Dziękuję.

Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na dodatkowe pytanie.

Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Matusiak. Mam pytanie do pana ministra odnośnie do sytuacji, która panuje na rynku węgla detalicznego.

Ja wiem, że, powiedzmy, zamieszanie, które wprowadziła Unia Europejska, dotyczące tzw. zielonej energii dzisiaj skutkuje tym, że właściwie jedyny opał, który jest wykorzystywany, który jest stabilny, to węgiel, którego obecnie brakuje na rynku. Panie Ministrze! Chciałem zadać pytanie: Jakie działania w tej sprawie zamierza podjąć rząd? Rozumiem, że teraz oczekujemy odpowiedzi od sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana Macieja Małeckiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Aktualne zapotrzebowanie na węgiel opałowy na rynku komunalno-bytowym w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 9 mln t rocznie. To zależy od warunków atmosferycznych, jakie panują w Polsce, bo te warunki mają bezpośrednie przełożenie na długość sezonu grzewczego i wielkość zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynków.

Dlatego nie da się w prosty sposób, np. przekierowując węgiel z innego sektora na ogrzewanie, zwiększyć ilości paliwa przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Ostatnia zima była zdecydowanie chłodniejsza, trwała dłużej.

Jak pokazują poprzednie lata, ta krzywa zakupów spada w miesiącach bezpośrednio przedzimowych.

Mówimy więc o sytuacji rynkowej, która zdarza się raz na kilkanaście lat. Wspomniałem, że banki i inne instytucje finansowe nie chcą finansować takich inwestycji, bo to wynika z ich polityki antywęglowej.

Wynika to z faktu, że tak jak wspomniałem, te ceny podlegają dynamicznym zmianom i może to się zmieniać w niedługim czasie. Mamy świadomość, że węgiel to paliwo wykorzystywane przez osoby, które są gorzej sytuowane, lub tam, gdzie nie ma jeszcze sieci gazowniczej. W Polsce jest ok. 10 tys. składów.

Np. w Polskiej Grupie Górniczej obowiązują ograniczenia w postaci sprzedaży do 3 t za gotówkę na wagach. W sklepie internetowym można kupić maksymalnie 5 t. Ograniczenia te nie dotyczą autoryzowanych sprzedawców, z którymi spółka ma podpisane wieloletnie umowy, dlatego można usłyszeć głosy, że z kopalni wyjeżdżają duże auta ciężarowe do 24 t, które są w pełni załadowane.

Sprzedaż, jak powiedziałem, jest dostosowana do rynku po to, żeby nie była powodem spekulacji, że ktoś spoza autoryzowanych dostawców wykupi większą część węgla w szczycie zapotrzebowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Panie Ministrze! Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Obserwując średnie ceny sprzedaży węgli opałowych w spółkach Skarbu Państwa, widać bardzo mocny trend sezonowy. Najniższe ceny pojawiają się w miesiącach luty-maj, natomiast najwyższe w okresie wrzesień-listopad.

Także informacje, które otrzymujemy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pokazują, że tam, gdzie mowa o podwyżkach z 900 zł do 1300 zł, to są działania sprzedawców detalicznych niezwiązanych ze spółkami Skarbu Państwa. Niektórzy sprzedawcy chcą wykorzystać ten run na rynku. Podam przykładowe ceny produktów spółek Skarbu Państwa, to jest cena brutto z podatkiem akcyzowym.

Trzeba też bardzo mocno powiedzieć, że w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze spekulacją na rynku gazu, widzimy już pierwsze, może nie pierwsze, kolejne, ale pierwsze tak bardzo widoczne, efekty czasem oderwanej od życia polityki klimatycznej Unii Europejskiej - tym właśnie skutkują dla odbiorców indywidualnych, ale też tym skutkują dla przemysłu. Takimi informacjami, tym przekazem też stale dzielimy się na arenie międzynarodowej, przekazujemy to naszym partnerom na forum Unii Europejskiej, po to żeby transformacja energetyczna Unii Europejskiej, transformacja pana Timmermansa i innych zwolenników tego radykalnego trendu, nie była prowadzona w oderwaniu od rzeczywistości, w oderwaniu od konkurencyjności gospodarki, w oderwaniu od dbałości o portfele rodzin.

Bardzo proszę, pan poseł Waldy Dzikowski jako pierwszy. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Nie będę przytaczał tutaj szczegółów technicznych ani zawiłości prawnych, bo to zostało opisane w naszym pytaniu. Będę mówił o ludziach.

Tu jest rola państwa, aby ochraniało ich i było strażnikiem ich bezpieczeństwa, w tym przypadku bezpieczeństwa energetycznego.

Najważniejsze jest to, żeby ludzie byli w państwie polskim traktowani dokładnie tak samo. Taka jest rola państwa polskiego. Każdy nasz rodak jest najważniejszy.

Bo polityka jest uprawiana w imieniu i dla ludzi. Wysoka Izbo! W tym wystąpieniu, mam nadzieję, podyktowanym troską, ale dosyć zaczepnym wobec rządu, pan poseł właśnie zmasakrował 30-letnią politykę prowadzoną przez liberałów w Polsce, szczególnie prowadzoną przez środowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Platformy Obywatelskiej. Bowiem państwo przez wszystkie lata od transformacji gospodarczej, transformacji politycznej opowiadaliście, że niewidzialna ręka rynku zrobi swoje, że nie jest ważne, kto jest właścicielem firm, że trzeba prywatyzować, wyprzedawać i państwo powinno się pozbywać różnych aktywów. Panie pośle, czy sieci gazowe w Opalenicy, w Tarnowie Podgórnym, w tych rejonach, zostały sprzedane przez samorządy?

Panie pośle, ma znaczenie, ma znaczenie.

Rząd nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób dana spółka prowadzi kontraktację gazu, w jaki sposób zabezpiecza się poprzez politykę zakupową, a tak naprawdę zabezpiecza swoich klientów przed zwyżkami cen gazu w dającej się przewidzieć perspektywie.

Z czego to wynika? Wynika to z tego, że gazociągi prowadzące z Rosji do Europy Zachodniej nie były wykorzystywane do wypełnienia magazynów gazu po bardzo mroźnej zimie. Mówiąc najprościej, Władimir Putin i Gazprom nie uzupełnili zapasów gazu po mroźnej zimie i dzisiaj mamy mniejszą podaż gazu w Europie.

Teraz widać, jak dalekowzroczna była polityka śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który po kolejnym szantażu gazowym Rosji uruchomił budowę terminala gazowego w Świnoujściu. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości finalizuje budowę gazociągu Baltic Pipe.

Jeszcze raz podkreślę, że rząd w żaden sposób nie miał wpływu na kontrakty zawierane przez spółkę, która nie jest w żaden sposób powiązana ze Skarbem Państwa, spółkę G.EN. i nie ma wpływu na warunki, w jakich ta spółka, jeszcze raz powtarzam, i z jakim wyprzedzeniem, kupuje gaz na kolejne okresy sprzedaży klientom, w jakich wolumenach i za jakie ceny.

Podkreślam, że rząd Polski podejmuje na arenie europejskiej działania zmierzające do tego, żeby właściwe organy unijne podjęły skoordynowane działania pozwalające zapobiec manipulacjom i niebezpiecznemu dla wszystkich uprzywilejowaniu gazociągu Nord Stream 2.

Niezależnie od tego, czy mówimy o gazie zaazotowanym, czy o gazie metanowym.

Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo!

Naprawdę mieszkańcy moich gmin, Kazimierza, Opalenicy, powiatu nowotomyskiego czekali na konkretne informacje.

A przecież nasz gaz, z naszych źródeł, nie musi być tak drogi jak ten gaz, o którym pan mówił, czyli gaz dostarczany z Gazpromu. My, panie ministrze, o to apelujemy, bo dysproporcje są zbyt duże. Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z zadowoleniem przyjmuję stanowisko posłów Platformy Obywatelskiej, którzy przyznają, że dotychczasowa polityka w postaci wmawiania Polakom, że niewidzialna ręka rynku zrobi swoje. i że wolny rynek rozwiąże wszelkie problemy, jest błędna. Państwo dzisiaj do tego się przyznaliście.

Ten projekt jest procedowany w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Chodzi o to, że projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada możliwość rozłożenia w czasie tego skokowego wzrostu cen gazu dla gospodarstw domowych. a wczoraj na posiedzeniu komisji nie poparliście tego projektu, nie poparliście rozwiązań korzystnych dla polskich odbiorców gazu.

W związku z tym podkreślam, że zaproponowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja Prawa energetycznego zakłada możliwość złagodzenia nagłego, skokowego wzrostu cen zakupu gazu poprzez przeniesienie wzrostu cen przez sprzedawcę w trakcie obowiązywania taryfy na kolejne okresy taryfowe.

I jednocześnie liczę, że ta sytuacja będzie taką okazją do refleksji, że nie wszystko można sprywatyzować, że nie wszystko można sprzedawać, tak jak były wyprzedawane sieci gazociągów, sieci ciepłownicze.

Dziękuję, panie ministrze.

Bardzo proszę, jako pierwsza pyta pani poseł Anita Czerwińska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo.

Pani Poseł! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście pojawiają się już informacje w przestrzeni medialnej na temat zamierzeń ministerstwa i całego rządu odnośnie do wynagrodzeń nauczycieli. Generalnie wychodzimy z założenia, że obecne wynagrodzenia są zbyt niskie i powinny ulec podwyższeniu. Co prawda w ostatnich kilku latach rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli łącznie o ok. 30%, ale nadal uważamy, że te wynagrodzenia powinny być wyższe. Jest to zawód szczególny, zawód, który decyduje o tym, jak będą wyglądały kolejne pokolenia Polaków, jak będzie wyglądała Polska za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Dlatego też zaproponowaliśmy w ramach dialogu ze związkami zawodowymi i samorządami propozycje wzrostu wynagrodzeń od września 2022 r. Ten wzrost wynagrodzeń będzie jednocześnie związany ze zmianą tzw. pragmatyki zawodowej, czyli m.in. zmianą w zakresie czasu pracy nauczycieli przy tablicy, redukcji obowiązków biurokratycznych, tak aby zbilansować te zmiany czasu pracy przy tablicy, także awansu zawodowego - jego uproszczenie, odbiurokratyzowanie - plus wprowadzenie nowej kategorii tzw. czasu dostępności nauczyciela, tak aby nauczyciel był dostępny w większym stopniu dla rodziców i uczniów. Te planowane wzrosty wynagrodzeń mają doprowadzić do tego, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o ok. 1 tys. zł na każdym stopniu awansu zawodowego. Jeśli chodzi natomiast o wynagrodzenie przeciętne, ten wzrost może sięgać nawet 1400 zł.

Mieliśmy wiele sygnałów - i my tak samo uważamy - że jest to stawka niezadowalająca i powinna zdecydowanie wzrosnąć. Po podwyżce, którą proponujemy, ta stawka będzie wynosiła 4010 zł. Najczęściej występujący stopień awansu zawodowego nauczyciela to nauczyciel dyplomowany, to mniej więcej 2/3 wszystkich nauczycieli pracujących w polskich szkołach. Dziś stawka wynagrodzenia zasadniczego takiego nauczyciela wynosi 4046 zł. Po podwyżce od września 2020 r. jego stawka ma, według naszej propozycji, wynosić 5130 zł. Przy czym mówię tylko i wyłącznie o wynagrodzeniu zasadniczym, a wynagrodzenie nauczyciela składa się także z kilku innych elementów, m.in. dodatku stażowego. W przypadku nauczycieli z 20-letnim i dłuższym czasem pracy, a to odnosi się najczęściej do nauczycieli dyplomowanych, ten dodatek będzie już wynosił 20%. Są także godziny ponadwymiarowe, dodatki funkcyjne, trzynastka i wiele innych elementów, podobnie jak z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Widać, że tu jest wyraźny wzrost o ponad 1400 zł. W przypadku nauczycieli dyplomowanych, tych najczęściej pracujących w naszej szkole, stawka obecnie obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia to 6510 zł.

Widać więc, że jest to wyraźnie różniąca się stawka zarówno wynagrodzenia zasadniczego, jak i wynagrodzenia przeciętnego.

Informacja o tym, że nauczyciel pracuje podobno tylko 18 godzin, jest nieprawdziwa. On przecież dodatkowo przygotowuje się do zajęć, sprawdza klasówki, przygotowuje te sprawdziany, spotyka się z rodzicami, ma konsultacje dla uczniów, jeździ na wycieczki, uczestniczy w radach pedagogicznych itd. Możemy więc porównać także to wynagrodzenie w 40-godzinnym czasie pracy.

Widać więc wyraźnie, że ministerstwo działało we współpracy z innymi resortami, bo potrzebna była tu decyzja pana premiera, Ministerstwa Finansów, potrzebne były dodatkowe środki w budżecie państwa, aby takie wynagrodzenia podnieść. Łączny koszt wzrostu wynagrodzeń, który planujemy, to jest ok. 8 mld zł - tyle dodatkowo w ciągu roku musi się pojawić w budżecie, aby te podwyżki można było zrealizować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, rezygnuję z pytania. Dziękuję bardzo.

Pierwsze pytanie zadają państwo posłowie Iwona Śledzińska-Katarasińska i Dariusz Joński. W lipcu br. wiceminister Jarosław Sellin, odpowiadając na moje i pani marszałek Kidawy-Błońskiej pytanie o funkcjonowanie tzw. fundacji patriotycznej, odpowiedział, cytuję: Otrzymane granty przeznaczone zostaną na różnorodne projekty promujące historię i dziedzictwo narodowe naszej ojczyzny oraz inicjatywy promujące postawy patriotyczne i obywatelskie. To były zapowiedzi, a wygląda to m.in. tak: prawie 4 mln zł otrzymały objęte protektoratem wicepremiera Glińskiego powiązane ze sobą organizacje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Straż Narodowa oraz Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości. Pytam wobec tego: Jaką historię i dziedzictwo narodowe promowały bojówki Roberta Bąkiewicza, lidera tych trzech skrajnie nacjonalistycznych organizacji, zakłócając śpiewanie hymnu państwowego przez dziesiątki tysięcy osób zgromadzonych na placu Zamkowym? Jakie postawy patriotyczne popchnęły członków tych bojówek do zakłócania wystąpienia pani Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki, bohaterki powstania warszawskiego? Wstyd i hańba, panowie ministrowie, wstyd i hańba, rządzie PiS. Mam takie pytanie: Czy już wystąpiliście, drogi rządzie, o zwrot tych pieniędzy i czy już je uzyskaliście z powrotem? Dziękuję. Wysoka Izbo! Pytam konkretnie o sprawę dofinansowań z Funduszu Patriotycznego dla dwóch Stowarzyszeń: Straż Narodowa i Marsz Niepodległości. Regulamin mówi wprost, że ocena dwóch ekspertów jest wiążąca. Mamy karty ocen, z których wynika, że jedno i drugie stowarzyszenie ocenione przez dwóch ekspertów w jednym i w drugim przypadku dostało po 184 punkty. Natomiast na stronie internetowej nagle okazuje się, że dostają 204 punkty i tym samym zostali zakwalifikowani do dofinansowania. Mam konkretne pytanie do pana ministra: Kto zmienił punktację, tak aby te dwa stowarzyszenia powiązane z panem Bąkiewiczem dostały pieniądze, i kiedy konkretnie zwrócą te pieniądze? Bardzo proszę, panie ministrze. Panie i Panowie Posłowie! Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Śledzińskiej-Katarasińskiej, to trudno mi na nie odpowiedzieć, bo nie ma czegoś takiego jak fundacja patriotyczna. ale domyślam się, że to było przejęzyczenie. Bardziej prawidłową nazwę przedstawił pan poseł Joński, mówiąc o programie Fundusz Patriotyczny. Jeśli chodzi o ten program, to jest to program własny. Tak, tak, właśnie domyśliłem się, pani poseł. Jeśli chodzi o ten program, to jest to program własny Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Chrześcijańsko-Demokratycznej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Takich programów grantowych mamy w ministerstwie i w podległych nam instytucjach ponad 30. W sumie w ciągu roku na ogół ok. 4 tys. podmiotów otrzymuje różnego rodzaju granty. Jak państwo się zainteresowali, z tych 4 tys. grantów przyznanych w ciągu roku dwoma grantami, ale nawet w tym programie, który tak szczególnie państwa zainteresował, czyli Fundusz Patriotyczny, chcę poinformować, że wniosków było 2 tys., a beneficjentów ostatecznie 150, oczywiście w ramach tych punktacji, które tam zgodnie z regulaminem były dokonywane. Od razu odpowiadam też na wątpliwość pana posła Jońskiego, że regulamin mówi, że rzeczywiście punktacji dokonuje dwóch ekspertów. Ale ten sam regulamin mówi o tym, że potem te punktacje oceniane są przez panel ekspertów, czyli szersze grono. A ostateczną decyzję co do punktacji i dotowania dokonuje dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Chrześcijańsko-Demokratycznej. A więc przyszło 2 tys. wniosków na ponad 550 mln zł.

Ten program, ta pierwsza edycja grantowa Funduszu Patriotycznego ma taką nazwę „Wolność po polsku” Państwo interesujecie się już od dłuższego czasu zresztą w przestrzeni medialnej tylko dwoma z tych 150 podmiotów, które te granty otrzymały.

Powtarzam: tylko pierwszą stronę.

Państwo interesujecie się tymi dwoma: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Stowarzyszenie Straż Narodowa, które otrzymały zgodnie z punktacją też taką dotację. Pani raczyła nazwać z trybuny sejmowej te organizacje bojówkami. To nie jest mój problem. To jest problem relacji między panią a tymi stowarzyszeniami. One być może się przysłuchują. Przysłuchują się tej debacie i nie wiem, jaka będzie reakcja. Ale ma pani prawo w ramach wolności słowa oczywiście takiego określenia użyć. Nie 4 mln w sumie na te stowarzyszenia przeznaczono, tylko 3 mln w ramach podziału tych środków, więc każde legalnie działające stowarzyszenie w Polsce w ramach szeroko pojętego ruchu NGO-sów ma prawo występować w państwie polskim zarówno do budżetu rządowego, jak i do budżetu samorządowego, różnych organów władzy samorządowej o granty i zgodnie z różnymi procedurami, regulaminami, programami, które są dedykowane poszczególnym programom grantowym, ma prawo takie granty otrzymywać. Z tego, co wiem, te stowarzyszenia, które są przedmiotem szczególnego państwa zainteresowania, są organizacjami legalnie działającymi w Polsce. Dziękuję. Teraz dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Michał Szczerba. Szanowni Państwo! Czy rządowi PiS nie jest głupio, że środków nie otrzymało Muzeum Powstania Warszawskiego na cele bezpieki, Fundacja Ośrodka KARTA czy też, panie marszałku, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie? Jak to jest możliwe, że po pół roku po zarejestrowaniu stowarzyszenia zwykłego z ułomną osobowością prawną Stowarzyszenie Straż Narodowa otrzymuje 1 mln 700 na zakup siedziby, mimo że Fundusz Patriotyczny nawet nie ma własnej siedziby i siedzi kątem w PKP? Szanowni Państwo! Z panem posłem Jońskim pokazaliśmy, że działaliście poza regulaminowo, że dwóch ekspertów oceniło wnioski na 184, a w punktacji, którą pokazaliście światu, było 204. Jak te 20 punktów zostało dodane? Ani panel ekspertów, ani dyrektor nie mają prawa zmieniać punktacji. Pan się do tego kompletnie nie odniósł. Ani poseł Joński, ani posłanka Śledzińska-Katarasińska, ani ja nie damy się zastraszyć w tej sprawie. Będziemy tę sprawę drążyć. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. To, że pan poseł nie da się zastraszyć, to ja wiem, bo pan słynie z odwagi i na trybunie sejmowej, i na różnych eventach pozaparlamentarnych. Skoro ja mam prawie 3 minuty na odpowiedź i skoro padły tutaj zarzuty, że ktoś nie otrzymał dofinansowania w ramach Funduszu Patriotycznego, to przypomnę jeszcze raz, że wniosków było 2 tys., a środki mogło otrzymać 150 podmiotów. Wnioski były na 550 mln, a do podziału było 30 mln.

A więc ja jeszcze sobie ten czas wykorzystam i przedstawię instytucje, które otrzymały. Fundacja Pokolenia Kolumbów, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Fundacja Humble 90, Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Na Skałce, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Archidiecezja Lubelska, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Drozdowie, Towarzystwo Salezjańskie, Fundacja Służba Niepodległej, Opatowski Ośrodek Kultury, Fundacja Obowiązek Polski, Fundacja Dobrej Rady, Fundacja Dziedzictwo Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, Fundacja na Rzecz Szpitala Ubogich im. Świętej Jadwigi Królowej w Bieczu, Fundacja świętego Benedykta, Fundacja Advocata Nostra, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego, Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji i Sztuki, Strzelcy Rzeczypospolitej. Fundacja Action-Life, Fundacja Projekt Patriotyzm, Stowarzyszenie Pro Artis, Fundacja edukacyjno-patriotyczna „Dumni z Polski” Stowarzyszenie Scena Kultury, Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Fundacja Rozwoju Kultury we Wrocławiu, Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki, Stowarzyszenie Sąsiedzi 05–123, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej, Fundacja Instytut Poznański, Fundacja Wspierania Myśli Polskiej, Fundacja Społeczno-Kulturalna Sarmatia. Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski, Fundacja Między Słowami, Koło Gospodyń Wiejskich Różanka w Kaniewie, Stowarzyszenie Bonum Publicum, Fundacja Obserwatorium Społeczne, Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, Fundacja Misji Obywatelskiej, Fundacja Tradycji Miast i Wsi, Fundacja Klubu Ronina, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Wielkopolscy Patrioci, Mrągowskie Centrum Kultury, Fundacja Rodziny Witaszków. Dziękuję, panie ministrze. Posłowie Krzysztof Gawkowski, Magdalena Biejat i Katarzyna Kotula wraz z grupą posłów pytają o działania rządu na rzecz zapobiegania wzrostowi ubóstwa. Bardzo proszę, jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Katarzyna Kotula. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę o udzielenie bieżącej informacji na temat prognoz i analiz realizowanych czy też zrealizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów w zakresie efektów, jakie Polski Ład wywrze na jakość i dostępność usług publicznych, i co za tym idzie - w zakresie tego, jak wpłynie on na strukturę wydatków gospodarstw domowych. Czy ministerstwo ma informacje, wykonało analizy i sporządziło prognozy dotyczące tego, w jakim stopniu spadki dochodów samorządów terytorialnych przełożą się na dostępność i jakość usług publicznych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, transportu, usług opiekuńczych, opieki społecznej, wsparcia osób najbiedniejszych, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów? Czy ministerstwo zamierza sporządzić prognozy dotyczące tego, w jaki sposób zmiany dostępności usług publicznych wpłyną na budżety gospodarstw domowych, w szczególności w rodzinach z dziećmi, rodzinach wielodzietnych oraz rodzinach osób z niepełnosprawnościami?

Obniżenie podatku dochodowego, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu progresji podatkowej do 120 tys. zł są sztandarowymi elementami Polskiego Ładu. Jest to świetna zmiana, Lewica upominała się o nią od ponad dekady, ale każde rozwiązanie, nawet najlepsze i najbardziej potrzebne, da się niestety zepsuć albo spartaczyć, czasem być może niechcący, a czasem całkiem świadomie. Mam coraz większa obawę, graniczącą z przekonaniem, że właśnie z tym mamy tutaj do czynienia. Na zmianach podatkowych ma skorzystać 18 mln obywateli, w których kieszeniach zostanie łącznie ok. 9 mld zł. Problem w tym, że jednocześnie w gminach i powiatach ubędzie ponad 14 mld rocznie, a to oznacza 14 mld mniej na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni zdrowia, komunikacji miejskiej, na remonty budynków i dróg, domy kultury i politykę socjalną. Rząd, pozostawiając te 9 mld w kieszeni obywateli, jednocześnie wycina w niej pokaźną dziurę. Środki zaoszczędzone na niższym PIT szybko rozejdą się na usługi, które przestaną być publiczne.

Bardzo proszę, pani minister. Szanowny Panie Marszałku! Państwo Posłowie! Odpowiadam na pytanie w sprawie działań rządu na rzecz zapobiegania wzrostowi ubóstwa, w tym wśród osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w kontekście raportu Poverty Watch i zmian w budżecie na 2022 r. Jak słyszałam, pani poseł poszerzyła zakres tematyczny pytania, zatem dalszą część, o którą pani dopytała, przedstawimy na piśmie. Przede wszystkim, szanowni państwo, z dużą ostrożnością należy interpretować dane dotyczące wzrostu ubóstwa skrajnego, ponieważ nie jest on związany ze spadkiem dochodów gospodarstw domowych, ale z ograniczonymi w przypadku niektórych grup, a mówimy tutaj o osobach z niepełnosprawnościami, możliwościami wydatkowymi. Przyczyn wzrostu ubóstwa skrajnego upatrywać można w zmianach dotyczących konsumpcji, związanych ze zmniejszeniem się wydatków gospodarstw domowych wynikającym z ograniczeń spowodowanych pandemią i lockdownem. Należy również podkreślić, że sukcesywnie spada liczba gospodarstw domowych, którym udzielona została pomoc społeczna z powodu ubóstwa. W 2020 r. takich gospodarstw było o 33 tys., a więc o 8 punktów procentowych, mniej niż w roku 2019. Są kierowane m.in. do osób z niepełnosprawnościami, ale także, co ważne, do ich rodzin.

Pozwolicie państwo, że podam kilka danych liczbowych. Programy rządowe i resortowe w tym zakresie realizowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który również realizują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Tutaj kwota dofinansowania to 250 mln zł. Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który w zakresie finansowania zadań związanych z ich utworzeniem, ale także z kontynuacją działań.

Oczywiście mamy program dotyczący rodzinnych ośrodków wsparcia - 15 mln zł.

Dodatkowo przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój” uruchomione zostały projekty mające na celu włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Włączenie wyłączonych” oraz projekt dotyczący opracowania projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Do działań rządu na rzecz przeciwdziałania ubóstwu należy również zaliczyć silną pomoc społeczną, a więc szeroko pojętą politykę pomocy społecznej państwa, której celem jest oczywiście umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne usprawnienia, ograniczone zasoby i możliwości.

Jest to spadek o blisko 18% w stosunku do roku 2018.

Do najważniejszych działań, które wpisują się w walkę z ubóstwem, w przeciwdziałanie ubóstwu, należy przede wszystkim wspieranie jednostek samorządu terytorialnego.

Mam nadzieję, że ta odpowiedź wyczerpuje wątpliwości państwa posłów. Jeśli coś wymaga doprecyzowania, oczywiście biuro pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami prześle resztę odpowiedzi na piśmie. Pani poseł Magdalena Biejat zada dodatkowe pytanie.

Teraz słychać. Mam pytanie doprecyzowujące. Powiedzmy jasno: drożyzna, inflacja, spadek dochodów w pandemii już dawno pochłaniają dużą część programów i bezpośrednich transferów, które państwo wprowadzają, takich jak 500+, którym państwo lubią się chwalić. Problemem tego programu, tak samo zresztą jak bardzo wielu programów, które państwo wprowadzają, jest to, że po prostu są to programy doraźne, które zajmują się tylko częścią problemu. Nie ma natomiast systemowych rozwiązań. Zamiast poprawy jakości życia, wzrostu płac, wyrównania płac kobiet i mężczyzn, dobrych usług publicznych są pieniądze do ręki co miesiąc i słowa: radź sobie sam. Efekt jest taki, że ewidentnie widać, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jednak gdzieś pokutuje cały czas duch prof. Balcerowicza, ponieważ macie podejście opierające się na tym, że trzeba dać przede wszystkim pieniądze i niech ludzie radzą sobie sami. Naprawdę prosiłabym o ustosunkowanie się do pytania pani posłanki Kotuli i mojego, które powtórzę. Panie marszałku, jeśli tylko mogę dosłownie w 15 sekund odnieść się do kwestii osób z niepełnosprawnościami, bo pani minister również miała możliwość dokończenia swojej myśli. Pani mówiła dużo o osobach z niepełnosprawnościami, tymczasem nadal nie jest wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego wyrównujący świadczenia dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. Nie ma nadal dostępnej asystencji osobistej, mimo że ciągle się chwalicie, że są na to pieniądze, a pieniądze w budżecie na 2020 r. na zasiłki, na dożywianie zostały obniżone, a generalnie budżet na pomoc społeczną w 2020 r. ulega raczej stagnacji lub lekkiemu obniżeniu, co w kontekście 6-procentowej inflacji jest de facto obniżeniem nakładów na pomoc społeczną.

Pani minister, bardzo proszę. Szanowna Pani Poseł!

Po drugie, wydawało mi się, że odpowiedziałam na pani wątpliwości, bo kwoty, które przeznaczamy na programy wspierania osób z niepełnosprawnościami, uruchamianie asystencji osobistej, centrów opiekuńczo-mieszkalnych, które mają wspierać osoby z umiarkowanym i lżejszym stopniem niepełnosprawności, które są w stanie funkcjonować poza jakimś, powiedzmy, zamkniętym ośrodkiem, tylko w mieszkaniu chronionym z funkcją asystenta i samodzielnie wchodzić w wykonywanie codziennych funkcji, funkcji życiowych, ograniczanych właśnie niepełnosprawnością, ewidentnie dowodzą tego, że wszystkie działania rządu i miliardy złotych, a ja tutaj przytoczyłam kilkanaście różnych wskaźników, w tym również wskaźników kwotowych, ewidentnie wskazują na to, że polityka rządu, w ramach której mieści się w tej kadencji, przypominam, pani poseł, przygotowanie w ramach spełnienia warunku podstawowego Unii i Komisji Europejskiej.

Jeśli to pani poseł nie satysfakcjonuje, to na dalszą część pytań odpowiemy na piśmie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego pytania. Posłowie Mieczysław Kasprzak i Jarosław Rzepa z Koalicji Polskiej pytają o likwidację wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych. Pierwszy pytanie zadaje pan poseł Jarosław Rzepa. Panie Marszałku! W ostatnich dniach społeczności powiatów pyrzyckiego i polickiego zmroziły informacje o pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie zamiaru likwidacji wydziałów zamiejscowych w Pyrzycach Sądu Rejonowego w Stargardzie i wydziałów zamiejscowych w Policach Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. W obu tych miastach powiatowych, które zamieszkuje ponad 100 tys. mieszkańców, funkcjonują obecnie wydziały karne i ksiąg wieczystych. Pani Minister! Przeniesienie spraw z Polic i Pyrzyc do Szczecina i Stargardu zmniejszy szybkość postępowań karnych i ksiąg wieczystych głównie z powodu oddalenia siedziby sądu od miejscowości w powiatach polickim i pyrzyckim. Dziś jest to zaledwie najwyżej kilkanaście kilometrów, a jutro może być to kilkadziesiąt. Bardzo utrudnione, a czasem nawet wykluczone, będą dojazd i obecność w sądzie ze względu na brak funkcjonujących połączeń środkami komunikacji publicznej. Głównie dotyczyć to będzie miejscowości wiejskich powiatu pyrzyckiego, które nie mają regularnego połączenia ze Stargardem. To samo dotyczyć również będzie miejscowości wiejskich gmin Dobra, Nowe Warpno czy Kołbaskowo w powiecie polickim. Niewątpliwie wzrosną koszty i wydatki ponoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niezwykle ważne, pani minister, powinno być to, żeby prokuratorzy zajmowali się swoimi zadaniami, funkcjonariusze Policji strzegli bezpieczeństwa obywateli, a nie poświęcali swój czas pracy na zbędne podróże do sądu oddalonego nie o kilka, ale o kilkadziesiąt kilometrów. Wreszcie pragnę wspomnieć o skutkach społecznych pani zapowiedzi. Pamiętać należy o osobach pokrzywdzonych, interesantach ksiąg wieczystych, osobach starszych, dla których wyprawa z ich miejscowości zamieszkania do Pyrzyc i Polic jest już dzisiaj sporym utrudnieniem i wyzwaniem. To jest, pani minister, fizycznie niemożliwe, nawet ze względu na sposób przydzielania spraw. Również sytuacja pracowników tych sądów może doprowadzić do ich indywidualnych decyzji o zakończeniu pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pani Katarzyna Frydrych. Wysoka Izbo! Wydaje mi się, że pytanie jest już bezprzedmiotowe. Pytanie brzmi: Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zlikwidować wydziały zamiejscowe sądów rejonowych? Są to wydziały zamiejscowe w Pyrzycach i w Policach. Decyzja w zakresie zaprzestania kontynuowania prac związanych ze zniesieniem tych wydziałów zamiejscowych została podjęta wcześniej, przed skierowaniem pytania. A zatem odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi, że aktualnie nie jest planowane zniesienie wydziałów zamiejscowych w tych sądach. Chciałabym tylko zaznaczyć - pan poseł zresztą już o tym mówił - że są to wydziały zamiejscowe, wydziały karne i wydziały ksiąg wieczystych. Historycznie rzecz ujmując, wydziały zamiejscowe w Policach funkcjonują na bazie poprzedniego sądu grodzkiego od 2001 r., natomiast wydziały zamiejscowe w Pyrzycach od 1 stycznia 2013 r. Jeśli chodzi o sytuację wydziałów zamiejscowych w Pyrzycach, to decyzja o utworzeniu tych wydziałów była podyktowana tylko i wyłącznie sytuacją lokalową w sądzie. W chwili obecnej sąd ma dobre, bardzo dobre warunki lokalowe i teoretycznie można byłoby dokonać przeniesienia tych wydziałów do sądu. Poruszona została również kwestia odległości pomiędzy Policami a sądem w Szczecinie i Pyrzycami a sądem w Stargardzie. Jeśli chodzi o Police, to odległość do siedziby wynosi 17 km, a z Pyrzyc do Stargardu 27,7 km. Ministerstwo Sprawiedliwości dokonuje zawsze dokładnej analizy, zanim podejmie decyzję w zakresie zniesienia jakiegokolwiek wydziału zamiejscowego. Kierujemy się dobrem obywateli, zapewnieniem im dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Bierzemy pod uwagę również okoliczności związane z obciążeniem orzeczników, bo to obciążenie tak naprawdę daje gwarancję szybkiego, sprawnego rozpoznania sprawy. Bierzemy pod uwagę wpływ, liczbę etatów, faktyczną obsadę w danej jednostce. I tak jak mówiłam, w chwili obecnej prace nie są kontynuowane, one zostały zaprzestane, zanim zostało skierowane pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani minister, za tę deklarację, mieszkańcy na pewno odetchną z ulgą.

Bardzo proszę o odpowiedź. Jeszcze raz odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pani Katarzyna Frydrych. Tak naprawdę jeśli chodzi o wydziały ksiąg wieczystych, można kierować wnioski elektronicznie, można kierować wnioski na piśmie, kwestia tylko dostępu do wydziałów karnych. W chwili obecnej - trzeba wziąć pod uwagę zapowiedź ze strony pana ministra sprawiedliwości dotyczącą reformy sądownictwa - trwają prace dotyczące kwestii związanej z tzw. nową siatką sądów i na pewno okoliczność, o której pan poseł był uprzejmy w chwili obecnej wspomnieć, o którą zapytał, będzie również przedmiotem dogłębnej analizy. Tak jak mówię, zawsze minister sprawiedliwości ma na względzie dobro obywateli i zapewnienie im dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani minister. Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Jarosław Gonciarz, Wojciech Szarama i Bożena Borys-Szopa z Prawa i Sprawiedliwości pytają w sprawie zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia i odwołania czasu letniego. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Jarosław Gonciarz. Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Pomysł odejścia od zmiany czasu pojawia się na forum krajowym oraz unijnym od kilku lat. W samym tylko Parlamencie Europejskim odbywały się na ten temat debaty i różnego rodzaju wysłuchania publiczne, zaś Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne w państwach członkowskich, zgodnie z którymi blisko 90% głosujących zadeklarowało chęć odejścia od zmian czasu. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu. Mając na względzie powracającą jak bumerang tematykę zmiany czasu oraz przesłanki, które wskazują na zaniechanie tej czynności w organizacji naszego życia, pragnę zapytać, czy ministerstwo pracuje nad przepisami, które zaprzestałyby nakazywać zmianę czasu z zimowego na letni i na odwrót. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani minister. Wysoka Izbo!

W związku z tym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą przygotować przepisy prawne wprowadzające w życie regulacje wynikające z powyższego komunikatu, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia i rozwiązania w tym zakresie. Polska od początku popierała podjęte przez Komisję Europejską w 2018 r. działania zmierzające do rewizji dyrektywy jako zgodne z oczekiwaniami społecznymi, ale jednocześnie, tak jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, zachęcała Komisję do przedstawienia kompleksowej analizy korzyści i skutków społeczno-ekonomicznych odstąpienia od dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu, która jednak do tej pory nie została przygotowana. Przedmiotowy problem jest wieloaspektowy, dotyczy wielu dziedzin życia, osobistego, społecznego, gospodarczego, oraz innych uwarunkowań w każdym z unijnych krajów, takich jak np. uwarunkowania geograficzne, kulturowe czy inne strefy czasowe. Polska, tak jak i inne kraje, uważa, że z ekonomicznego punktu widzenia najważniejsze jest zachowanie harmonizacji w kwestii czasu pomiędzy państwami członkowskimi, głównie ze względu na konieczność takiej harmonizacji na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Gdyby doszło do odejścia od zmian czasu i przejścia na jeden wybrany czas, wszystkie kraje członkowskie musiałyby mieć czas konieczny na wypracowanie stanowiska co do tego, jaki czas powinien obowiązywać w danym kraju w powiązaniu z tym, jaki czas będzie obowiązywał w krajach sąsiadujących w danym regionie Unii Europejskiej. Jednak na forum unijnym od końca 2019 r. nie były podejmowane działania w zakresie wypracowania ostatecznego kształtu dyrektywy znoszącej sezonowe zmiany czasu, co wiązałoby się również z intensyfikowaniem prac zmierzających do wypracowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zharmonizowanego stanowiska co do obowiązującego czasu. Obecnie, m.in. również w związku z trwającą pandemią, nie są podejmowane prace w tym zakresie na forum Unii Europejskiej. Tym samym na chwilę obecną nie jest wiadome, jakie będą dalsze losy tego projektu i czy ostatecznie odejdziemy od sezonowych zmian czasu. Kolejne pytanie również pan. Japończycy wyliczyli, że stosowanie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. t i pomóc zaoszczędzić do 930 mln l paliwa.

Dziękuję. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pani Olga Ewa Semeniuk. Bardzo proszę, pani minister. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle!

Bardzo dziękuję. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Elżbieta Duda i Mariusz Trepka z Prawa i Sprawiedliwości zadadzą pytanie w sprawie mobilnych aplikacji dla osób poszukujących pracy. Jako pierwsza zadaje pytanie pani poseł Lidia Burzyńska. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat wprowadza instrumenty mające na celu rzecz bardzo ważną dla społeczeństwa, mianowicie niwelowanie stopy bezrobocia. Sukcesywne podnoszenie płacy minimalnej, realizowanie programów społecznych i aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i wykluczonych przynoszą wymierne skutki w postaci spadku bezrobocia.

Od marca br. poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce systematycznie spadał. Według wstępnych danych na koniec września 2021 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 936 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu ze stanem z końca sierpnia br. liczba ta zmniejszyła się o prawie 25 tys. osób, czyli o ponad 2,5%. To oznacza, że tempo spadku było niemal dwukrotnie większe niż miesiąc wcześniej. Szanowny Panie Ministrze! Jak dane dotyczące rejestrowanego bezrobocia przedstawiały się w poszczególnych województwach, ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego? Dziękuję bardzo. Na to pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pan Stanisław Szwed. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za te pytania. To bardzo ważny temat, związany z sytuacją na rynku pracy.

A jeżelibyśmy to rozłożyli w perspektywie rocznej, to jest to spadek o 10% w stosunku do poprzedniego okresu 10-miesięcznego.

Czyli w skali całego kraju mamy najniższą stopę bezrobocia w województwie wielkopolskim, a drugie województwo to województwo śląskie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoki Sejmie! Dziękuję bardzo panu ministrowi za udzielenie wyczerpującej informacji na temat działań podjętych przez rząd w zakresie ochrony miejsc pracy, szczególnie w sytuacji pandemii, która nas dotknęła. Chciałabym zapytać, panie ministrze, o bezpłatną aplikację mobilną przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla osób poszukujących pracy. W jakim terminie możliwe jest wdrożenie tej aplikacji i na jakie efekty jest obliczone jej przygotowanie dla osób poszukujących pracy? Bardzo dziękuję. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Dziękuję, panie marszałku.

Czyli ta aplikacja w zdecydowany sposób pomoże pracodawcom w poszukiwaniu osób, które szukają pracy. I odwrotnie: dla pracowników, którzy potrzebują i szukają pracy, jest oferta wolnych miejsc pracy. 52% użytkowników korzysta z Centralnej Bazy Ofert Pracy na smartfonach, 45% na komputerach stacjonarnych, 3% na tabletach, to też się będzie zmieniać.

Wszystkie te działania, które podejmowaliśmy w ramach rządu, pozwalają nam, że jesteśmy w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o wdrażanie Polski cyfrowej, która jest niesłychanie istotna dla naszych mieszkańców i dla tego, co jest potrzebne w bieżącej działalności. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jako pierwsza zadaje pytanie pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek. Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Centra integracji społecznej działają od ponad 18 lat. Funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej m.in. osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 11 tys. osób. Nie wszyscy bezrobotni kwalifikowali się do możliwości objęciach ich pomocą przez CIS-y. Aktualnie przygotowywana jest nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Głównym celem tej nowelizacji jest dostosowanie jej przepisów do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych w kraju. Panie ministrze, moje pytanie brzmi: Jakie propozycje zmian w zakresie funkcjonowania centrów integracji społecznej przewiduje projekt nowelizacji ustawy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie.

Pamiętajmy, że rozmawiamy o zatrudnieniu socjalnym, o ekonomii społecznej, która dotyka osób, które najbardziej takiego wsparcia potrzebują.

Tak jak już powiedziałem, będzie okazja, żeby w czasie prac parlamentarnych jeszcze raz państwu o tym powiedzieć.

Temu przyświecają zmiany, jeśli chodzi o kwestie zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Warunkiem uczestnictwa w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a nawet korzystania z jednorazowego indywidualnego poradnictwa specjalistycznego w KIS jest realizacja kontraktu socjalnego zawartego w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Obowiązujące rozwiązanie jest często sporym utrudnieniem głównie dla organizacji pozarządowych prowadzących kluby integracji społecznej w małych miejscowościach lub gminach wiejskich, gdzie świadomość potrzeby podejmowania aktywnych form zapobiegania wykluczeniu społecznemu nie jest wystarczająco wysoka nawet wśród pracowników socjalnych. Panie Ministrze! Czy podstawą objęcia pomocą przez KIS mogłaby być bezpośrednia umowa reintegracyjna zawierana pomiędzy uczestnikiem a podmiotem prowadzącym klub integracji społecznej?

Dziękuję. Oczywiście w ramach ustawy chcemy też rozszerzyć katalog podmiotów uprawnionych do tworzenia centrów integracji społecznej. W zmianach w ustawie nie mamy takiego bezpośredniego przepisu, ale jesteśmy jeszcze ciągle w trakcie prac nad ustawą, tak że warto się jeszcze również zastanowić nad tymi propozycjami, o których pani poseł mówiła. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przystępujemy do następnego pytania.

Jako pierwszy zadaje pytanie pan poseł Sławomir Nitras. Panie Ministrze! Panie ministrze, zadajemy pytanie w imieniu zachodniopomorskiego i Szczecina. Szczecin to wyjątkowe miasto, bo położone najdalej od stolicy, od Warszawy - ponad 600 km. Pan zapewne wie, że dzisiaj pociągiem do Szczecina jedzie się 9 godzin.

Nie ma takiego województwa i niestety nawet w planach dotyczących centralnego portu lotniczego nie uwzględniliście Szczecina jako miasta, z którego można dojechać do tego portu. Chciałbym zapytać pana dzisiaj o dwa kluczowe projekty z punktu widzenia aglomeracji szczecińskiej. Szczecin jest miastem, przez który przechodzi droga krajowa nr 10. Na północy Szczecina są wielkie zakłady produkcyjne w Policach i cały transport przechodzi przez miasto. Żeby zorganizować transport w Szczecinie, potrzebujemy dwóch projektów.

Będą oddane te projekty, które są samorządowe, czyli będziemy mieli przystanki, będziemy mieli dojazdy do przystanków, ale nie będziemy mieli kolei, bo za to odpowiada państwowa już dzisiaj spółka, która po prostu nawaliła z przetargami.

Pan premier, pan Brudziński, pan minister Adamczyk obiecali nam, że w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na obejście zachodnie Szczecina. Bez tych dwóch projektów Szczecin sprowadzacie do XIX w. Mam nadzieję, że jest to odpowiedź: za rok, za dwa, za trzy, a nie za 12. Dziękuję. Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że ostatnie rozstrzygnięcia Polskiego Ładu dają temu największy wyraz. Ale także działania Ministerstwa Infrastruktury, które są podejmowane w ostatnich latach, są dowodem na to, że chcemy rozwijać komunikację nie tylko w samym Szczecinie czy przy Szczecinie, ale w ogóle w województwie zachodniopomorskim, ponieważ w naszej ocenie na dane miasto należy patrzeć z perspektywy całego regionu. Ośrodki takie jak Szczecin, Poznań, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra są ośrodkami, które są stolicami danych regionów i przez ten pryzmat należy patrzeć na całość, bo to daje taki kompleksowy obraz rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej. Szanowni Państwo!

Skoro Szczecin jest wykluczony komunikacyjnie - w mojej ocenie aż tak źle nie jest, a będzie jeszcze lepiej - to oznacza, że przez lata nie robiono nic, żeby ta sytuacja się zmieniła. Przypomnę, że przecież 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej to fakt. Jeżeli chodzi o zachodnią obwodnicę Szczecina, to potwierdzam następujący fakt: zachodnia obwodnica Szczecina została wpisana do rządowego „Programu budowy dróg krajowych”, który na najbliższą perspektywę będzie w ramach Polskiego Ładu realizowany. Kiedy te środki będą potrzebne do uruchomienia, zostaną uruchomione. W tej chwili szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie przygotowywania przetargu, który niebawem zostanie ogłoszony na zaprojektowanie, a później docelowo oczywiście zbudowanie zachodniej obwodnicy Szczecina. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Inną ważną inwestycją drogową, która usprawni komunikację Szczecina nie tylko z Warszawą, nie tylko z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ale w ogóle z centralną Polską, jest budowa drogi ekspresowej S10.

Jeżeli chodzi o kolejne odcinki w kierunku skrzyżowania z drogą ekspresową S11 i dalej w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy, Torunia, następnie w kierunku Warszawy, te odcinki są w trakcie przygotowywania. Pracujemy nad złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Zapewniam panów posłów, że środki finansowe na budowę drogi ekspresowej S10 na całym odcinku, i w województwie zachodniopomorskim, i w województwie kujawsko-pomorskim, i w województwie wielkopolskim, a także w mazowieckim, również są zapewnione.

W tej chwili w trakcie realizacji jest odcinek między Koszalinem a Bobolicami - 48 km drogi w budowie.

Tak wygląda kwestia związana z inwestycjami drogowymi. Jeżeli chodzi o skomunikowanie Pomorza Zachodniego, warto też w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym programie, który ułatwia komunikację, który jest ważny dla samorządowców z województwa zachodniopomorskiego. To rządowy program rozwoju dróg.

Myślę, że samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego doceniają to i dostrzegają. Dziękuję, panie ministrze. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Arkadiusz Marchewka. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Powiedział pan, że Szczecin jest miastem ładnym i wspieranym przez rząd. Z tym pierwszym się zgodzę, to prawda, ale to drugie to jest kompletna bzdura. Mam wrażenie, patrząc na to, co robicie, że Szczecin spisaliście kompletnie na straty. Minister infrastruktury mówił przecież, że w czerwcu będzie ogłoszony przetarg na zachodnią obwodnicę Szczecina. Jest prawie listopad i nie stało się zupełnie nic. Oczekuję od pana, panie ministrze, konkretów. Kiedy ten przetarg będzie zrealizowany? Przecież posłowie PiS kilkanaście miesięcy temu pięknie pozowali do zdjęć, kiedy była podpisywana umowa na tę kolej.

Czy jest pewność, że tych pieniędzy nie trzeba będzie zwracać? Dziękuję. Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Rafał Weber. Dziękuję bardzo. Jak sam pan poseł wspomniał, umowa na budowę kolei metropolitalnej w Szczecinie jest podpisana. Zgodnie z harmonogramem umownym termin wykonania i zakończenia tej inwestycji to 2023 r.

Zatrzymując się na inwestycjach kolejowych, powiedziałem na początku swojego wystąpienia, że nie działamy w próżni, że musimy pewne kwestie po naszych poprzednikach posprzątać. Warto wspomnieć o tym, jak o polską kolej, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, dbali politycy Platformy Obywatelskiej albo politycy, którzy zostali przez Platformę Obywatelską przygarnięci. Mówię tutaj np. o premierach Leszku Millerze czy Marku Belce, którzy przecież są europosłami z Koalicji Europejskiej, bo tak bodajże nazywał się komitet wyborczy w 2018 r. Z informacji, która jest też ogólnodostępna, wynika, że w latach, kiedy ci panowie rządzili Polską, a także wtedy, kiedy Polską rządzili Donald Tusk i Ewa Kopacz, na Pomorzu Zachodnim zostało zlikwidowanych, szanowni państwo, 300 km linii kolejowych. W opiłowywaniu jesteście specjalistami.

Teraz ostatnie już z serii pytań.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jezdnie autostrady A4 na odcinku węzeł Balice - ul. Kąpielowa o długości 17 km ze względu na występujące na nim duże natężenie ruchu zostaną poszerzone o trzeci pas, a węzły Kraków Balice i Kraków Skawina zostaną rozbudowane. Proszę o wskazanie zakresu prac, a także przewidywane daty zakończenia inwestycji. Dziękuję. Pani poseł Barbara Bartuś. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Bardzo często jeżdżę tą autostradą i szczególnie chcę zapytać o wjazd z lotniska Balice. Faktycznie te dwa pasy, które zostały zaprojektowane i wybudowane, to jest znacząco za mało do tego, żeby to nazywać w ogóle autostradą. Te dobre informacje, które otrzymaliśmy, napawają dużą nadzieją, bo zwykle na tym odcinku autostrada stoi. Ale nasuwa się też pytanie, jakie były przyczyny tego, że tak szybko wyczerpała się przepustowość autostrady. Dlaczego tak szybko doszło do tego, że ta przepustowość się wyczerpała?

Wszyscy - my, Małopolanie, ale nie tylko Małopolska, także Śląsk, wszyscy, którzy się tamtędy poruszają, a szczególnie korzystają z naszego lotniska w Balicach - bardzo tego wyczekują. No i Kraków. Dziękuję. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Rafał Weber. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Autostrada A4 jest główną osią komunikacyjną naszego kraju na linii wschód - zachód. Ważne jest więc, aby była drogą bezpieczną, komfortową, ale też o odpowiedniej przepustowości, tak aby można było z tej drogi korzystać w sposób nieograniczony i nieskrępowany. Dlatego w ostatnich, można powiedzieć, miesiącach zostały podjęte polityczne decyzje, które oczywiście są wynikiem merytorycznej analizy, aby autostradę A4 rozbudować - nie tylko przy Krakowie, ale szerzej.

Mamy na to zapewnione środki finansowe w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych, niemałe, bo to ponad 35 mld zł. To pokazuje, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego chce rozwijać polską infrastrukturę drogową, że dostrzega te problemy, które w tej chwili występują, i robi wszystko, aby te problemy rozwiązać. Jeżeli chodzi o A4 w okolicach Krakowa, to faktycznie jako obwodnica Krakowa pełni ona istotną funkcję w obsłudze komunikacyjnej ruchu tranzytowego, jest też równocześnie cennym uzupełnieniem układu komunikacyjnego samego miasta. W trakcie analiz, które zostały przeprowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury, uznano, iż kluczowym elementem rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu powinien być w pierwszej kolejności odcinek od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie. Obecnie funkcjonujący układ w postaci przekroju po dwa pasy ruchu w każdą stronę wyczerpuje już swoją przepustowość, co może powodować okresowe utrudnienia w ruchu i zmniejszenie przewidywalności w korzystaniu z tego odcinka autostradowej obwodnicy Krakowa. To właśnie te ogromne potrzeby transportowe, uzasadnione przez panujący na tym odcinku ruch, w dobitny sposób potwierdzają konieczność rozbudowy. Pozwolę sobie przytoczyć dane dotyczące średniorocznego ruchu drogowego według generalnego pomiaru ruchu i to będzie odpowiedź na pytanie pani poseł Bartuś.

Oczekiwany jest dalszy wzrost ruchu na autostradowej obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłem Balice a ul. Kąpielową - szacujemy, że w 2040 r. możemy się na tym odcinku spodziewać nawet 90 tys. pojazdów na dobę. Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej o trzeci pas ruchu będzie dotyczyć rozbudowy samej autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej, rozbudowy węzła Kraków Balice II, a także rozbudowy węzła Kraków Skawina. W nawiązaniu do rozbudowy węzłów należy wskazać, że działanie to przyczyni się nie tylko do poprawy przepustowości, ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Takim rozwiązaniem spełniającym oba te kryteria będzie rozbudowa obecnego węzła Kraków Skawina od układu półkoniczyny, z takim układem w tej chwili mamy do czynienia, do układu pełnej koniczyny. Jeżeli chodzi o harmonogram realizacyjny tego zadania, to w ostatnich dniach minister Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji w odniesieniu do prac przygotowawczych.

Planowane uzyskanie decyzji środowiskowej powinno nastąpić w 2024 r. Na późniejszym etapie będą podejmowane decyzje o tym, w jakim trybie będzie prowadzony przetarg wykonawczy - czy będziemy realizować tę inwestycję w trybie „projektuj i buduj”, czy też najpierw będzie przetarg na projekt, a później przetarg na budowę.

Chcemy, aby ta inwestycja została ukończona jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby rozbudowy autostrady A4 i z ogromną konsekwencją i determinacją będziemy to zadanie realizować. Dziękuję bardzo serdecznie, panie ministrze, za tę nadzieję, która płynie z pana słów.

Natomiast patrząc z naszej strony, ze strony korzystających z tych autostrad, jest troszeczkę smutno, że musimy aż tak długo czekać, ale pewnie inaczej tych procedur nie da się przeskoczyć. Jeżeli mówimy o trzecim pasie, to są miejsca, gdzie ten trzeci pas jest.

Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Poseł! Pełna zgoda, jeżeli chodzi o to, co może być, nie daj, Panie Boże, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie odpowiadało za sytuację w naszym kraju. Nawiązując do autostrady A4, chcę wspomnieć, że zgodnie z założeniami naszych poprzedników ta droga miała zostać zbudowana na Euro 2012, które odbywało się u nas i na Ukrainie. Miała ona połączyć przecież Polskę i Ukrainę, areny, na których mistrzostwa Europy się odbywały. Natomiast kiedy przyszło do realizacji, autostrada A4 nie została w całości zbudowana nawet na mistrzostwa Europy, które odbywały się w roku 2016 we Francji. Ostatnie odcinki przy Łańcucie były otwierane bodajże już w sierpniu czy we wrześniu 2016 r. Tak że nie daj, Panie Boże, aby ci, którzy wtedy odpowiadali za inwestycje infrastrukturalne, powrócili. To po pierwsze. Po drugie, autostrada A4 zostanie rozbudowana między Tarnowem a węzłem Krzyżowa w województwie dolnośląskim. Tam, gdzie w tej chwili funkcjonują dwa pasy, zostanie ona rozbudowana o jeden pas, czyli będą funkcjonowały trzy, natomiast tam, gdzie funkcjonują trzy pasy, również zostanie dokonana rozbudowa o kolejny pas. Tak jak powiedziałem, również będą rozbudowywane węzły, tak aby one mogły obsługiwać większą liczbę pojazdów w sposób przede wszystkim bezpieczny. Wygoda i komfort to jedno, ale przede wszystkim bezpieczeństwo - na tym skupiamy głównie naszą uwagę. Jeżeli chodzi o harmonogram realizacyjny, wiem, że każdy oczekuje od Ministerstwa Infrastruktury, abyśmy prowadzili nasze inwestycje dobrze i szybko. Oczywiście robimy, co możemy, żeby tak się działo, natomiast nie jesteśmy jedynym resortem, który uczestniczy w procesie inwestycyjnym. Naprawdę wiele zależy od tego, w jakim tempie wydawane są przede wszystkim decyzje środowiskowe, bo to jest w tej chwili coś, co zabiera nam najwięcej czasu, to jest coś, na czym w głównej mierze się koncentrujemy. Oczywiście jakość dokumentacji, jakość wszystkich badań środowiskowych, które są dokonywane, też ma znaczenie, ale kwestia uzyskania decyzji środowiskowej, która powinna być nie tylko ostateczna, ale również prawomocna, zabiera najwięcej czasu. Tak że liczymy na tych, którzy chcą nam w tym procesie inwestycyjnym pomóc. Jeżeli będą padały w łonie Wysokiej Izby czy w łonie komisji sejmowych propozycje legislacyjne, które pozwolą na skrócenie czasu procesu inwestycyjnego, to jako Ministerstwo Infrastruktury jesteśmy na nie bardzo otwarci. Pytanie to kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Ogłaszam 3 minuty

Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Barbarę Bartuś. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Fundusz jest impulsem dla gospodarki, która ucierpiała w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Co bardzo ważne, program wpisuje się w model zrównoważonego rozwoju. Ma wyrównać szanse rozwojowe poszczególnych jednostek czy regionów, które dotąd nie szły do przodu w tym samym tempie. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami były m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, gospodarowanie odpadami, inwestycje społeczne, tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Dzięki rządowemu funduszowi Polski Ład mamy szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, gmin, powiatów czy województw. Niezależnie od różnych pojawiających się problemów potrafimy budować finansowanie, które daje perspektywę rozwoju. Właśnie tam zostało skierowane kolejne wsparcie finansowe. Chcemy, aby mieszkańcy naszych miast i wsi nie musieli czekać latami na realizację podstawowych inwestycji. Poprzez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych poprawi się komfort życia wszystkich Polaków. Dziś Polska, korzystając ze środków budżetowych i zdrowych finansów publicznych, pokazuje, czym jest rzeczywisty rozwój gospodarczy, który służy wszystkim Polakom. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego programu inwestycji strategicznych rządowy Polski Ład. Z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego wspieramy zrównoważony rozwój i nowe inwestycje w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska, o czym już mówiłam. Ponad 2780 gmin, powiatów, miast, miasteczek otrzymuje dofinansowanie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów. Z tego wynika jednak, że ok. 3% samorządów nie otrzymało, np. w moim okręgu nowosądeckim otrzymało 58 gmin, pięć powiatów, ale dwie gminy nie otrzymały.

Czy te samorządy, które nie otrzymały, mają szansę je uzyskać w kolejnym naborze?

Czy te samorządy, które może miały problem ze stworzeniem właściwego wniosku, mogą liczyć w kolejnym naborze na jakieś merytoryczne wsparcie przy przygotowywaniu wniosków?

Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też dodatkowe wsparcie dla gmin popegeerowskich. Mam więc też pytanie, które płynie od moich samorządów, które skorzystały już z dofinansowania z tego programu dla gmin popegeerowskich. Były to niestety nie tak duże środki, jak teraz mówimy, bo to było po kilkaset tysięcy, ale mam pytanie: Czy ten program będzie kontynuowany, czy też jakoś on będzie zmodyfikowany? Teraz proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Pawła Szefernakera. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Chciałbym rozpocząć to wystąpienie od podziękowań dla praktycznie wszystkich samorządów w Polsce, dla wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków województw, którzy wzięli udział w tym pierwszym, pilotażowym naborze w ramach funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład.

Szanowni Państwo!

W trakcie rozpatrywania tych wniosków trzeba było przyjąć jakąś zasadę, która pozwoli, aby jak najwięcej wniosków było rozstrzygniętych.

Szanowni Państwo! Dofinansowanie otrzymało ostatecznie 4040 wniosków i, szanowni państwo, procedowaliśmy w ramach tych możliwości, które każda gmina stworzyła. Każda gmina, każdy powiat, każda jednostka samorządu terytorialnego miały możliwość złożyć trzy wnioski: jeden wniosek bez limitu kwoty, jeden wniosek do 30 mln i jeden wniosek do 5 mln zł. Szanowni Państwo! Ostatecznie dofinansowanie uzyskało 97% samorządów. Te 3% samorządów, które nie uzyskały.

W przeważającej większości - oprócz tych samorządów, które nie złożyły wniosków - samorządy, które nie otrzymały wniosków w pierwszym naborze, to samorządy, które złożyły wnioski albo bez limitu kwoty, albo na bardzo duże kwoty, czyli do 30 mln zł, co niestety przekraczało możliwości tego naboru. Szanowni Państwo! Namawiamy wszystkich, także Bank Gospodarstwa Krajowego razem z wojewodami będzie organizował w tym i kolejnym tygodniu we wszystkich województwach w Polsce spotkania z samorządowcami, tak żeby przekazać informacje, wnioski z pierwszego naboru, tak żeby wszyscy mogli jak najlepiej przygotować się do kolejnych naborów.

Szanowni Państwo! Kwota przyznanego dofinansowania w podziale na najważniejsze inwestycje.

Wśród tych największych gmin, ale także tych małych ewidentnie jest to najważniejszy problem inwestycyjny, największa potrzeba, gdzie nie ma też środków zewnętrznych z innych programów na to, aby gmina czy powiat były beneficjentem środków zewnętrznych i mogły inwestować. W związku z tym najwięcej, bo właśnie blisko 17 mld zł, przeznacza się na infrastrukturę drogową, na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Szanowni Państwo! Pan premier zapowiedział kolejny nabór w ramach funduszu inwestycji strategicznych. Ten nabór odbędzie się jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku będzie specjalny komponent programu dedykowanego gminom z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W związku z tym te nabory będą jeszcze w tym roku. W najbliższych tygodniach będzie o nich informowana opinia publiczna, jak tylko decyzje, w postaci uchwały Rady Ministrów, dotyczące tych naborów zostaną podjęte. Szanowni Państwo! Dziś również otrzymałem pismo od Związku Miast Polskich, gdzie wskazano parę przypadków w kraju. Włodarze gmin, części miast uważają, że nie otrzymali środków w wymiarze proporcjonalnym.

Szanowni Państwo!

Wczoraj rozmawiałem choćby z panem burmistrzem Lądka-Zdroju, który pytał mnie o to, z czego wynikają takie, a nie inne wyniki. Także Bank Gospodarstwa Krajowego jest otwarty na to, aby rozmawiać z samorządami.

Przygotowujemy się do kolejnych rozdań.

Chciałbym również podziękować pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy z nami pracowali. Chodzi o opiniowanie ponad 8 tys. wniosków. Pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pragnę złożyć podziękowania na ręce obecnej tutaj pani minister Izabeli Antos. Pozostajemy do państwa dyspozycji, do dyspozycji parlamentarzystów, samorządowców.

Bardzo dziękuję panu ministrowi. Informuję, że zgłosili się posłowie do dyskusji. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zapisać się do głosu? Bardzo proszę. Po panu pośle zamykam listę mówców.

Tym samym państwo ograniczycie liczbę wystąpień, jeżeli. Są podzielone głosy. Bardzo proszę, pani poseł Borowiak. Bardzo dziękuję. Ponad 1250 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład dla województwa kujawsko-pomorskiego, w tym ponad 737 mln na 140 inwestycji, które zmienią oblicze mojego regionu, to 140 przykładów realnego wsparcia ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości dla samorządów i dla mieszkańców.

To konkrety, nie puste obietnice. Pytanie: Kiedy samorządy mogą zacząć realizować inwestycje, na które otrzymały bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Budżet państwa to jest ten dokument, w którym powinno się szukać informacji o programach rozwojowych, ale w tym budżecie niczego takiego nie znajdziemy. Znajdziemy za to blisko 40 mld środków mniej dla samorządów. To efekt zmniejszenia dotacji i wpływu z podatku dochodowego 12 mln zł. Nic dziwnego, że dzisiaj PiS w obliczu katastrofy dyplomatycznej w Brukseli i blokady środków z Krajowego Planu Odbudowy, za którą ponosicie pełną odpowiedzialność. Ratujecie sytuację, uruchamiając po raz kolejny pozabudżetowe środki z emisji obligacji, zadłużając nas na kolejne dziesiątki miliardów złotych. I od razu zaznaczę: te pieniądze, cytując klasyka, samorządowcom się po prostu należą. Zresztą ten wasz ład to zaledwie 10% Krajowego Planu Odbudowy, a do samorządów miało przecież trafić 30%. To taka PiS-owska sprawiedliwość. Jeszcze w niedzielę mieli mieć 27 mln zł. Proszę powiedzieć, który z sądeckich posłów zabiegał o mniejszą kasę dla Nowego Sącza. Chcemy znać to nazwisko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Program inwestycji strategicznych ma zmienić Polskę biedną w Polskę bogatą, tylko jest pytanie, w których regionach. W ramach tego wielkiego PiS-owskiego programu Bydgoszcz ma otrzymać zaledwie 35 mln zł na inwestycje, tj. 100 zł na jednego mieszkańca. Niestety w Inowrocławiu jest jeszcze gorzej, bo mają otrzymać 69 zł na jednego mieszkańca i w sumie 5 mln zł. A w poprzednich programach wsparcia rządowego Inowrocław nie otrzymał pieniędzy na żaden ze złożonych wniosków. W związku z tym mam pytanie: Jakie są oficjalne przyczyny takiej polityki rządu, że mieszkańcy Bydgoszczy, Inowrocławia nie zasługują na te pieniądze? Jakie są wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące zakwestionowania tych wniosków? Mieszkańcy oczekują dokonania korekt przez rząd w podjętych decyzjach dotyczących przyznawania tych środków. Natomiast mam pytanie: Gdzie w budżecie państwa zawarte są pieniądze na rozdawanie tych środków? Gdzie te pieniądze są? Ile Polacy będą musieli ostatecznie zwrócić pieniędzy, na które zadłużyliście w tym momencie państwo? Bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie, do kiedy budżet będzie musiał zwrócić te pieniądze. Czy będzie drugi konkurs i czy w ramach tego konkursu nadrobicie te działania, w których chociażby taki Inowrocław ma 69 zł (Dzwonek) na jednego mieszkańca?

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Ten wasz Polski Ład to tak naprawdę brak ładu i składu, a przede wszystkim brak odpowiedzialności za finanse państwa i brak odpowiedzialności za finanse samorządów. Samorządy lokalne na waszych zmianach podatkowych będą tracić ok. 10 mld rocznie. Na stronie natwojkoszt.pl, bo to jest na koszt nas wszystkich, samorządy polskie podsumowały, że w ciągu 10 najbliższych lat na zmianach podatkowych stracą niemal 150 mld zł. Jeszcze gorzej jest, kiedy analizujemy poszczególne przypadki. Dąbrowa Górnicza w waszym arkuszu Excela otrzymała 20 mln na drogę, ale straci w przyszłym roku 48 mln wpływów do budżetu. Miasto Tychy, moje rodzinne miasto, otrzymało 47 mln na budowę dwóch wiaduktów, o które zresztą prosimy od wielu, wielu lat. Ale w przyszłym roku stracimy 52 mln wpływów do budżetu. Ja wiem, projektujecie tzw. rekompensatę, ale ta rekompensata to tylko połowa środków, które normalnie do budżetu by wpłynęły. Rybnik nie otrzyma nic, a straci 31 mln zł. Te środki są poza długiem, one są poza budżetem, one są poza regułą wydatkową. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Lidia Burzyńska, klub Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Program Inwestycji Strategicznych pokazuje, szanowni państwo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma i realizuje program, na który umówił się z Polakami. Zrównoważony rozwój naszej ojczyzny, a nie, tak jak totalna opozycja chciała i realizowała, dyfuzyjność, pokazuje, że środki nie trafiają według podziału na liczbę mieszkańców, bo to jest dyfuzyjność, tylko trafiają do samorządów. Przykładem tego, szanowni państwo, jest. okręg nr 28, z którego mam zaszczyt być posłem. Na cały okręg, czyli 5 powiatów, 344 mln trafiły do samorządów. Powiat kłobucki - 77 mln. Na co są przeznaczone? Ano na to, czego nie otrzymały, kiedy państwo rządziliście, na infrastrukturę drogową, na infrastrukturę sportową, na budowę przedszkoli, na kanalizację, na bazę sportową.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Każda złotówka przeznaczona na inwestycję w samorządzie jest szczególnie cenna, bo samorządy od lat generują 3/4 inwestycji publicznych w Polsce i oglądają dokładnie każdą złotówkę. Ograbialiście i ograbiacie od lat budżety samorządów, że ledwo już, można powiedzieć, zipią, więc dobrze, że w końcu postanowiliście oddać część tych środków.

Zapowiadacie, że to będzie jeszcze wyższa kwota. Dlaczego zadłużacie budżet państwa na następne pokolenie, kiedy wystarczy dopiąć tylko Krajowy Plan Odbudowy, z którego możemy dostać 110 mld zł bezzwrotnych dotacji? To po pierwsze. Dlaczego udzielacie samorządom tylko promes? Samorząd będzie więc musiał wyłożyć na całość inwestycji swoje pieniądze, a dopiero potem może te pieniądze zostaną zwrócone. Wyobraźmy sobie gminkę, która ma budżet wynoszący 30 mln i dostaje środki na inwestycje - 8 mln.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Rozmawiamy dzisiaj o Programie Inwestycji Strategicznych, w szczególności o pierwszej edycji dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego. Na sali we wprowadzeniu padły słowa, że wyboru dokonano z uwagi na preferowane inwestycje dla małych, lokalnych, rodzimych przedsiębiorstw, które mogą zrealizować te inwestycje lokalnie. Panie Ministrze! Bardzo proszę pana o informację, czy i kiedy będzie druga edycja. Kiedy środki z pierwszej edycji trafią do jednostek samorządu terytorialnego oraz skąd dokładnie będzie czerpane źródło finansowania tych inwestycji? Bardzo proszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Takim miastem jest np. Bielsko-Biała.

Tymczasem okazuje się, że jeżeli popatrzymy na województwo śląskie, to miasto Bielsko-Biała, jeżeli chodzi o kwotę dofinansowania, jest dopiero niemalże na samym końcu, znajduje się na czwartym miejscu od końca.

Panie Ministrze! Co decydowało o tym, że takie miasta jak Bielsko-Biała, które utraciły status województwa, które dzisiaj potrzebują tego wsparcia, tego wsparcia nie otrzymują? To jest wbrew temu, co powtarzacie, czyli wbrew wspieraniu mniejszych ośrodków.

Panie Ministrze! Polski Ład wraz z Programem Inwestycji Strategicznych są odpowiedzią na potrzeby Polaków, a także samorządów i samorządowców. Jest on, co podkreślałem wielokrotnie, największym takim programem w historii wolnej i demokratycznej Polski.

Dziękując za 2 mld zł wsparcia dla samorządu województwa śląskiego, chciałbym poprosić o wskazanie największych inwestycji w województwie śląskim, z uwzględnieniem Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Będzina, Zawiercia. Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, iż łączna kwota dofinansowania w skali kraju to 23 mld zł. Chciałbym zapytać o Program Inwestycji Strategicznych, kolejne edycje. Czy takowe są planowane?

Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! PiS najpierw okradł samorządy niczym kontenery PCK [[Oklaski]] - w dodatku nazwał ten proceder Polskim Ładem - po czym kilka dni temu z przytupem ogłosił, że samorządom coś daje. A wystarczyło nie zabierać. Premier Morawiecki oszukuje, gdy mówi, że to jest największy projekt inwestycyjny w samorządach. Jest tylko jeden warunek. Rząd PiS-u ma nie wypowiadać III wojny światowej Unii Europejskiej, tylko wykonać wyrok TSUE. Popłyną strumienie pieniędzy do polskich samorządów, dużo większe i w dodatku nie z długu, bo te tekturowe czeki, które rozdajecie, to są obligacje, to jest dług, w dodatku to obciąży budżet za 10 lat. PiS rozdaje, kolejne rządy i pokolenia będą spłacać. Te pieniądze rozdajecie poza kontrolą Sejmu. Bo chociaż jest Komisja, to - uwaga - przepisy, które sami stworzyli, pozwalają, żeby premier Morawiecki jednoosobowo przekreślił werdykt Komisji i nawet wstawił tam swoje projekty. Czyli będzie jak z funduszem Ziobry, tylko jeden rozdaje miliony, drugi będzie rozdawał miliardy. To jest wreszcie likwidacja autonomii samorządów. Będzie decydował nawet, która ulica. Dziękuję bardzo.

Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Każde wsparcie państwa w realizacji inwestycji samorządów jest ważne. My możemy toczyć spór dotyczący kontroli wydatkowania tych środków finansowych, zaciągania długu na przyszłość, niemniej jednak z punktu widzenia społeczności lokalnych środki te są istotne i ważne w kontekście rozwoju.

Chciałem zapytać, czy ten program będzie kontynuowany i czy będą również kierowane środki na wyrównanie dostępu do infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, ale także dostępu do świetlicy wiejskiej czy strażnicy. Drugie pytanie dotyczy mimo wszystko nierównego potraktowania w tej edycji niektórych samorządów.

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Samorządy działają w imieniu mieszkańców, dla swoich mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców, dlatego wsparcie samorządów, wsparcie mieszkańców musi być sprawiedliwe. Stąd moje wielkie zdziwienie, że w regionie świętokrzyskim dwa powiaty, sandomierski i buski, nie otrzymały ani złotówki.

Sądzono, że teraz zrobi się coś dla mieszkańców. Busko-Zdrój też nie otrzymało ani złotówki. Czy ten błąd to, mam nadzieję, niedopatrzenie zostanie naprawione w najbliższym czasie, przy kolejnych podziałach, aby po prostu. Bo wiemy, że takie sytuacje powodują ogromne niezadowolenie wśród mieszkańców. Pamiętajmy, że te kryteria muszą być przejrzyste, muszą być obiektywne, nie może być uznaniowości. Wiemy, że w sam raz te.

Wysoka Izbo! Ja z wielką satysfakcją przyjąłem informację o wynikach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, bo to wielka szansa na zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski - to 2785 miasteczek, powiatów i gmin, do których trafi ponad 23 mld zł na dofinansowanie ponad 4 tys. inwestycji, zwłaszcza inwestycji lokalnych, z których codziennie korzystamy i które bezpośrednio wpływają na jakość i komfort naszego życia. To jest budowa i rozbudowa szkół, żłobków, przedszkoli, a także obiektów sportowych, przychodni zdrowia, terenów rekreacyjnych i to są liczne inwestycje drogowe. Z kolei lokalni przedsiębiorcy, realizując te inwestycje, mogą rozwijać swoje firmy, tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się tym samym do rozwoju niemal każdej gminy w Polsce, czyli miejsc, w których mieszkamy, żyjemy i realizujemy nasze codzienne potrzeby życiowe. Krótko mówiąc, Rządowy Fundusz Polski Ład to jedyny od dziesięcioleci program na miarę naszych marzeń, potrzeb i oczekiwań społecznych, za który chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Cóż, tak już będzie: jedną ręką rząd samorządowcom zabiera i zmusza do cięć, wydatków, a drugą bez kryteriów i zasad rozdziela tylko część zabranych wcześniej pieniędzy. Pomimo tego, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, tylko te pochodzące z podatków Polaków, uruchomił rozdawniczą rządową maszynę propagandową w gminach, miastach i powiatach. Drugi i trzeci etap w przypadku Funduszu Inwestycji Lokalnych pokazał rozdawnictwo publicznych pieniędzy, które rząd potraktował jak polityczny łup i rozdał bez trybu, lekceważąc mieszkańców tych miejsc, gdzie nie dotarła ani jedna złotówka.

Ale nie, bo sprawiedliwość po waszemu w rekompensowaniu strat samorządom nadal pokazuje olbrzymie dysproporcje.

Samorządowcy mówią wyraźnie: decentralizacja postępuje, rząd niszczy samorządność, rząd ubezwłasnowolnia samorządy, publiczne pieniądze rząd rozdaje bez kryteriów.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Elżbieta Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pani poseł? Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Polski Ład to ponad 160 mln zł dla samorządów województwa małopolskiego, rekordowa kwota dla królewskiego miasta Krakowa.

Dzięki dotacji rządowej przebudowany zostanie w końcu rynek w Słomnikach i rynek w Mogilanach. Polska pięknieje. Szanowni Państwo! Chciałabym z tego miejsca w imieniu samorządowców województwa małopolskiego podziękować. za wspaniałą współpracę rządu z samorządami. Pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Pani Marszałek!

Ale wy prowadzicie politykę pod hasłem: po nas choćby potop. Traktujecie pieniądze z długu tak samo jak te pieniądze, które moglibyście pozyskać, gdyby nie Ziobro, z Krajowego Planu Odbudowy i z funduszy europejskich. Kiedyś ktoś będzie spłacał, ale teraz już płaci za to ze swojej kieszeni każdy Polak, ponieważ najnowsze dane mówią o drożyźnie: 6,8% według CBOS. Co to oznacza? Wasza polityka to jest polityka wydawania pieniędzy, których nie macie. Wasza polityka to jest polityka zadłużania przyszłych pokoleń. Wasza polityka to jest polityka zakładająca, że kupimy sobie przychylność samorządów w ten sposób, że w tej chwili pożyczymy pieniądze po to, żeby rozdać. A moglibyśmy mieć pieniądze z Unii Europejskiej, gdyby nie Ziobro. Płacimy za wasze nieumiejętności, płacimy za wasze niezgulstwo i płacimy za wasze silne poczucie bycia bezkarnymi. A wystarczyłoby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i kilkadziesiąt miliardów euro trafiłoby do Polski. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pamięć, szczególnie opozycji, gdy była władzą, jest ulotna.

Przepisy te spowodowały, że gminy z dnia na dzień nie miały skąd wziąć środków na wkład własny do programów unijnych. Więc co z tego, że były programy unijne, skoro nie było pieniędzy na to, żeby można było inwestować. Taka była prawda, 60%.

Przez te wszystkie lata nie było skąd wziąć na wkład własny. Kończąc, chciałbym bardzo podziękować za 110 mln dla powiatu piotrkowskiego. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie z PiS-u! Krótką macie pamięć. Ale teraz mówimy o stanie obecnym. Inflacja, drożyzna+.

Każecie im zapłacić za długi szpitali. Nie wykonujecie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zabraliście pieniądze samorządom w Polskim Ładzie.

Bilans tego rozważenia 6 lat dla samorządów to mniej niż zero. Mniej niż zero. Pytanie do pana ministra: Dlaczego w powiecie mieleckim samorząd gminy Przecław (Dzwonek) nie otrzymał pieniędzy? Po pierwsze, gdzie. i kto miał upoważnienie do rozdawania [[Dzwonek, oklaski]] tekturek? Panie pośle, bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Cóż można powiedzieć o pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład?

Osobne słowa podziękowania mam dla kierownictwa Banku Gospodarstwa Krajowego na czele z panią prezes Beatą Daszyńską-Muzyczką. Dziękują Kołobrzeg i wszystkie gminy powiatu kołobrzeskiego. Dziękują Koszalin i gminy powiatu koszalińskiego. Dziękują Szczecinek i gminy powiatu szczecińskiego. Dziękują miasto Sławno i powiat sławiński. Dziękuje gmina Darłowo itd., itd., itd. Panie Premierze! Panie Ministrze! Pani Prezes! Wspaniały okres zrównoważonego rozwoju małych ojczyzn, regionów Polski. Wkrótce, proszę państwa, żadna gmina w Polsce nie będzie funkcjonować daleko od szosy. Jeszcze kilka lat temu minister finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL-u twierdził, że nie ma pieniędzy i nie będzie. Okazuje się, że pieniądze są i będą. Na spotkaniu w Wałczu samorządowcy stwierdzili, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Wysoka Izbo! Rządowy fundusz inwestycji strategicznych. Cztery słowa, a w każdym kłamstwo.

Tworzy w to miejsce mechanizm iście feudalny, w którym samorządy idą po prośbie do pana i władcy, a ten w łaskawości swojej, za przyczyną lokalnych dworzan, [[Oklaski]] wręcza im uroczyście tekturowe czeki, po czym następują równie uroczyste podziękowania za starania miejscowych kacyków. W rezultacie mamy system wasalny, w którym wszystko, nawet oczyszczanie przydrożnego rowu lub trawa na boisku, zależy od pańskiego oka władzy na Nowogrodzkiej.

Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Do powiatu zduńskowolskiego, w którym rządzi Platforma Obywatelska - 55 mln zł.

Na co może liczyć gmina Wieluń? Panie pośle, dziękuję. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! O Wieluniu będzie dziś często słychać, bo to jest jedyna gmina w województwie łódzkim, która została pominięta. I jest oświadczenie burmistrza Wielunia. Gmina Wieluń po raz kolejny została pominięta przy podziale środków rządowych, tym razem w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy jedynym miastem w województwie łódzkim, które nie otrzymało dotacji z dotychczas ogłoszonych przez rząd konkursów. To wstyd. To także hańba dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jesteście rekordzistami, gdy chodzi o hipokryzję, jesteście rekordzistami, gdy chodzi o inflację, jesteście rekordzistami, gdy chodzi o zadłużanie Rzeczypospolitej. Te długi będą spłacały następne pokolenia. Ale przypomnę, że rząd Platformy Obywatelskiej rozpoczął wielką budowę Rzeczypospolitej, [[Oklaski]] wielką budowę samorządów, samorządów, które wy ograbiacie.

Pani poseł Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi, bardzo dziękuję rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że te środki możemy wykorzystać na drogi, na przedszkola, na stadiony, na oczyszczalnie, na wodociągi, które są bardzo potrzebne w województwie podkarpackim. Dlatego tyle środków przeznaczono dla województwa podkarpackiego, ponieważ tam są wieloletnie zaniedbania. Nie dbaliście o Bieszczady, nie dbaliście o miasta, nie dbaliście o małe miasteczka. Dzięki tym środkom w moje rodzinnej miejscowości może zostać zmodernizowana oczyszczalnia, mogą zostać wybudowane drogi w Bieszczadach.

Potrzebują one na oczyszczalnie, jak np. gmina Krasne, która potrzebuje prawie 26 mln zł. Pan poseł Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Samorząd realizował wielkie inwestycje infrastrukturalne, wielkie inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej. To jest praktyka życia w Polsce od 30 lat. Były próby ograniczania wpływów samorządu terytorialnego, ale nikt nie zrobił tego tak jak wy. Znowu wracamy do modelu PRL-owskiego, w którym decyzję o sprawach lokalnych, sali gimnastycznej, jak tutaj słyszeliśmy, drogach, zapadają w Warszawie, centralnie. To jest powrót do komuny. Przecież ten fundusz inwestycji strategicznych to jest de facto fundusz propagandy wyborczej PiS-u. Gdybyście te pieniądze podzielili według algorytmu, to nie trzeba byłoby pisać żadnych wniosków, nie trzeba byłoby armii urzędników rządowych, żeby przyznawać te pieniądze. Samorządy powinny (Dzwonek) te pieniądze dostać według algorytmu. Pan poseł Lipiec. Pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziś jest szczególny dzień, kiedy możemy otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych - mówił w ostatni poniedziałek premier Morawiecki. I kontynuował: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o wielkości powyżej 23 mld to program jedyny i największy przez ostanie 30 lat w czasach wolnej Polski. Panie Premierze! Która to już największa księga inwestycji otwierana przez pana w ciągu ostatnich 6 lat? Która to już księga bajek? Przypominam, że był plan Morawieckiego, była piątka Morawieckiego na 100 dni, później Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Nie ma tanich 100 tys. mieszkań.

Przykładem jest choćby moje miasto Bielsko-Biała. Kogo pan, panie premierze, tym razem chce oszukać? Zaczęłam cytatem z pana premiera i zainspirowana sięgnęłam do książki „Pinokio”

Pani poseł Ewa Malik, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W tym naborze przeznaczono na inwestycje prawie 24 mld zł. Z ciekawości zapytam: Jaką kwotę pan premier Morawiecki przeznaczy w kolejnym naborze na właśnie tak liczne, wspaniałe inwestycje? że program będzie dostosowywany do potrzeb gmin, więc to też jest ciekawą dla mnie rzeczą. Ale, tak szczerze mówiąc, występuję w imieniu mieszkańców gmin i miast usytuowanych w moim okręgu wyborczym. Duże miasta na prawach powiatu, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, pięknie dziękują nam za bardzo duże pozyskane środki. Także dwa ziemskie powiaty, będziński i zawierciański, z ogromną radością przyjęły właśnie otwarcie przed nimi tych wszystkich możliwości dodatkowego inwestowania na rzecz potrzeb, które zamieściły we wnioskach, bo to wcale nie jest tak, jak tutaj pani poseł z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że przyznajemy pieniądze, że rząd przyznaje pieniądze, ale tak naprawdę przyznaje je jakby bez wiedzy gmin. Otóż nie.

Dziękuję. Wysoka Izbo! Wasz Program Inwestycji Strategicznych w ramach tzw. polskiego nieładu to nic innego jak propaganda i szczyt manipulacji. Zasady rozpatrywania wniosków samorządów to w dużej mierze skopiowane procedury, jakie obowiązywały w Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nadal są one mało transparentne i pozwalają na wydanie dużej części pieniędzy według partyjnego klucza. Doskonale widać to na przykładzie mojego regionu. Miasto Bielsko-Biała, które według narzędzia wyliczającego koszty Polskiego Ładu stworzonego przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich straci 86 mln rocznie, na remont kąpieliska Panorama otrzyma zaledwie 25 mln zł. Takie są relacje. Bez wyjątku - na wszystkie, które zgłosiły. Przykład ten pokazuje, że znowu próbujecie rozdzielać pieniądze w myśl zasady „swoi+” Poprzez zadłużenie Polaków na 24 mld zł w obligacjach chcecie zrekompensować samorządom stratę 150 mld zł z tytułu utraconych dochodów, ale jak zwykle robicie to nieudolnie. Kiedy wreszcie przyjmiecie nową ustawę o (Dzwonek) dochodach jednostek samorządu terytorialnego? Inflacja blisko 7%. Pani poseł, bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pierwsza edycja pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za nami. Uzyskane fundusze są cennym wsparciem działań samorządów, oczywiście tych, które je otrzymały. Moje pytanie brzmi: Czy jest możliwość zmiany projektu po uzyskaniu promesy na wykonanie konkretnej inwestycji? Dotyczy to czasu realizacji inwestycji. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Samorządy od lat czekają na uczciwą relację z rządem, na realne pokrywanie kosztów zadań, jakie realizują w imieniu państwa. Oczekują partnerstwa i zaufania, wiary, że znają lepiej potrzeby mieszkańców i lepiej zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze. Rząd daje, a w zasadzie zadłuża Polskę, nie potrafiąc skutecznie pozyskać 110 mld zł dotacji z Unii Europejskiej, i wreszcie ogranicza dochody samorządu terytorialnego. PiS niestety nie rozumie samorządu. Zamiast rozdawać promesy, papierowe czeki, zostawcie te pieniądze w gminach, powiatach i województwach. Byłoby przynajmniej sprawiedliwie. Ale jest, jak jest. Proszę zatem o udzielenie informacji, jakie kryteria decydują o życzliwości rządu i czy samorządy mogą odwołać się od tych decyzji, które są podejmowane. Wysoka Izbo! Polski Ład to systemowy program zadłużania Polski. Można by sparafrazować słynny cytat i powiedzieć: Jeszcze nigdy tak wielu nie zostało zadłużonych tak bardzo przez tak nielicznych. Dziękuję. Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych jest programem, który dowodzi, że współpraca rządu z samorządem jest bardzo dobra. Ja się nie dziwię, że taką wściekłość u państwa budzi ten program, bo wytrącamy wam ten argument z ręki - nie możecie już powtarzać, że rząd nie współpracuje z samorządami. 99% samorządów otrzymało dofinansowanie. W powiecie brzeskim wszystkie samorządy otrzymały środki finansowe na ważne inwestycje, które nie były realizowane od wielu lat. W powiecie bocheńskim to np. przedszkola, drogi, mosty. To są konkretne zadania, które będą realizowane w ramach Polskiego Ładu. Szanowni Państwo! Tak bardzo narzekacie, że na Polskim Ładzie tracą samorządy. To jest nieprawda.

Podam konkrety na przykładzie gminy Brzesko.

Ponieważ powoli zbliżamy się do końca tego punktu, apeluję do wszystkich państwa, by przede wszystkim nie przedłużać i naprawdę skracać wypowiedzi, żeby każdy mógł zadać pytanie. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zadam pytanie: Dlaczego rząd ograbił niektóre samorządy? Mówicie o podziałach na województwa. Wszędzie tam, gdzie są wasi wyborcy, są oni wynagradzani. Dlaczego to robicie? Mówicie, że za waszych rządów jest tak dobrze, ale ludzie, z którymi się spotykam na co dzień, mówią zupełnie co innego.

Jak gmina głosuje na PiS, wtedy ma większe dotacje. Słucham i nie przeszkadzam. Natomiast chciałam państwu powiedzieć, że dokładnie pamiętam PRL. Pamiętam, jak to wyglądało. U was jest podobnie. Przyjeżdża cała świta, żeby otworzyć kawałek drogi.

Odbyłem w województwie podlaskim, z którego sprawuję mandat poselski, w ostatnich dniach cały szereg spotkań z samorządowcami. Wszyscy wyrażają naprawdę wielką wdzięczność polskiemu rządowi, podkreślając, że jeszcze nigdy takich pieniędzy, tak dużych środków finansowych na rozwój Polski lokalnej w gminach, powiatach, miastach i regionach nie było.

Przecież, szanowni państwo, to jest niebywała sytuacja. Jeżeli ktoś to kwestionuje, po prostu nie chce rozwoju Polski. To jest po prostu działanie na szkodę przyszłości. Jeszcze raz powtarzam: szanujmy się nawzajem i skracajmy swoje wypowiedzi, żeby każdy mógł zabrać głos. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W ubiegły poniedziałek na zamku w Nidzicy panowała wielka radość - spotkanie samorządowców z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Proszę, mogliście państwo tam być. Ja byłam tam obecna.

To są fakty, szanowni państwo.

Szanowni państwo, w moim okręgu wyborczym wsparcie otrzymały wszystkie gminy, wszyscy samorządowcy są szczęśliwi. Dzięki tym pieniądzom powstaną nowe odcinki dróg, infrastruktura sportowa, oczyszczalnie ścieków. Pan poseł Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Premier Mateusz Morawiecki na początku tygodnia ogłosił wyniki rządowego funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład. To ponad 23 mld zł na poprawę infrastruktury i podniesienie jakości życia mieszkańców miast, miasteczek i wsi. To szansa na zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do życia dla Polek i Polaków, również dla mieszkańców Wielkopolski, także południowej Wielkopolski. Do samorządów województwa wielkopolskiego na strategiczne inwestycje trafi ponad 1980 mln zł. Będzie ona przeznaczona na remonty dróg, obiektów sportowych, tras rowerowych, także sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wymianę źródeł ciepła z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Niektóre z tych inwestycji do tej pory nie miały szans na realizację, np. droga Przygodziczki - Biskupice w powiecie ostrzeszowskim. I tak, do samorządów powiatu kępińskiego trafi ponad 64 mln zł, powiatu ostrzeszowskiego - ponad 52 mln zł, powiatu ostrowskiego - ponad 82 mln, powiatu krotoszyńskiego - 32 mln, powiatu pleszewskiego - ponad 32 mln, powiatu jarocińskiego - ponad 32 mln, powiatu kaliskiego - prawie 70 mln zł plus 44 mln zł dla miasta Kalisza. Cieszę się, że do południowej Wielkopolski spłyną aż tak duże środki, za to bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi i panu ministrowi. Pani poseł Ewa Szymańska, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Jak już tu przedmówcy wspomnieli, pierwsza edycja Polskiego Ładu za nami. Samorządy otrzymały prawie 24 mld zł. Na tej sali były ze strony opozycji głosy, że nie stosuje się algorytmów, że nie bierze się pod uwagę liczby mieszkańców gmin. Proszę państwa, przy braniu pod uwagę liczby mieszkańców niektóre gminy nie dostałyby w ogóle pieniędzy. Co ma zrobić mała gmina popegeerowska na dużym obszarze, jak nie miała wkładu własnego i nie była brana w związku z tym pod uwagę, nie mogła złożyć wniosku? Tam drogi są fatalne, nie ma infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej, mimo że w sąsiednich gminach, bogatszych, inaczej świat wygląda. Dzisiaj te gminy dziękują nam, że wzięliśmy pod uwagę inne kryteria. Pieniądze były dzielone na wnioski, nie na widzimisię naszego rządu czy kogokolwiek innego. A moje pytanie dotyczy kolejnych edycji Polskiego Ładu.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Czas płynie, a narracja opozycji jest taka sama. Kiedy w lipcu 2020 r. rozstrzygnięty został pierwszy nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, też mówiliście o czekach bez pokrycia, o tekturkach i o karteczkach. A za te pieniądze, które wtedy trafiły do samorządów, wykonano naprawdę bardzo wiele potrzebnych inwestycji. Województwo świętokrzyskie, piękne, ale nie największe, otrzymuje blisko 1 mld. Mój powiat ostrowiecki na budowę stadionu lekkoatletycznego dla młodzieży z zespołu szkół mistrzostwa sportowego dostaje 16 mln i są to pieniądze, na które czekano kilkanaście lat.

I to marszałek wnioskował o to, żeby w moim mieście to zrobić. Szanowni Państwo! Ja naprawdę dziękuję za ten program i z nadzieją oczekuję na kolejną edycję. Pan poseł Aleksander Mrówczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Do opozycji totalnej: wasze 8 lat rządzenia. Damy radę. Wyście rozwijali duże aglomeracje, a my dochodzimy do małych gmin. Zrównoważony rozwój. Wasi samorządowcy nam dziękowali, a wy cały czas krzyczycie, zawsze to robicie. Polacy na to się już nie dadzą nabrać, absolutnie nie. Nie kłamcie, każdy samorząd otrzymał środki, chyba że o zbyt duże środki występował. Szanowny Panie Ministrze! Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować z serca jako poseł rządowi Zjednoczonej Prawicy z Mateuszem Morawieckim na czele. Moje pytanie: Czy w kolejnej edycji tego programu samorządy będą mogły składać wnioski o środki na rozwój linii światłowodowej? Pan poseł Włodzimierz Tomaszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Moje podstawowe pytanie do opozycji jest takie: Ile ta opozycja dała, kiedy była przy władzy, samorządom na inwestycje?

To są niebotyczne kwoty. Jeżeli Platforma mówi, że dodawała samorządom, to pokażcie, ileście dodawali. Chcę państwu przypomnieć: realizowałem te ustawy dotyczące kompetencji powiatów i województw, ale jeśli chodzi o decentralizację finansów publicznych, to przecież samorządy dostały 25% mniej, niż miała to administracja rządowa. A teraz dopiero dodaje się te pieniądze i to jeszcze najważniejsze - inwestycyjne. Będzie wspólne dobro, ponieważ będą przez te inwestycje wzrastały wpływy podatkowe do samorządów i do budżetu państwa i będą miejsca pracy. Pan poseł Jerzy Paul, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Rok 2020 był chyba rokiem najtrudniejszym po II wojnie światowej dla gospodarki, służby zdrowia, edukacji czy wielu innych dziedzin naszego życia. Rok 2021 jest czasem odbudowy po koronawirusie, ale również przygotowania się do wielkich inwestycji, które będą realizowane w roku następnym. Z wielkim optymizmem patrzymy na rok 2022, bo to rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył i sfinansował program Polski Ład. Te 23 mld zł, które trafią do polskich samorządów, pozwolą zrealizować inwestycje, których wykonanie ze względu na brak środków finansowych było przekładane przez lata. Wiem, o czym mówię, bo kiedy byłem burmistrzem miasta i gminy Nowa Sarzyna w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, pieniędzy na wszystko brakowało, a właśnie szczególnie na inwestycje, które były wtedy praktycznie wstrzymywane. A teraz polski rząd wsparł finansowo prawie każdą gminę w Polsce, nie patrząc na przynależność partyjną czy na poglądy polityczne. Dlatego jako poseł z Podkarpacia i ziemi leżajskiej w imieniu swoim i samorządowców dziękuję panu premierowi i polskiemu rządowi za miliardy złotych, które trafią do wszystkich miast i gmin w całej Polsce. Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Więc idźcie do swoich prezydentów, wójtów, burmistrzów i powiedzcie: nie bierzcie pieniędzy z tego funduszu. A te inwestycje, które były inwestycjami marzeń za waszych rządów, zrealizujecie być może, jak wy przejmiecie władzę, w co wątpię. Szanowni Państwo! Dziękuję bardzo za prawie 2 mld zł dla Wielkopolski, za ponad 44 mln dla Kalisza i wielu innych miast południowej Wielkopolski. Kiedy rozmawiałem z burmistrzami i prezydentami, wójtami, sołtysami z PSL-u, z Lewicy, z Platformy, z PiS-u, mówili jedno: dzięki tym środkom realizujemy marzenia, bo to, co opisali we wnioskach, to były nasze marzenia sprzed lat, raczej nie do zrealizowania. Więc dziękujemy rządowi Mateusza Morawieckiego za te pieniądze, bo będziemy mogli zrealizować inwestycje, na które czekają obywatele. I moja prośba już na koniec, panie ministrze. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Otrzymujemy telefony, otrzymujemy e-maile od włodarzy gmin, od mieszkańców gmin z ogromnymi podziękowaniami, bo wreszcie znajdują się takie miejscowości, że będzie w takim, a nie innym miejscu zrobiona zapomniana droga i choćby nie wiem, jak państwo chcieli zaklinać rzeczywistość, szanowna opozycjo, niestety ta rzecz się dzieje i rzeczywiście miliardy płyną do samorządów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Niektóre gminy w ogóle nie otrzymały dofinansowania, bo 97% jednostek samorządu terytorialnego to dofinansowanie otrzymało.

Jest jednym z największych powiatów obszarowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest ubogim powiatem. Chciałabym zapytać, czy przy następnym naborze tego typu jednostki samorządu terytorialnego mają szansę na to, żeby być potraktowane priorytetowo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

To są fakty. Pozwolę sobie z tego miejsca zacytować słowa pani burmistrz Byczyny z ramienia PSL: To wielki dzień dla Byczyny, dla gminy najbardziej zadłużonej w naszym województwie i jednej z najbardziej zadłużonych w Polsce. Jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu na rok 2022 i widzimy, że nie stać nas by było na żadną inwestycję, gdyby nie środki w ramach programu rządowego Polski Ład. Szanowna Opozycjo! Wiele osób zadaje pytanie, jaki ma program Platforma Obywatelska. Pan poseł Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Władysław Kurowski.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Koleżanki i Koledzy! Okręg nr 12 cieszy się z kilkuset milionów złotych. Natomiast ja chciałem wyrazić swoje podziękowanie w imieniu wszystkich samorządowców ziemi myślenickiej, powiatu myślenickiego, bo mnie o to prosili i zobligowali, żeby podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i panu, panie ministrze, za środki w kwocie ponad 100 mln zł dla powiatu myślenickiego. To środki kierowane do samorządów, ale to przede wszystkim środki kierowane do mieszkańców powiatu myślenickiego. Serdecznie dziękujemy i liczymy na więcej w następnym rozdaniu.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przede wszystkim za to, że pieniądze trafiły do wszystkich gmin i były skierowane na te programy, na te zadania, których one wcześniej nie mogły wykonać, bo raz było na drogi takie, raz było na domy kultury, natomiast samorządy same wiedzą, jakie mają potrzeby. Właśnie na te potrzeby, o których samorządy wiedzą najlepiej, te pieniądze zostały skierowane.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na wstępie bardzo dziękuję za trud wykonanej pracy zarówno panu premierowi, jak i panu ministrowi, a także wszystkim osobom, które nadzorowały ten program. Tytaniczna, benedyktyńska praca, która przynosi sukcesy. Te programy to nie propaganda, te programy to konkret, to są działy, które pozwalają myśleć o przyszłości.

W związku z tym, moi drodzy państwo, ta edycja i przyszłe to przyszłość samorządów terytorialnych, to przyszłość naszego narodu, przyszłość społeczeństwa i rozwój tego potencjału. Chcemy, żeby gminy stawały się coraz bardziej samodzielne. Dzięki tym inwestycjom, dzięki temu, że nadgonią te zapóźnienia, będą mogły same realizować ambitniejsze plany w ciągu wieku. Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Do okręgu wyborczego nr 22 południowej części województwa podkarpackiego trafia z tego naboru 860 mln zł na inwestycje, przede wszystkim drogowe, wodno-kanalizacyjne, ale także na budowę farm fotowoltaicznych w gminie Fredropol, kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Birczy, przebudowę budynku szkół w Radymnie, budowę wiejskiego domu kultury w Woli Węgierskiej, gminnego parku selektywnej zbiórki odpadów w Tarnowcu czy parku turystyki i kultury w Skołyszynie. To są znakomite inwestycje oczekiwane przez lokalne społeczności. To jest prawdziwa realizacja zasady zrównoważonego rozwoju.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Opozycja mówi, że te kryteria były niesprawiedliwe, bo nie wszystkie gminy czy powiaty dostały, ale to jest nieprawda, bo wnioski składały gminy i powiaty.

Panie Ministrze! Bardzo serdecznie dziękuję za ten fundusz strategiczny, dziękuję panu premierowi i wszystkim członkom komisji, które się napracowały. W imieniu samorządów proszę, aby dalej było to kontynuowane z korzyścią dla mieszkańców całej Polski. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Tym bardzo dobrym przykładem jest gmina Byczyna rządzona przez świetną burmistrz z Polskiego Stronnictwa Ludowego panią Iwonę Sobanię.

To jest właśnie konkretny przykład, jak rząd Zjednoczonej Prawicy pomaga samorządom.

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo!

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Ministrowie!

Panie ministrze, zwracam się do pana ministra Pawła Szefernakera, wielkie podziękowania od wszystkich za tytaniczną pracę, którą pan [[Oklaski]] wykonał jako przewodniczący komisji, która te wnioski rozpatrywała. Tych wniosków było bardzo dużo. 23 mld zł, które zostały przeznaczone, to są bardzo duże pieniądze. Oczywiście samorządy, mogąc korzystać z dofinansowania nawet 95% inwestycji, te wnioski składały, większość z nich te wnioski składała.

My dopiero nadrabiamy prace przy infrastrukturze np. wodno-kanalizacyjnej. Nie ma wody, nie ma kanalizacji. Dzięki tym środkom to się zmienia. Panie ministrze, kolejny nabór w tym roku, ale czy rozstrzygnięcie też? Bo wszyscy na to czekają. Szanowni Państwo! Za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u były też inwestycje, z dużym opóźnieniem były, i kto je wykonywał? naszych podwykonawców, którzy do dzisiaj walczą z tym, że nie otrzymali zapłaty.

Opozycja krzyczała - niewielu państwa się zapisało do głosu, bo faktycznie, o czym mówić - a wypadałoby powiedzieć: dziękuję, ale tego nie zrobiliście. Mówiliście, że samorządowcy muszą zapłacić, że potem dopiero dostaną jakieś papierowe czeki, z których nic nie wynika. Inwestycje z RFIL są już oddawane. I to nie premier decyduje, to właśnie wasi włodarze składają wnioski, to oni decydują, czy wnioski.

Jestem z powiatu gorlickiego, cały powiat, wszystkie 10 gmin plus powiat otrzymały środki, i to znaczące środki.

Reasumując: krzyczeliście, że teraz jest dobrze, a jak odejdziemy, to będzie źle, więc wniosek jeden: Prawo i Sprawiedliwość musi rządzić dalej, żeby Polska dalej mogła się rozwijać i żeby ludziom żyło się coraz lepiej. Dziękuję, pani poseł. Uprzejmie proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana ministra Pawła Szefernakera. Szanowni Państwo! Jest po czasie, pani nawet nie chce usłyszeć odpowiedzi na pani pytanie, którą przygotowałem. Po co tyle nienawiści, szanowna pani? A jeżeli chodzi o tę nienawiść, które zionęła z państwa strony, to ktoś kiedyś powiedział: nienawiść spowodowała wiele problemów na świecie, ale jeszcze ich nie rozwiązała. A my tym programem rozwiązujemy konkretne problemy, na które to rozwiązania ludzie czekali przez lata.

Jakie ręce? Proszę pana, ja mam czyste ręce. A pan?

Dziękuję za wykonaną pod pańskim kierunkiem pracę komisji rozpatrującej wnioski jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Inwestycji Strategicznych, której efekty spotkały się z uznaniem ogromnej [[Oklaski]] większości samorządowców. Byłem przekonany, że przy jakichkolwiek wątpliwościach państwa będziecie jednak potrafili podejść obiektywnie, ale nie potraficie tego zrobić. My wydajemy 6 mld rocznie. Szanowni Państwo! Spróbuję odpowiedzieć na zdecydowaną większość pytań. Kiedy inwestycje mogą ruszyć? Otóż, szanowni państwo, na początku przyszłego tygodnia będą wystawione promesy Banku Gospodarstwa Krajowego i cała dokumentacja związana z rozpoczęciem przetargów będzie mogła już ruszyć, tak żeby w ciągu pół roku wszystkie przetargi zostały ogłoszone.

Dzięki projektowanym zmianom dochody samorządowe z PIT, CIT i subwencji ogólnej wyniosą w przyszłym roku według prognoz Ministerstwa Finansów 149 mld zł.

Państwo uważają, że nie należy podnieść tej kwoty, bo jeżeli podnosimy kwotę wolną od podatku, państwo uważają, że stracą. Jak się podnosi kwotę wolną, to będą zawsze mniejsze kwoty, które będą wpływały do budżetu państwa i budżetu samorządów, to jest podstawa ekonomii. Naprawdę niedużo trzeba wiedzieć, żeby się w tym zorientować. Pracujemy nad tym, żeby zrekompensować samorządom straty. Tak jak powiedziałem, dzięki algorytmowi, który przyjęliśmy w ustawie, za którą głosowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość - dziękuję większości parlamentarnej, że to poparła - ta ogólna subwencja rozwojowa będzie mogła być wydawana w ramach dochodów własnych samorządów. Tak jak powtarzam, jeżeli chodzi o dochody samorządowe z PIT, CIT i subwencji ogólnej, to wyniosą one więcej niż w tym roku według prognoz Ministerstwa Finansów. Szanowni Państwo! Państwo pytali, dlaczego tylko 35 mln dla Bydgoszczy. Zrealizowane zostały dwa wnioski dla Bydgoszczy, trzeci wniosek był na kwotę 425 mln. Największy wniosek to było 160 mln dla województwa małopolskiego. Jeden z panów posłów rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia: ten wasz Polski Ład. Szanowni państwo, tak, nasz Polski Ład, my się go nie wstydzimy, jesteśmy dumni, [[Oklaski]] a jeżeli wy macie jakieś inne łady czy wstydzicie się tego, że on jest polski, to już wasz problem.

Jestem przekonany, że wtedy Rybnik otrzyma środki. Pieniądze tam po prostu nie dotrą. Za waszych rządów byłoby to niemożliwe. Szanowni Państwo! Szanowni państwo, pokażcie mi samorządowca, który płaci z góry za wykonanie roboty. Płaci się albo w transzach, albo na końcu. To jest matematyka.

Kto komu płaci z góry za wykonaną robotę? Szanowni Państwo! Program dla terenów popegeerowskich będzie kontynuowany także w ramach inwestycji sportowych. Inwestycje sportowe będą w dalszym ciągu realizowane na terenach popegeerowskich. Żaden taki wniosek w Polsce w tym rozdaniu nie został rozstrzygnięty.

Szanowni Państwo!

Inne gminy również muszą je otrzymać. Będziemy namawiać gminę do tego, żeby w kolejnym naborze te wnioski były mniejsze. Będziemy chcieli realizować Polski Ład razem z takimi gminami jak gmina Przecław i gmina Wieluń. Szanowni Państwo!

Już teraz można było je składać. To był IV priorytet, 20% wkładu własnego. Nadal będzie można składać wnioski na inwestycje związane z światłowodami. Szanowni Państwo! Postarałem się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. W ostatnim zdaniu chciałbym powiedzieć, że państwo bardzo często mówili, jak wspaniale było za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Pan Andrzej Porawski odpowiedział: Mnie najtrudniej było z rządem Donalda Tuska, który deklarował prosamorządowość, ale jej nie realizował. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1661 i 1669) Uprzejmie proszę pana posła Zbigniewa Babalskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 1661. Marszałek Sejmu, na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierowała w dniu 13 października 2021 r. powyższy projekt uchwały do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych do pierwszego czytania. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm przyjąć raczył projekt uchwały z druku nr 1661 bez poprawek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Kazimierz Smoliński. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu wobec zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zawartej w druku nr 1661. Jako klub pozytywnie opiniujemy i będziemy popierali ten projekt, bardzo krótki, zawierający upoważnienie dla Prezydium Sejmu do określenia zasad i sposobu doręczania posłom uchwał oraz powiadomień o zarządzeniach, o których mowa w przepisach rozdziału, w którym znajduje się art. 25a.

Tak jak w innych przypadkach będzie to możliwe poprzez pocztę elektroniczną. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicja Obywatelska wobec projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druki nr 1661 i 1669. Regulamin Sejmu powinien być jasny i czytelny oraz nie budzić wątpliwości. Projekt uchwały zakłada, że Prezydium Sejmu ma określić zasady i sposób doręczania posłom uchwał i zarządzeń, które dotyczą obniżenia diety parlamentarnej lub uposażenia poselskiego. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych uregulowań w tym zakresie, co stanowi problem natury praktycznej. Po zmianie regulaminu to Prezydium Sejmu będzie miało delegację do określenia tego, jak danemu posłowi zostanie doręczona uchwała lub zarządzenie o obniżeniu diety lub uposażenia. Pan poseł Marek Rutka w imieniu klubu Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wniesiony projekt uchwały dotyczący zasad i sposobu doręczania posłom uchwał i zarządzeń w sprawie obniżenia uposażenia poselskiego pewnie nie byłby rozpatrywany, gdyby nie specyficzny sposób bycia jednego z posłów, znanego z negowania istnienia pandemii COVID-19. Ze zrozumiałych względów nie przytaczam nazwiska owego posła, aby nie propagować jego postaci. Warto jednak przybliżyć szczegóły sprawy, która stała się bezpośrednią przyczyną proponowanej zmiany w regulaminie Sejmu. Wobec posła znanego z umiłowania do monarchii i popierającego pomysł formalnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski zastosowano najsurowszą z możliwych kar finansowych zawartych w art. 25 regulaminu Sejmu. Oczywiście powodem zastosowania kary nie były osobliwe poglądy pana posła, a słowa skierowane podczas obrad plenarnych Sejmu w stronę ministra zdrowia, cytuję: Będziesz pan wisiał. Każda kara, w tym również kara finansowa, powinna spowodować pożądaną zmianę zachowania. Co istotne, na jednym z portali zajmujących się zbiórkami pieniężnymi prowadzona jest zbiórka, której celem jest wsparcie działalności owego posła. Nie ma co ukrywać, że prowadzona zbiórka ma związek z karą finansową nałożoną na pana posła. Na dziś na godz. 11.45 na koncie zbiórki znajdowało się 419 626 zł. Zebrana kwota wielokrotnie przekracza łączną sumę kary nałożonej na pana posła zgodnie z art. 25 regulaminu Sejmu. Przytoczony przykład podaję, aby ukazać, że nałożona kara finansowa w żaden sposób nie spełniła swojego zadania.

Dziękuję. Pan poseł Jan Łopata, Koalicja Polska. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska mam zaszczyt zaprezentować stanowisko w sprawie omawianej w tym punkcie obrad. Jak już wielokrotnie padało z tej mównicy, celem proponowanej zmiany jest dodanie w dziale I w rozdziale 4 przepisu, który będzie stanowił podstawę do określenia przez Prezydium Sejmu sposobu doręczania posłom uchwał i zarządzeń dotyczących obniżenia uposażenia poselskiego lub diety parlamentarnej.

Wydaje się, że te techniczne w sumie zmiany, bez potrzeby przywoływania konkretnego przypadku, tylko dla usprawnienia komunikacji, są dobre. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Artur Dziambor w imieniu koła Konfederacja. Wysoka Izbo! Na początek krótki komentarz do tej ustawy.

Grzegorz Braun, który przez to, że trzymał się pryncypialnie zasad i trzymał się pryncypialnie prawa do wykonywania mandatu poselskiego w taki sposób, jaki uważa za wolny, był wielokrotnie wypraszany z tej sali i karany finansowo przez marszałka Zgorzelskiego, marszałka Czarzastego, przez marszałek Witek wielokrotnie. Ale to się dobrze skończy dla pani, bo ostatecznie nie będzie pani później w przyszłości odpowiedzialna. Mamy tutaj ekspertyzy prawne o bezprawności nakazu noszenia maseczek przez posłów. Jedna z nich jest napisana przez prof. Marka Chmaja, a druga z nich jest napisana przez panią prof. Sabinę Grabowską, która tę analizę wykonała dla Biura Analiz Sejmowych. Obie te analizy jednoznacznie stwierdzają, że ograniczanie mandatu posła i wypraszanie posła z sali dlatego, że nie założył maseczki zgodnie z waszym widzimisię, było bezprawne. Bezprawne było również odbieranie mu uposażenia, ponieważ wbrew temu, co wy opowiadacie, to nie jest tak, że dotychczas Grzegorz Braun migał się od odpowiedzialności. Nie było żadnego migania się od odpowiedzialności. Pieniądze, które mu zabierało Prezydium Sejmu, były pobierane z jego wypłaty przez ostatni ponad rok. To znaczy, że nie Grzegorz Braun, tylko jego rodzina była brana na zakładnika Prezydium Sejmu przez to, że odbierane były mu pieniądze, dzięki którym tę rodzinę może utrzymywać. Te pieniądze były od niego zabierane, a teraz jeszcze otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary finansowej, co spowodowało, że trzeba było uruchomić zbiórkę na to, żeby mógł normalnie dalej funkcjonować. Szanowni Państwo! W przyszłości trzeba się będzie oczywiście poważnie zastanowić nad tym, czy Prezydium Sejmu, czy marszałek Sejmu, czy ktokolwiek ma prawo wymierzać kary finansowe posłom za to, że zachowują się albo mówią coś, z czym nie zgadza się większość parlamentarna, ponieważ ta większość parlamentarna, którą wszyscy państwo od lewa do prawa, a właściwie lewa, lewa, centrum stworzyliście, ta sytuacja doprowadziła do tego, że dzisiaj musimy dokonywać takich absurdalnych zmian. Niestety, szanowni państwo, przekroczyliście swoje uprawnienia, te ekspertyzy mówią o tym jasno. Proszę bardzo, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Wysoki Sejmie! Tak, to jest epokowe wyzwanie, jak usprawnić proces doręczania posłom zawiadomień o obniżeniu poborów. Przypomnę tylko, że dzieje się to w Sejmie, którego regulamin w ogóle nie widzi dokumentów cyfrowych. Przypomnę, że ma to miejsce w Sejmie, gdzie elektroniczne pisma przesyłane przez ministrów są drukowane na papierze i w tej formie doręczane posłom - na kartkach. Dzieje się to w Izbie, w której marszałek wbrew regulaminowi dopuszcza na mównicę osobę niedysponującą mandatem poselskim, żeby mogła głosić swoje homofobiczne frazesy i epatować mową nienawiści, a jednocześnie nic zdrożnego nie widzi w tym, żeby czas wypowiedzi posłów w debacie ograniczyć do 30 sekund. Następnym razem proponuję może 15 sekund albo 7 sekund. Dzieje się to w Izbie, w której można ogłosić reasumpcję przegranego głosowania i naściemniać posłankom i posłom, że się zasięgnęło w tej sprawie opinii pięciu prawników. Tak, zdecydowanie usprawnienie procesu doręczania posłom zawiadomień o obniżeniu uposażeń jest bardzo ważnym wyzwaniem. Posłanki i posłowie ruchu Polska 2050 oczywiście poprą to rozwiązanie. Przechodzimy do pytań. Zamykam listę osób chcących zadać pytanie. Zapisało się sześciu parlamentarzystów. Bardzo proszę jeszcze, po dopisaniu się pana. Wyznaczam czas na zadanie pytania - pół minuty. Wysoka Izbo! Mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem przesłanki, jakie powodowały autorami tego projektu podczas jego pisania. Mniemam, że szanowne Prezydium, pewnie podobnie jak pan premier, szykuje się na wojnę i w związku z tym stara się nadać swoim działaniom bardziej formalnego charakteru.

Pan poseł Jakub Kulesza, koło Konfederacja.

Wysoka Izbo! Nie potrzebujecie tej uchwały, zmiany regulaminu Sejmu, by brać za zakładników rodziny posłów, ograniczać im mandat poselski, wykluczać ich z porządku obrad. Dzisiaj już nikt nie ma tej maseczki, pomimo że mamy rzekomo czwartą falę.

Jak sama nazwa wskazuje, to jest posłaniec wysłany przez wyborców, powinien być nietykalny dla swoich kolegów. Jest niedopuszczalne, żeby koledzy z jego ław recenzowali jego wypowiedzi i karali go finansowo.

Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Osobiście nie popieram sytuacji, w której karze się posła za to, że powiedział coś do innego lub, nie wiem, nie założył maseczki. Jeśli inny poseł się obraził, to są sądy powszechne, powinni się pozwać i tam załatwiać sprawę. Ale ja w innej sprawie.

Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! A ja dziękuję za tę uchwałę, bo jeśli nie można inaczej, to można po prostu tak.

Chciałabym, żeby poseł Braun, kiedy pojawia się na posiedzeniach komisji, pracował faktycznie merytorycznie, tak jak mówili, bronili go tutaj koledzy hipokryci, którzy pewnie się zaszczepili, ale po prostu o tym nie mówią, bo mogliby zapłacić za to polityczną cenę. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

I nawet mandat poselski musi się podporządkować tym zasadom.

Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Mam bardzo krótkie pytanie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1631) Uprzejmie proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Macieja Miłkowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Posłowie! Jest mi niezmiernie miło przedstawić państwu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem tej ustawy jest stworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ma to na celu skoncentrowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej. Planowane jest połączenie aktualnie dwóch instytucji podległych ministrowi zdrowia: Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skupienie działań w tym podmiocie pozwoli na połączenie tematyki uzależnień behawioralnych i uzależniających substancji psychoaktywnych na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie edukacji, profilaktyki, szkolenia kadr, leczenia, rehabilitacji i działalności badawczej. Obecnie te dwie instytucje realizują zadania ustawowe zbliżone w swoim zakresie i zadania Narodowego Programu Zdrowia związane z odrębnymi rodzajami uzależnień, mimo że jest uzasadnione w wielu zakresach połączenie tych zadań w odniesieniu do profilaktyki i rozwiązywania problemów w ogóle związanymi z uzależnieniami czy monitorowania realizacji polityki państwa w zakresie uzależnień. Centrum będzie działało w sposób skoordynowany i spójny, co przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania problemami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych, wpisującymi się w zagrożenia dla zdrowia publicznego. Powstanie jedna instytucja, która w imieniu ministra zdrowia będzie odpowiadała za cały ten sektor.

Tak że to jest głównym celem połączenia tych dwóch jednostek w jedną. Drugi element zmiany dotyczy ustanowienia gminnych programów w obszarze profilaktyki uzależnień, chodzi o to, żeby scalić działania w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej, ponieważ w bardzo wielu podmiotach, w bardzo wielu samorządach gminnych te dwa zadania są realizowane w ramach jednej strategii.

Planujemy włączenie tego systemu kształcenia do systemu szkoleń określonego w ustawie o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Będzie to skutkowało tym, że będziemy mieli jednolity system kształcenia, jednolite umiejętności poszczególnych specjalistów. Aktualnie istnieją trzy ścieżki uzyskiwania certyfikatu. Dwie ścieżki są obsługiwane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, jedna ścieżka jest obsługiwana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak że wszyscy będą kończyli ten sam cykl specjalizacyjny w zakresie psychoterapii uzależnień. Ujednolicamy w tym zakresie standardy treści kształcenia i sposób realizacji, co przyczyni się na pewno do podniesienia jakości kształcenia. Jednocześnie te przepisy zakładają uznanie równoważności certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień z dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ta rada, tak jak do tej pory, będzie zajmowała się monitorowaniem i koordynowaniem działań w zakresie realizacji polityki państwa w obszarze uzależnień i zaleceniami rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym uzależnień. Projekt przewiduje okresy przejściowe tego połączenia.

Koszty te będą realizowane w ramach aktualnych kosztów tych dwóch jednostek. Tak że organizacyjnie dla Ministerstwa Zdrowia w przypadku całego zakresu to połączenie będzie uzasadnione. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Katarzyna Sójka. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1631. Projektowana ustawa wprowadza zmiany głównie w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Proponowane zmiany mają na celu utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projektowane zmiany mają na celu skupienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z różnymi rodzajami uzależnień w jednej jednostce organizacyjnej jako państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Skoncentrowanie działań w jednym podmiocie decyzyjnym, jakim będzie centrum, pozwoli na połączenie tematyki różnych uzależnień czynnościowych i chemicznych, uzależnień od substancji legalnych i od substancji nielegalnych, na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Obecnie funkcjonujące jednostki działają osobno w odniesieniu do problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z pominięciem innych uzależnień, które w tym zakresie pozostają poza regulacjami prawa powszechnie obowiązującego. Aktualnie każda z tych jednostek realizuje swoje zadania ustawowe i zadania Narodowego Programu Zdrowia związane z odrębnymi rodzajami uzależnień, mimo że w wielu przypadkach ich połączenie byłoby zasadne i korzystne, ponieważ oba podmioty realizują zadania o zbliżonym zakresie przedmiotowym. Zadania podmiotów odnoszą się wspólnie do profilaktyki, do leczenia uzależnień, do edukacji publicznej oraz wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji przez nie ustawowych zadań dotyczących odpowiednio profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Czynnikiem różnicującym zakres zadań obu tych podmiotów nie są obszary problemowe czy formy oddziaływania społecznego, a jedynie podział na substancje, których używanie powoduje szkody i problemy społeczne. Centrum zajmujące się w sposób kompleksowy problematyką uzależnień umożliwi prowadzenie polityki państwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w sposób skoordynowany i spójny, co przyczyni się do bardziej skutecznego niż dotychczas osiągania planowanych celów. Wprowadzenie proponowanych zmian zwiększy efektywność działań, zmniejszy obciążenia administracyjne, pozwoli na poprawę obecnie funkcjonującego rozwiązania organizacyjnego i lepsze wykorzystanie środków z budżetu państwa, a przede wszystkim poprawi efektywność prowadzonych działań i zadań. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Rajmund Miller w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1631. Projekt ustawy wprowadza połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku tego utworzone zostanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Celem powołania centrum jest skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej jako państwowej jednostce budżetowej, utworzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W miejsce Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powołana zostanie Rada do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zakładane są również zmiany w zakresie ustanawiania wojewódzkich i gminnych programów w obszarze profilaktyki uzależnień. Projekt oddziałuje na następujące podmioty: na Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i na Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na populację osób uzależnionych i współuzależnionych, na jednostki samorządu terytorialnego i na organizacje pozarządowe. Wysłuchałem dokładnie pana ministra. Mamy trochę zastrzeżeń do zapisów tej ustawy. Uważamy, że pominięto w tym zapisie prawa osób pozostających w procesie kształcenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień czy instruktora terapii uzależnień, prowadzonego na dotychczasowych zasadach, oraz osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień, do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin. Obecnie osoby te stanowią ponad 50% świadczeniodawców zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnień. Praca z pacjentami uzależnionymi, członkami ich rodzin warunkuje możliwość uzyskania certyfikatu specjalisty czy instruktora na bazie dotychczasowych przepisów lub możliwość podjęcia kształcenia specjalistycznego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. W takim razie musimy uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki akt prawny będzie gwarantował dalszy dostęp tych osób do pacjentów.

Jest tu jeszcze kilka innych zapisów. Mamy również wątpliwości co do tego, że nastąpi upolitycznienie nowo tworzonego ciała, ponieważ to pan premier będzie miał decydujące zdanie, kto w skład tego ciała wejdzie. Trzeba zaznaczyć, że trochę inny jest profil i sposób działania agencji do spraw narkomanii, która zajmuje się ok. 60 tys. przypadków w Polsce.

Jeżeli ci ludzie nie znajdą się w odpowiednim, powiedzmy, składzie tej rady, to uważamy, że będzie istniało zagrożenie dla funkcjonowania działań w zakresie uzależnień od alkoholu. Oczywiście proponujemy dalszą pracę nad tą ustawą. Będziemy prosić o rozważenie naszych poprawek, które do tej ustawy wniesiemy. Dziękuję, panie pośle. W imieniu klubu Lewica głos zabierze pan poseł Zdzisław Wolski. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałoby się powiedzieć: wreszcie. Projekt ustawy powinien być uchwalony przez Sejm, Senat, pana prezydenta już lata temu, a już na pewno powinno to się zacząć w roku 2019, a ci, którzy bliżej się interesują, wiedzą dlaczego. Wreszcie jest akt porządkujący dotychczasową rozproszoną walkę z uzależnieniami, przede wszystkim prowadzoną przez PARP-ę, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Pan poseł Miller o tym mówił, o alkoholu.

Jest ok. 6 mln osób, których to dotyka wprost, łącznie z osobami współuzależnionymi, czyli przede wszystkim rodzinami i bliskimi.

Jest to przecież problem o olbrzymim znaczeniu społecznym, również ludzkim.

Będzie zajmowało się m.in. nie tylko tzw. psychotropami, ale i nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi, czyli tzw. dopalaczami, przy okazji, to już pan minister mówił.

Umożliwi lepszą koordynację działań, jako że, tak jak mówiłem, one się wzajemnie przenikają. Oczywiście oby tylko były prawidłowo realizowane i wdrażane. Wiele wątpliwości technicznych czy innych w Komisji Zdrowia na kolejnych etapach będziemy omawiali. Dziękuję. Zgodnie z art. 1 pkt 8 projektu ustawy członków Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów. W skład tej rady będą wchodzili: jako przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, a poza tym jeszcze 12 reprezentantów w randze ministra bądź wiceministra z poszczególnych resortów. Natomiast przedstawiciel strony samorządowej to będzie tylko jedna osoba. Wobec tego, że w zakresie wdrożenia tej ustawy dużo zależeć będzie od działalności strony samorządowej, wydaje się, że skład tej rady jest głęboko nierównoważny, jeśli idzie o kwestię dotyczącą reprezentacji strony samorządowej.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt rządowy jest teoretycznie prosty i jasny. Dotyczy utworzenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z pierwszych spostrzeżeń jest to, że w projekcie aż roi się od słów „koncentracja”, „centrum” i innych synonimów słowa „centralizacja” W projekcie ustawy zaproponowano zmiany w zakresie ustanawiania wojewódzkich i gminnych programów w obszarze profilaktyki uzależnień. Autorzy ustawy wskazują, że istotnym źródłem polityki scalenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej są także działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza na poziomie gminnym. Uważam, że rząd niepotrzebnie wtrąca się w sprawy lokalnej i regionalnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom, zamiast skupić się na koordynacji działań wespół z resortami, ministerstwami, które odpowiadają za edukację, naukę, sport czy oczywiście zdrowie. Tutaj jest klucz do właściwej krajowej polityki przeciwdziałania uzależnieniom, a nie ingerowanie w szczegółowe, ukierunkowane na charakterystykę danej społeczności lokalnej i regionalnej, polityki profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. To, co jest ważne z punktu widzenia nowej instytucji w relacjach z gminami i województwami, to odpowiedni i sprawny system raportowania i przekazywania właściwych danych, wyników i wniosków z wdrażanych strategii, które powinny służyć jako przedmiot w kształtowaniu polityki krajowej względem problemu uzależnień. Kolejna sprawa to cel tego nadzoru nad ustanawianiem wojewódzkich, a w szczególności gminnych programów. Czy czasem w odpowiednich nowych rozporządzeniach do ustawy nie znajdą się przepisy ingerujące dalej, w kolejne przepisy, np. dotyczące koncesji i związanych z tym opłat? Uważam, że trudno wskazać, żeby połączenie ww. instytucji stworzyło także nowe obowiązki dla nowej instytucji, bo chyba nie należy do nich na siłę wpisane do ustawy tzw. budowanie systemu monitorowania problemów alkoholowych występujących na terenie Polski. Za stworzeniem nowej instytucji powinno iść w mojej opinii stworzenie nowej jakości, nowych sposobów radzenia sobie z problemami, nowych mechanizmów oraz instrumentów, a przede wszystkim wspieranie lokalnych i regionalnych odpowiedników. A co mamy? W moim przekonaniu bezwiedne, administracyjne połączenie dwóch instytucji. Mankamentem w procedowaniu nad rządowym projektem jest kolejny raz brak prekonsultacji. Jak ważnym elementem są prekonsultacje procesu legislacyjnego, wskazuje choćby raport z obowiązkowych konsultacji, gdzie uwzględniono np. uwagi Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, które wskazywało na chaotycznie wymienione zadania centrum - pod kątem ich zakresu, poziomu szczegółowości, kolejności, powtarzalności - w których całkowicie pominięto zadania związane np. z: pomocą osobom dorosłym, rodzinom, członkom rodzin, partnerom osób uzależnionych; kontynuowaniem do 2024 r. systemu kształcenia specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień dotychczas realizowanego osobno w PARPA i w krajowym biurze; brakiem regulacji dotyczących ścieżki przygotowania i certyfikowania superwizorów w dziedzinie psychoterapii uzależnień; brakiem regulacji dotyczących stałych kadencyjnych ciał merytorycznych, eksperckich przy krajowym centrum - doradczych i opiniujących szkolenia i projekty; brakiem powołania komisji odpowiedzialności zawodowej.

Pytanie jest takie: Czy po połączeniu PARPA i krajowego biura będzie można śmiało stwierdzić, że nowa instytucja będzie lepsza, sprawniejsza i silniejsza niż działające osobno biuro i agencja? W uzasadnieniu argumentów jest bardzo mało, natomiast wcale nie ma argumentów, że efekt działań nie ulegnie pogorszeniu, a o tym także - uważam - autorzy tego projektu powinni jasno powiedzieć. Pytania, które mam, zadam w serii pytań. Pan poseł Grzegorz Braun w imieniu koła Konfederacja.

Tutaj, w Wysokiej Izbie, jak zwykle najpierw tworzy się problemy, żeby potem je rozwiązywać, najlepiej administracyjnie tworząc jakieś superministerstwa, superresorty, nowe instytucje. Tu oczywiście trendem, z naszego punktu widzenia może nawet obiecującym, jest jakaś komasacja, że z dwóch szyldów robi się jeden. Ale z drugiej strony nasza niewiara w instytucjonalne rozwiązywanie problemów jest tak daleko posunięta, że musimy być sceptyczni wobec projektu jako całości, zwłaszcza że występujecie z tym projektem najbezczelniej po 1,5, ach, już prawie 2 latach wpędzania Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych, w uzależnienia. Polityka walki z mniemaną pandemią doprowadziła, szanowni państwo, powie wam to każdy terapeuta, pediatra, psychiatra, do wzniesienia fali depresji, nerwic, ach, także problemów społecznych - wzrost liczby zamachów samobójczych wśród nieletnich o 1/3. Zaprzestańcie działań, które generują choroby, nieszczęście, tragedie i patologie. Przestańcie szkodzić, a może wtedy nie będziemy musieli wszyscy tyle pomagać. Weźmiemy ten projekt na warsztat, zaproponujemy do niego nawet przynajmniej jedną poprawkę. Skoro w pierwszym punkcie mowa o kreowaniu postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych oraz zapobieganiu uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, to - wiecie państwo - może po prostu załączymy jako poprawkę społeczny projekt: Stop LGBT plus, który tutaj późnym wieczorem wczoraj był procedowany, właśnie dlatego, że ludzi, którzy popadli w kłopoty na tle uzależnień behawioralnych, trzeba traktować z należytą troską. Trzeba im przyjść z pomocą, trzeba umożliwić im leczenie, zamiast promować ich schorzenia. A zatem (Dzwonek) dobry sposób na to, żeby projekt: Stop LGBTQ itd., plus był jednak procedowany. Pan poseł Wojciech Maksymowicz w imieniu koła Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zagadnienie uzależnienia jest oczywiście bardzo złożone i same instytucje rządowe czy też samorządowe na pewno nie załatwią tego problemu, konieczne jest wspólne działanie, praktycznie całego społeczeństwa.

Projekt zakładający utworzenie jednego krajowego centrum w wyniku połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma zwiększyć efektywność działań realizowanych przez oba podmioty. Dodatkowo nowa instytucja ma zająć się wszelkimi innymi typami uzależnień. Również gminne i wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki uzależnień mają być scalane. To na pewno może pomóc realizować gminne programy samorządowe, bo przecież problem dotyczy też obszarów jak najbliższych mieszkańcom i społeczności.

A jedna z uwag, która się nasuwa przy analizie propozycji projektu, powinna być dyskutowana w komisji. Mianowicie chodzi o jednego przedstawiciela obecnego ministra edukacji i nauki w Radzie do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Nie wiadomo też, czy w przyszłości nie będzie podjęta decyzja o kolejnym przyporządkowaniu tych działów do dwóch ministerstw. Edukacja na poziomie szkolnym, przedszkolnym na pewno ma inną specyfikę i powinna być bardzo wyraźnie brana pod uwagę, tak samo jak i inna jest specyfika szkolnictwa wyższego. Dziękuję bardzo. Popieramy przekazanie do dalszych prac. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu koła Polskie Sprawy pan poseł Andrzej Sośnierz. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Konstrukcja prawidłowa, sam pomysł wydaje się słuszny. Teoretycznie. Ale chcę zwrócić uwagę, że wiele teoretycznie dobrych pomysłów wcale potem w praktyce nie funkcjonuje. I dziwię się, że Lewica też popiera ten projekt, bo w lewicowym myśleniu zawsze jest takie założenie, że jak stworzymy instytucję państwową, centralną, to będzie dobrze.

Ale czy będzie lepiej? Zauważyłem, że najczęściej nieumiejętność koordynowania różnych podmiotów przez kogoś zarządzającego - w tym przypadku państwo, rząd - zastępuje się centralizacją.

Nie, to jest pogłębiający się upadek tej instytucji. Czy sanepid scentralizowany tak niedawno działa lepiej niż poprzednio? Nie. Więc z zainteresowaniem będziemy słuchali, jakie argumenty przekonały, że po raz kolejny pomysł centralizacyjny tym razem się uda. Bo, jeszcze raz podkreślam, one się ciągle wydają słuszne i cały świat wraca co chwilę do takich rozwiązań socjalistycznych. Czy tylko są takie intencje? Z zainteresowaniem przeczytałem kryteria, które ma spełnić przyszły dyrektor tego centrum, i okazuje się, że właściwie on niewielkimi osiągnięciami musi się wykazać, poza takim enigmatycznym zdaniem, że musi wiedzieć, czym kieruje. Tak jest tam napisane: że musi posiadać wiedzę. Ale jak to? Przecież każdy z nas ma jakąś wiedzę o narkomanii i każdy z nas coś wie o alkoholu, więc takie miękkie kryterium być może jest przygotowane dla kogoś, kto nie będzie w ogóle nic albo niewiele wiedział.

Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuje Ministerstwu Zdrowia za przygotowanie tego projektu, ponieważ te nowe rozwiązania znacznie ułatwią wspieranie osób, które borykają się z uzależnieniami. Do tej pory te dwie instytucje prowadziły niezależną działalność związaną z profilaktyką uzależnień od alkoholu oraz profilaktyką uzależnień od innych substancji, w tym narkotyków. Wiemy, że obecnie uzależnienia bardzo często są krzyżowe. Bardzo rzadko spotyka się u pacjentów wprost uzależnienie od jednej substancji. Bardzo często jest tak, że jeżeli jesteśmy uzależnieni od alkoholu, to równocześnie też występuje uzależnienie od leków czy innych substancji. W tej chwili ta koncentracja sił i środków, możliwości, także potencjału (Dzwonek) intelektualnego na pewno będzie sprzyjała lepszej realizacji tych zadań. To uprości też funkcjonowanie samorządom, ponieważ.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście pytanie będzie dotyczyło tej nowej instytucji, która ma powstać przez połączenie dwóch istniejących, w tym jednej bardzo doświadczonej w realizacji programów antyalkoholowych. Czy mamy, panie ministrze, dokładne prognozy, jakie będą koszty funkcjonowania tej instytucji w kolejnych latach, w szczególności jeśli chodzi o nabór pracowników, o kwestie organizacyjne, finansowe? Chciałbym również upewnić się, czy zostanie wykorzystany cały potencjał ludzki istniejącej państwowej agencji w nowej instytucji.

Bardzo bym prosił, aby pan minister odpowiedział mi na piśmie, jaki jest rzeczywisty cel dublowania instytucji zajmujących się bliźniaczymi tematami. Czy pieniądze z budżetu będą wydatkowane na prace w terenie, czy tylko na tworzenie kolejnej scentralizowanej jednostki, której głównym zadaniem ma być organizowanie pracy jednostkom terenowym, które do tej pory świetnie sobie radzą bez tworzenia tej czapy rodem ze zjednoczenia? Uprzejmie proszę też o informację, w jaki sposób potencjał jednostek, które podlegają połączeniu, zostanie wykorzystany w nowej jednostce. Raz jeszcze uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska, i zapowiedziane pytania. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Można oczywiście tworzyć kolejne instytucje, sytuować je w zasięgu władzy centralnej, tylko pytanie, czy to będzie efektywne. Czy nie lepiej iść w stronę wykorzystania potencjału instytucji, potencjału ludzkiego, który już dzisiaj istnieje? Powiem szczerze, że ze zdumieniem obserwuję kolejne pomysły Ministerstwa Edukacji Narodowej zarządzanego przez już osławionego - myślę, że nie tylko w Polsce - pana ministra Czarnka, który forsuje różnego typu ideologiczne ofensywy. Natomiast tam jest dzisiaj naturalna przestrzeń do tego, żeby rozpocząć w najmłodszym wieku wśród młodzieży profilaktykę antyuzależnieniową i na to zwracać uwagę. Chciałem zapytać, czy rozważano, aby właśnie na bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dzwonek) usytuować tego typu materię. Pan poseł Jakub Kulesza, koło Konfederacja. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Łączycie dwie instytucje w jedną, ale te instytucje po prostu należy zlikwidować, dlatego że w tych instytucjach, tak jak PARPA, panuje XX-wieczny przesąd, że prohibicją narkotykową, alkoholową można rozwiązać problemy uzależnień. Otóż nie można, wręcz przeciwnie.

Takie są fakty. Tak wygląda współczynnik przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych (Dzwonek) na 100 tys. mieszkańców. To nie działa. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Otóż przewiduje się, że do tej rady będą delegowani przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędach wielu ministrów, czyli mają to być jednym słowem urzędnicy. Pytanie, dlaczego ta rada została tak pomyślana, tak skonstruowana. Wydaje się, że urzędnicy wiele mogą radzić, natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiste pomysły i rzeczywistą sprawczość, to raczej jest ona w rękach tych, którzy mają doświadczenie, i kolokwialnie mówiąc, zjedli zęby na pomocy takim osobom. Dlaczego jest taka systematyka, że będą to urzędnicy, a nie ludzie kompetentni, którzy znają się na rzeczy, którzy rozumieją ten świat i rzeczywiście mogliby pomóc, tworząc takie pomysły i takie wzorce, które (Dzwonek) skutkowałyby pozytywnie? Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wspominał pan, że ok. połowa jednostek samorządowych prowadzi w zasadzie z tymi samymi ludźmi dwa oddzielne programy. Jeżeli chodzi o skutki, to skutki bardziej się różnią niż przyczyny. Czy to połączenie, panie ministrze, przyczyni się do lepszego zwalczania przyczyn powstawania wszelkiego rodzaju uzależnień, zarówno alkoholowych, narkotykowych, dopalaczowych, jak i wszelkich innych, które w coraz większym stopniu wyrównują się między dużymi miastami a małymi gminami? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Nie ma pana posła. Pan poseł Zdzisław Wolski, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Lewica nie popiera centralizacji i zjawiska jedynie słusznych decyzji z fotela ministerialnego. Ten projekt popiera tylko dlatego, że na poziomie gmin, stowarzyszeń rozproszenie, alkoholizm, narkomania, behawioralne uzależnienie itd. wreszcie zostaną scalone. Ale przechodzę do pytań. Art. 10 i 11 o uzyskiwaniu kwalifikacji. Art. 10 zrównuje certyfikat specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień z dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty, czyli są to dokumenty równoważne.

Czy osoby w trakcie (Dzwonek) specjalizacji mogą pracować przy pacjencie, czyli udzielać świadczeń? Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W marcu 2018 r. w województwie łódzkim zbudowaliśmy regionalne centrum diagnozy i terapii FASD dla dzieci i dla opiekunów, rodziców. To jest działanie fakultatywne dla samorządu województwa, nieobowiązkowe, ale mimo to stworzyliśmy przy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej tego typu ośrodek, który do dzisiaj cieszy się dużym zainteresowaniem, wielu osobom pomaga. To jest pytanie do ministerstwa.

Bo widzimy, jak wielki to jest niestety ciągle problem w polskim społeczeństwie. Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom to bardzo rozsądny krok i kierunek, jednakże chciałem zapytać, panie ministrze, jak wygląda to na dole, w Polsce powiatowej. Czy dzieci i młodzież mają tam taki sam dostęp do programów profilaktycznych, jak młodzież i dzieci z większych ośrodków? Mówił pan tutaj o tym, że ta ustawa będzie regulowała również zapisy dotyczące psychoterapeutów uzależnień.

Chciałem zapytać w tym kontekście o regulacje dotyczące zawodu psychologa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Dość niezrozumiały jest dla mnie skład rady. Dlaczego w radzie znalazło się tylko jedno miejsce dla przedstawiciela samorządów i zabrakło miejsca dla specjalistów do spraw leczenia uzależnień? Wynika z tego, że rada będzie ciałem głównie politycznym, a merytorycznym nie bardzo. Ale tak naprawdę bardziej interesuje mnie to, czy ta centralizacja rzeczywiście poprawi sytuację osób uzależnionych, czy poprawi sytuację rodzin, które doświadczają przemocy.

Czy rodziny i dzieci osób uzależnionych będą miały dostęp do opieki psychologicznej i wsparcia? Bo tego cały czas brakuje.

Kiedy wreszcie ministerstwo się tym zajmie i kiedy wreszcie będzie to sytuacja normalna, kiedy osoba uzależniona będzie leczona, a rodzina dzięki temu nie będzie cierpiała? Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Problem alkoholizmu i narkomanii to rzeczywiście poważny temat, przyczyna dramatu wielu osób, wielu rodzin, dlatego chciałbym zadać konkretne pytania. Jakie są plany rządu dotyczące zwiększenia ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi? Sama centralizacja i łączenie instytucji niczego nie rozwiążą. Czy rząd dysponuje danymi dotyczącymi tego, jaka jest skala problemu, jaka jest dynamika, wzrost, spadek, liczby uzależnień? Jak wygląda współpraca w tym zakresie, przede wszystkim z resortem edukacji, ale także z ministerstwem spraw wewnętrznych? Czy planowana jest zmiana możliwości finansowania niektórych zadań w tym zakresie? Wreszcie czy rząd posiada badania dotyczące relacji pomiędzy ochroną zdrowia psychicznego a problemem alkoholizmu i narkomanii? Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dlaczego upolityczniacie ten organ? W zakresie psychoterapii nie ma rozwiązań. Zapomnieliście o tym? Mam pytanie: Czy zgodnie z zapowiedziami osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień i osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień udzielające świadczeń medycznych w tym zakresie wykonują zawód medyczny? Jak to jest? Ustalacie gminne i wojewódzkie programy rozwiązywania problemów alkoholowych. Jakie są zastrzeżenia co do tych komisji, skoro powołujecie nową instytucję? W mojej ocenie zbędne jest tworzenie nowej instytucji. Ostatnie pytanie zada pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Będziemy mieć z tym coraz większy problem. Niestety uważam, że to dotyczy nie tylko Polski, ale i całego świata. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się dzisiaj, stan polskiej psychiatrii, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi i młodzieżą, jest wręcz tragiczny. Po pierwsze, profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Profilaktyka w szkołach. Musimy w to bardzo mocno włączyć szkoły.

Proszę państwa, chodzi o to, żeby w tych organach znaleźli się ludzie, którzy mają wiedzę (Dzwonek), umiejętności i doświadczenie, bowiem tylko w ten sposób będziemy mogli coś z tym problemem zrobić. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo serdecznie, pani przewodnicząca.

To jest bardzo jasno zapisane w ustawie.

Była również mowa, że oczekujemy, że ustawa o innych zawodach medycznych będzie niezwłocznie procedowana. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień i zostanie ona przekazana do konsultacji. Faktycznie jest to jedna z najistotniejszych ustaw, która dopina system związany z zawodami medycznymi. Część zawodów medycznych ma swoje własne ustawy, z których dwie przegłosowaliśmy w poprzedniej kadencji.

Pytanie brzmiało: Dlaczego muszą przystępować do egzaminu specjalizacyjnego?

W tym zakresie bardzo mocno współpracuje i pracuje PARPA.

Bardzo wiele informacji, bardzo wiele szkoleń w tym zakresie jest procedowanych.

Ale jednocześnie bardzo mocny jest udział, wzrasta udział w szkoleniu profesjonalistów medycznych, lekarzy w tym zakresie.

Oczywiście każdy samorząd jest samodzielny.

Jeśli chodzi o pytanie. Zresztą dwa pytania były na piśmie: pana posła Szopińskiego, a w szczególności pana posła Grzegorza Rusieckiego, który zadał bardzo szerokie pytanie.

To zostanie przygotowane. Oczywiście zgadzam się, tak jak powiedziałem na wstępie, że problem będzie narastał.

Cały czas widzimy, że uzależnienia od nowych technologii internetowych są bardzo mocne.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu psychicznym oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 1631, do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (druki nr 1136, 1317, 1355 i 1548) Proszę pana posła Piotra Babinetza o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Myślę, że zacząć trzeba od tego, że pamięć o Ignacym Łuksiewiczu jako twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego jest bardzo żywa w Polsce. Dowodzą tego choćby różne wnioski o ustanowienie roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Pan Ryszard Rabski wraz z panią dyrektor Barbara Olejarz prowadzi bardzo ważną instytucję kultury - muzeum w Bóbrce w miejscu, gdzie Ignacy Łukasiewicz w 1854 r. otworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej.

Wsparcia tej inicjatywie udzieliła też marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Elżbieta Witek.

Wreszcie marszałek Sejmu skierowała projekty uchwał do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja Kultury i Środków Przekazu zajęła się tymi projektami na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r.

Została wprowadzona istotna poprawka, którą zgłosił pan poseł Marek Rząsa z Platformy Obywatelskiej, również z Podkarpacia.

Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata. Ignacy Łukasiewicz urodził się w Zadusznikach pod Mielcem, w zubożałej rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach. Po śmierci ojca - uczestnika Powstania Kościuszkowskiego, ze względu na sytuację finansową musiał porzucić gimnazjum w Rzeszowie i podjąć pracę jako pomocnik aptekarski. Zdobytą wiedzę i umiejętności rozwinął w trakcie studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wiedniu. Działał we Lwowie, pracując w aptece Piotra Mikolasha, gdzie razem z Janem Zehem w procesie destylacji ropy naftowej wydzielił z niej naftę. Pracował także w Gorlicach, Jaśle i Krośnie. W powiecie krośnieńskim, w Bóbrce, współpracując z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą-Zrenckim, utworzył w 1854 roku pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Z kolei w Ulaszowicach, w Klęczanach, w Polance, a później w Chorkówce uruchomił rafinerię ropy naftowej. Jako twórca przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów i Rumunów. Był też wynalazcą lampy naftowej. W 1853 roku przy świetle skonstruowanej przez niego lampy wykonano pierwszą nocną operację w szpitalu na Łyczakowie we Lwowie. Zmarł w Chorkówce, a pochowany został w Zręcinie koło Krosna. Ignacy Łukasiewicz, wraz ze swoją siostrą Emilią Stacherską, angażował się w działalność niepodległościową, za konspirację w okresie Powstania Krakowskiego był więziony przez Austriaków. Wspierał finansowo Powstanie Styczniowe, a później udzielał schronienia i umożliwiał pracę jego uczestnikom. Był też posłem na Sejm Krajowy i radnym krośnieńskiej rady powiatowej, przewodził Towarzystwu dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa w Galicji. Pełnił wiele funkcji społecznych. Jako wielki filantrop fundował szkoły, szpitale, kościoły, drogi i mosty. Utworzył Towarzystwo Zaliczkowe w Krośnie. Organizował kasy zapomogowe, które jako pierwsze takie instytucje w Europie zabezpieczały robotników na wypadek choroby czy inwalidztwa. Jako pierwszą założył w kopalni Bóbrka kasę bracką, czyli nowoczesny system ubezpieczeń społecznych robotników. Dbał również o rozwój oświaty i kultury oraz edukację pracowników przemysłu naftowego. Za działalność charytatywną papież Pius IX nadał mu tytuł szambelana papieskiego i odznaczył go Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. Jako twórca i organizator przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz doprowadził do rozwoju Podkarpacia, a stopniowo znacznej części polskich ziem pod zaborami, tworząc bardzo wiele miejsc pracy i podnosząc poziom życia mieszkańców. Jego liczni następcy - przemysłowcy naftowi doprowadzili do rozkwitu tej gałęzi polskiej gospodarki. Na zapoczątkowanym przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. Także dzisiaj jest patronem przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego w Polsce, a Jego dziedzictwo powinno być mocno i stale rozwijane oraz propagowane w Europie i na świecie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza” Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tutaj już właściwie cały życiorys i dokonania Ignacego Łukasiewicza zostały przedstawione.

Ignacy Łukasiewicz był bardzo zaangażowany w konspirację niepodległościową od początku lat 40. XIX w., szczególnie w Rzeszowie. W okresie powstania krakowskiego działała też jego siostra Emilia Stacherska. Później w trakcie pracy w kopalni w Bóbrce, która powstała w 1854 r., i destylarni, a później w rafinerii w Chorkówce, która powstała w 1865 r., udzielał schronienia powstańcom styczniowym oraz chętnie zatrudniał ich w przemyśle naftowym. Mieli oni wielki wpływ na rozwój techniczny kopalni i rafinerii, a tym samym rozkwit przemysłu naftowego na Podkarpaciu.

Aktywnie pracowali w nim późniejsi oficerowie jak Stefan Torma czy bardzo zasłużeni dla Polski walczący przez kilkadziesiąt lat o niepodległość Marian Ocetkiewicz zamordowany potem przez Niemców w Auschwitz czy Jan Szczurek-Cergowski, który przez chwilę był nawet prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Oni oczywiście wcześniej walczyli też w Legionach Polskich i w wojnie przeciwko bolszewikom.

Odwiedził on wówczas rafinerię nafty w Krośnie, siedzibę „Strzelca” i dom dyrektora Władysława Wachala. Tak to ziarno niepodległościowe zasiane w Krośnieńskiem przez Ignacego Łukasiewicza sprowadziło do Krosna Józefa Piłsudskiego.

Myślę, że rok Ignacego Łukasiewicza przyczyni się do tego, że takie działania będą prowadzone z jeszcze większą intensywnością w przyszłym roku w całej Polsce. Odbędą się również spotkania międzynarodowe z udziałem Amerykanów, Rumunów i Kanadyjczyków, tych, którzy później na wzór Ignacego Łukasiewicza rozwijali przemysł naftowy. Prawo i Sprawiedliwość z radością popiera uchwałę o uchwaleniu roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Bardzo proszę, pan poseł Marek Rząsa, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Swoje wystąpienie w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza zacznę trochę nietypowo, bo od zadania pytania: Co łączy leki i wyroby farmaceutyczne, zabawki, telewizory, komputery, kleje i farby, włókna i tworzywa sztuczne, materiały wybuchowe, mosty, drogi, kosmetyki, opony, środki transportu od morskiego poprzez drogowy, skończywszy na lotnictwie? Każdy z tych otaczających nas przedmiotów istnieje dzięki surowcowi, który jest fundamentem współczesnej cywilizacji, techniki i gospodarki mającym podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej, a przede wszystkim będącym jednym z najważniejszych surowców energetycznych. Jest także ważnym czynnikiem kształtującym międzynarodowe stosunki gospodarcze, społeczne i polityczne, czego byliśmy w historii świata niejednokrotnie świadkami, choćby w momencie kryzysów energetycznych i paliwowych. Tym globalnym i ponadczasowym surowcem jest oczywiście ropa naftowa. A z jaką osobą kojarzy się ta ciekła kopalina? Naturalnie i oczywiście z naszym wybitnym rodakiem, mieszkańcem Galicji i Podkarpacia Ignacem Łukasiewiczem, pionierem światowego przemysłu naftowego, odkrywcą procesów przeróbki ropy naftowej, wreszcie konstruktorem pierwszej w świecie lampy naftowej. Był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego. Farmaceuta, chemik, przedsiębiorca, filantrop to najczęściej wymieniane zawody i rodzaje jego działalności zawodowej i społecznej. Praca, odkrycia naukowe, wynalazki, konstrukcje nie przysłoniły mu jednak najważniejszej sprawy dla ówczesnych Polaków - walki o niepodległość i wolność ojczyzny.

Był prekursorem szeregu rozwiązań socjalno-bytowych, m.in. ubezpieczeń społecznych robotników czy tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych. Był fundatorem nowych szkół, szpitali, kościołów. Uważał edukację dzieci i dorosłych za dziejową konieczność.

Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Lewica z wielką satysfakcją i dumą zagłosuje za ustanowieniem roku 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza. Żył, realizując swoje pasje, ale nie zapominał o dobru innych, przede wszystkim uboższych. W procesie destylacji ropy naftowej wydzielił naftę. Skonstruował pierwszą lampę naftową, która zrewolucjonizowała ówczesny świat i bardzo pomogła ludziom w ich codziennym życiu.

Wyprzedził swoją epokę także w działalności społecznej. Organizował m.in. kasy zapomogowe, które jako pierwsze tego typu instytucje w Europie zabezpieczały robotników na wypadek choroby lub inwalidztwa. Dbał o oświatę, inicjował budowę szpitali, sadzenie drzew owocowych. O Ignacym Łukasiewiczu powinno być głośno. Naszym obowiązkiem jest propagowanie czynów i osiągnięć tego człowieka.

W ten sposób chcą oddać hołd temu wielkiemu człowiekowi, patriocie, społecznikowi i jednemu z najwybitniejszych polskich naukowców. Mamy nadzieję, że to odznaczenie zostanie przyznane. Proszę, pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po otrzymaniu uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza napisałem projekt uchwały, aby rok 2022 był rokiem Ignacego Łukasiewicza. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie z kolegami i koleżankami posłami możemy z dumą powiedzieć, że przyszły rok będzie rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Oprócz tego był patriotą, pomagał ludziom, to wielka rzecz.

Tych szkół jest wiele.

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo!

Opowiadalibyście różne straszne rzeczy i żadne szyby naftowe nie wyrosłyby w tym pionierskim zagłębiu.

Aptekarstwo. Mój Boże, przy współczesnym, jak to nazywacie, uregulowaniu tej branży Ignacy Łukasiewicz w ogóle nawet nie miałby szansy terminować w jakiejkolwiek aptece w Łańcucie czy w Rzeszowie, ponieważ wasze regulacje zamykają także i ten fach. Młodzi przedsiębiorcy, rzutcy, łebscy ludzie muszą szukać pracy na obczyźnie zamiast w ojczyźnie. Świeć, Panie, nad jego duszą. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Był przecież aptekarzem, a w nafcie początkowo widział lek. Bardzo jestem dumny, że nazwisko Łukasiewicza przetrwało w nazwie i w koncepcji polskiej sieci naukowo-badawczej. Szczerze mówiąc, miałem pewne wątpliwości, kiedy ogłaszano ten projekt, ale nie ze względu na postać wybitnego Polaka, ale ze względu na nasilenie znaków diakrytycznych występujących w tej nazwie. Poprzemy ten projekt uchwały. Jest dobry. Ten wielki Polak naprawdę zasługuje na najwyższy rodzaj upamiętnienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zapisać się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Wysoka Izbo!

Znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Dopiero w wieku 30 lat obronił dyplom. Ten aspekt jego życia jest bardzo ważny. Chciałbym, żebyśmy my jako posłowie opowiadali o nim, bo jest to przykład człowieka, który sam, powiedziałbym, ze zubożałego ziemiaństwa, dzisiaj powiedzielibyśmy: gdzieś z rodzin o niskich dochodach, potrafił się wybić na przepiękną postać, patriotę, wybitnego naukowca i człowieka, który stworzył cały przemysł nafciarski w Polsce. Dziękuję.

Pani Marszałek! Ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza staje się faktem. Pragniemy w ten sposób oddać hołd wielkiemu patriocie i społecznikowi, jednemu z najwybitniejszych polskich naukowców, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju przemysłu naftowego. Projekt był poprzedzony ogromnym zainteresowaniem Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środowisk naukowych. Zarząd województwa podkarpackiego powołał komitet honorowy obchodów i zaplanował wiele przedsięwzięć, by godnie uczcić 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza. Jest jeszcze jedna inicjatywa marszałka województwa podkarpackiego, prezydenta miasta Rzeszowa, rektora Politechniki Rzeszowskiej, by odznaczyć Ignacego Łukasiewicza pośmiertnie Orderem Orła Białego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. List intencyjny w tej sprawie (Dzwonek) przekazuję na ręce pani marszałek i proszę o wsparcie tego działania. Przy wsparciu Prezydium Sejmu uda się w porozumieniu z prezydentem RP postulat samorządowców spełnić. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Inicjatywa ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza jest godna uznania, bo jest on patronem przemysłu naftowego i rafineryjnego w Polsce, a jego dziedzictwo powinno być propagowane w Europie i na świecie. Ten rok można wykorzystać do różnych działań edukacyjnych. W Bydgoszczy np. znakomicie funkcjonuje Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym zwracam się z tego miejsca z gorącym apelem do pana ministra Czarnka o opracowanie w roku 2022 programu na rok Łukasiewicza dla szkół noszących jego imię, programu, który będzie obejmował integrację tych szkół, środki na konkursy, rozgrywki sportowe, dotacje na sprzęt badawczy i wyposażenie pracowni chemicznych, wycieczki do polskich rafinerii i wycieczki szlakami Ignacego Łukasiewicza. Szanowny panie ministrze, gdyby pan zapomniał, to ja w tej sprawie wystosuję do pana interpelację. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Wysoka Izbo! Oczywiście dla wielu miast, dla wielu miejscowości i regionów w Polsce nazwisko Łukasiewicz jest niezwykle ważne, wiąże się m.in. z tym, że tam, gdzie powstał przemysł nafciarski, był on szansą na dynamiczny rozwój tych regionów. Tak jest także w naszym rejonie, w Czechowicach-Dziedzicach. Świadectwem tego jest również jedna ze szkół, która nosi imię Łukasiewicza, jest on patronem tej szkoły. W związku z tym mam pytanie do rządu i bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie. Jestem pewien, że ten rok będzie takim momentem, w którym zarówno historia, jak i dokonania Łukasiewicza będą stanowiły o pewnych, powiedziałbym, imprezach, będą stanowiły ważny element tego roku. Czy będą środki finansowe przewidziane w budżecie na realizację takich zadań? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jako osoba zajmująca się pomocą społeczną z radością przyjęłam inicjatywę uczczenia pamięci Ignacego Łukasiewicza. Ignacy Łukasiewicz w świadomości społecznej zapisał się jako ojciec Ignacy. Na wsiach organizował kasy gminne udzielające chłopom bezprocentowych, krótkoterminowych pożyczek spłacanych w cotygodniowych drobnych ratach. Pożyczał pieniądze chłopom wożącym ropę z kopalni do rafinerii na zakup i utrzymanie koni i wozów. Udzielał pomocy finansowej chłopskim synom podejmującym studia. Odstępował drzewo z lasu na budowę domów. Leczył chłopów za darmo. W kopalni w Bóbrce utworzył kasę bracką, prototyp dzisiejszego ZUS-u, 3-procentowy potrącony podatek od zarobków zabezpieczał bezpłatne leczenie, lekarstwa i było 20 centów dziennego chorobowego dla robotnika. Jak napisał jego kolega ze studiów, Anczyc: Nikt nie wie, ile i komu Łukasiewicz dobrodziejstw świadczył i do kawałka chleba dopomógł, bo czynił to jak najciszej i nieraz dobry uczynek przez siebie spełniony innym przypisywał. I właśnie takie informacje powinny się znaleźć w programach szkolnych. Bardzo dziękuję. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Jest pan poseł? Wysoka Izbo! Prometeusz na ludzką miarę” to tytuł biografii Ignacego Łukasiewicza, która jest najlepszym podsumowaniem tego pięknego życiorysu wielkiego, wybitnego Polaka, twórcy przemysłu naftowego, a przede wszystkim polskiego patrioty. Sam w 2016 r. zainicjowałem jako wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wielki program społeczny, edukacyjny, którego szósta edycja odbywa się w tym roku pod auspicjami PGNiG, „Być jak Ignacy” Ten program jest znakomitą podstawą naukową, aby wszystkie samorządy, wszystkie szkoły, które chcą w 2022 r. uczcić pamięć i promować dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza, uczyniły to. W mojej ocenie kopalnia Bóbrka powinna być obowiązkowym punktem na mapie wycieczek szkolnych wszystkich uczniów z całej Polski.

Dziękuję bardzo.

Miało być pytanie, jest sprostowanie, bo tutaj czcigodna koleżanka zagalopowała się w swojej laudacji śp. Ignacego Łukasiewicza i wyliczywszy jego piękne dzieła filantropii, niewymuszonej, bez terroru państwowego socjalu. Wy tego nienawidzicie.

Zgroza, abominacja, nic podobnego. Przynależność do kasy brackiej nie była wymuszona. Przynależność do kasy brackiej nie była ukrytą formą wyzysku fiskalnego.

Proszę zatem jednego z drugim nie porównywać. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad tym projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań.

Proszę pana posła Piotra Babinetza o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W zasadzie można powiedzieć, że był głównie mojego autorstwa, natomiast bardzo serdecznie dziękuję panu prof. Krzysztofowi Dybciakowi za cenne uwagi, które pozwoliły uzupełnić ten projekt. Pani marszałek skierowała go do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wprowadzono drobne, stylistyczne poprawki.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza. Dzieciństwo i młodość spędził na Wileńszczyźnie. Od stycznia 1919 roku, czyli już jako siedemnastoletni ochotnik, walczył przeciwko bolszewikom w Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a później na własną prośbę - w 13. pułku ułanów, dowodzonym przez majorów - braci Jerzego i Władysława Dąmbrowskich. W tym czasie zetknął się z rosyjskimi i białoruskimi sojusznikami w oddziałach generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. W 13. pułku walczył aż do zwycięstwa nad bolszewikami. Po wojnie odbył studia przyrodnicze na uniwersytetach w Warszawie i Wilnie. Rozpoczął współpracę z wileńskim pismem 'Słowo', redagowanym przez swojego starszego brata - Stanisława Cat-Mackiewicza, i dał się poznać jako patriota wielonarodowego i wielowyznaniowego dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W latach 30. ukazały się jego pierwsze utwory literackie: nowele, sztuka teatralna, powieść kryminalna oraz tom reportaży pt. 'Bunt rojstów' Po wybuchu II wojny światowej, gdy Wilno zajęli Litwini, przez kilka miesięcy wydawał polski dziennik 'Gazeta Codzienna' W Wilnie przetrwał okupację sowiecką, a po tym, kiedy to miasto trafiło pod okupację niemiecką - odmówił wydawania kolaboracyjnego pisma w języku polskim. Gdy zamieścił w 'Gońcu Codziennym' kilka antybolszewickich tekstów, został oskarżony o współpracę z Niemcami. Od wyroku skazującego uratowali go kierownik Biura Informacji i Propagandy Okręgu AK Wilno Zygmunt Andruszkiewicz oraz wybitny pisarz i żołnierz Sergiusz Piasecki. Po wojnie został oczyszczony z zarzutu kolaboracji. W maju 1943 roku, za zgodą polskich władz podziemnych, był świadkiem prowadzonej przez Niemców ekshumacji ciał oficerów zamordowanych przez Sowietów w Katyniu. W 1944 roku Józef Mackiewicz, wraz z żoną Barbarą Toporską, uciekł do Warszawy, a następnie do Krakowa, gdzie napisał broszurę pt. 'Optymizm nie zastąpi nam Polski' Następnie małżonkowie przedostali się do Rzymu. Tam powstał reportaż 'Ponary-Baza' - wstrząsający opis ludobójstwa dokonanego przez Niemców na Żydach oraz raport pt. 'Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów' ze wstępem generała Władysława Andersa. Józef Mackiewicz publikował też artykuły w pismach: 'Wiadomości', 'Kultura', 'Wilno i Lwów' oraz w rosyjskiej, litewskiej, ukraińskiej i białoruskiej prasie emigracyjnej. W 1947 roku przeniósł się do Londynu, gdzie wydano pierwszą napisaną przez niego po angielsku książkę o sowieckim ludobójstwie na Polakach pt. 'The Katyn Wood Murders' W 1952 roku zeznawał przed komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych do zbadania zbrodni katyńskiej. W 1955 roku Mackiewiczowie przenieśli się ostatecznie do Monachium, gdzie mieszkali do końca życia. W kolejnych latach powstawały jego najważniejsze dzieła literackie oraz kolejne teksty publicystyczne, niektóre napisane wspólnie z Barbarą Toporską. Były to przede wszystkim powieści: 'Droga donikąd', 'Karierowicz', 'Kontra', 'Sprawa pułkownika Miasojedowa', 'Lewa wolna', a także zbiory esejów i publicystyki: 'Zwycięstwo prowokacji', 'Ściągaczki z szuflady Pana Boga', 'Nie trzeba głośno mówić', 'W cieniu krzyża', 'Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy', 'Droga Pani...', 'Fakty, przyroda i ludzie' W warstwie faktograficznej, o którą Mackiewicz szczególnie dbał, przedstawiał życie mieszkańców pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego na tle przełomowych wydarzeń historycznych i odwoływał się do tradycji wielonarodowej I Rzeczypospolitej. Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu, poszukiwał wszystkiego, co mogłoby łączyć mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w tym antybolszewicką opozycję w Rosji, na drodze ku wolności narodów. Od strony artystycznej były to teksty łączące fakty z fikcją literacką, zawierające znakomite opisy przyrody i mistrzowskie przedstawienie psychologicznych motywów działania bohaterów powieści. Stworzył oryginalny model powieści fabularno-dokumentalnej epicko przedstawiający obraz rzeczywistości. W wielu reportażach pisarz ukazywał bezpowrotnie utracone Kresy Wschodnie wielkiej Rzeczypospolitej. Jego życiowe motto stanowiły słowa: 'Tylko prawda jest ciekawa' Oboje zostali pochowani w Londynie. W PRL twórczość Mackiewicza była zakazana i niemal niedostępna. Jej poznanie stało się możliwe dzięki rozwojowi wydawnictw drugiego obiegu. Od 2002 roku przyznawana jest Nagroda Literacka imienia Józefa Mackiewicza. Jego twórczość cieszy się wielkim uznaniem krytyków i badaczy literatury. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w stulecie urodzin wybitnego pisarza - uznając wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi, oraz uniwersalne wartości jego prozy literackiej - ustanawia rok 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza” Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. I znowu pan poseł Piotr Babinetz, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Rzeczywiście transmisja, wywiad telewizyjny zakłóca nam. Ale teraz dajmy panu posłowi prawo. Dziękuję bardzo.

Chodzi o fragment „Drogi donikąd”, właściwie wstępu. Drugą częścią tej dylogii było „Nie trzeba głośno mówić”

Oto ten wstęp. Poza powieściowymi osobami wszystko jest autentyczne w tej relacji. Ludzie, zwierzęta i rzeczy; zdarzenia, tajne dokumenty i daty; nazwy wsi; świt i zachód o czasie moskiewskim, linia przebiegająca rojstami, która dzieliła litewską i białoruską republiki sowieckie, a także kierunek każdej drogi. Autentyczne są nazwiska oficerów ludowego komisariatu bezpieczeństwa państwowego NKGB. Autentycznym nazwiskiem jest również: Wiśniewski. Znałem go bardzo mało, prawie przelotnie, a imienia nie wymienię. Gdy przed laty, w tamtym okresie, opracowywałem pierwsze szkice do niniejszej powieści, on, Wiśniewski, pożyczył mi maszynę do pisania. Powiedziałem wtedy: 'Panie Wiśniewski, jeżeli kiedykolwiek wydam tę książkę, podziękuję panu na jej wstępie' On tylko odkiwnął głową z niedowierzaniem, powiedziałbym nawet, że z tego rodzaju lekceważeniem, jakie się w ciężkich opresjach życia posiada dla projektów pozornie nierealnych. Nie wiem, czy i gdzie żyje w tej chwili Wiśniewski: w litewskiej, białoruskiej czy w polskiej republice sowieckiej? Autor” Rzeczywiście wyjątkowa była ta dbałość Józefa Mackiewicza o szacunek dla dobrych ludzi, ale też o dokładność, precyzję i fakty, wszak zresztą mówił przecież: „Tylko prawda jest ciekawa” Był Józef Mackiewicz konsekwentnym wrogiem bolszewizmu i komunizmu, ale i każdego totalitaryzmu. Zarazem był chyba największym mistrzem słowa wśród największych polskich pisarzy - prozaików i publicystów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Józef Mackiewicz bezsprzecznie nie jest najbardziej znanym polskim pisarzem, i szkoda.

Moje pokolenie w ogóle nie miało szansy poznać jego powieści, ponieważ, wiadomo, nie uznawał Mackiewicz PRL-u jako legalnej formy państwowości polskiej. Był tu zresztą zwalczany ze wszystkich sił.

Jeśli państwo pozwolicie, posłużę się tutaj cytatem z prof. Włodzimierza Boleckiego, który tak oto charakteryzuje i postać, i twórczość: „Myślenie Mackiewicza nie było związane z żadną doktryną i jest całkowicie antyideologiczne (jedyną ideologią jest w niej antykomunizm) Dlatego też jest nieporozumieniem wpisywanie myśli Mackiewicza w terminy współczesnego życia politycznego. Szczególnym nonsensem jest dziś czynienie z pisarza patrona polskiej prawicy. Ci, którzy tak robią, zdają się zapominać, że Mackiewicz był najbardziej zaciekłym przeciwnikiem polskiej myśli narodowej (...), a jego. stosunek do Kościoła, polityki Watykanu, czy mniejszości narodowych zbliżał go zdecydowanie do postawy, można powiedzieć, nawet liberalnej - w najbardziej potocznym znaczeniu tego słowa. Dewizą pisarza były po prostu słowa: 'żyj i daj żyć innym' Doceniając wielkość prozy Mackiewicza i nietuzinkowość także jego myśli publicystycznej, politycznej, sądzę, że wart jest, aby się znaleźć nawet w kanonie literatury, lektury szkolnej. To naprawdę jest znakomita proza i to naprawdę Mackiewicz udowadnia, czemu służy literatura i jakie są zobowiązania pisarza. Klub Koalicji Obywatelskiej (Dzwonek) oczywiście popiera ten projekt i ten wniosek, aby to był Rok Józefa Mackiewicza. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Józef Mackiewicz - pisarz, dziennikarz, publicysta, ale także furman i drwal. Jeśli życie potrafi być skomplikowane, a nasze wybory trudne, to właśnie życie Mackiewicza takie było.

Oskarżono go więc o kolaborację, a AK wydało nawet wyrok śmierci. Mackiewicz wierzył, że jego zadaniem jest przekazywanie wiedzy o świecie, ale miał odwagę swoją twórczością burzyć mity i legendy, naruszać stereotypy zbiorowej wyobraźni historycznej. Głównym tematem jego twórczości był rozpad wielonarodowej wspólnoty na terenach byłego Księstwa Litewskiego, za który winił nacjonalizm oraz ekstremistyczną politykę bolszewików i hitlerowców. Głównym bohaterem jego twórczości był zawsze pojedynczy człowiek zaplątany w wiry wydarzeń i ideologii. Cała twórczość Mackiewicza jest oskarżeniem XX-wiecznej polityki o deformowanie i niszczenie życia jednostek i narodów. Jego utwory wywoływały gorące polemiki. Był oskarżany o naruszanie politycznego i narodowego tabu, czyli np. o podważanie legendy Piłsudskiego, kwestionowanie polityki AK czy rzekome pomniejszanie martyrologii Polaków podczas II wojny światowej. Pisarz uważał antykomunizm za swój światopogląd, ale równie krytyczny był wobec nacjonalizmu. Uważał, że nacjonalizm jest źródłem największych nieszczęść Europy i Polski. Twierdził, że błędem II Rzeczypospolitej były mocarstwowe rojenia, które prowadziły do konfliktów z narodami zamieszkującymi wschodnie obszary kraju, a błędem było traktowanie ich jako obywateli drugiej kategorii. Był zwolennikiem różnorodności, wielojęzyczności i wielokulturowości. Podkreślał: natura nie zna ani rasizmu, ani nacjonalizmu. Ma więc polska prawica czego się uczyć od Mackiewicza. W publicystyce powojennej odróżniał naród niemiecki od hitleryzmu i analogicznie rozróżniał naród rosyjski i system komunistyczny. Pisał, że obwinianie wszystkich Niemców za hitleryzm jest takim samym absurdem, jak obwinianie wszystkich Rosjan za komunizm czy zbrodnie katyńskie. Jako pierwszy potępił niszczenie przez aliantów niemieckich miast w końcowej fazie wojny. Jako szczecinianka znająca piękno niemieckiego Sztetina tylko z fotografii podpisuję się pod tymi słowami. Jeśli osobiście (Dzwonek) mogę za coś cenić Mackiewicza, to za jego odwagę. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki, wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać” Od tak mądrych i trafnych słów wybitnego pisarza Józefa Mackiewicza chciałbym rozpocząć tę dzisiejszą wypowiedź. Tak jak ponadczasowa jest ta sentencja, podobnie niezapomniany powinien być jej autor. Już jako gimnazjalista walczący ochotniczo w wojnie polsko-bolszewickiej, w późniejszych latach piszący liczne felietony i reportaże dotyczące politycznej sytuacji w państwie i na świecie, był wzorem zaangażowanego i aktywnego obywatela.

Przez całe swoje życie miał przeciw sobie wszystkie najważniejsze centra opiniotwórcze polskiego życia publicznego. W roku 1942 został on nawet skazany na karę śmierci, jednak na szczęście odpowiednio szybko został uniewinniony. I mimo tych wydarzeń nie zniechęcił się jednak do działania. Przez to uważam, że powinien być on wzorem dla wszystkich, również współczesnych ludzi. Mackiewicz nie bał się poruszać tematów tabu oraz wyrażać głośno i klarownie własnej opinii. Takiej postawy mogliby się uczyć od niego niejedni, którym brak odwagi do działania i przeciwstawienia się temu, co według nas złe, w obawie, że może być to kontrowersyjne. Dużo miejsca w swojej literaturze powyższy autor poświęcił także prawdzie, mówiąc, że jedynie ona jest ciekawa. Jeszcze wiele biograficznych przywołań mogłoby pokazać, że postać Józefa Mackiewicza jest inspirująca i powinna zostać pokazana tym, którzy nie mieli okazji o nim usłyszeć, oraz przypomniana tym, którym niestety udało się o niej zapomnieć. Szukajmy wzorców dla naszych dzieci w ludziach z wiarą we własne przekonania i odwagą, by je wyrażać. Pokazujmy im na przykładzie tego właśnie pisarza, że działanie nie zawsze jest proste, że czasami warto jest przyjmować trudności na takiej drodze, aby żyć w zgodzie z samym sobą. Zróbmy to wszystko poprzez ten dzisiejszy projekt.

Czytajcie go, państwo, którzy tutaj recytujecie te lekcje „wytnij - wklej” z Wikipedii.

Tak jak za PRL-u surowo przestrzegał przed przyzwalaniem na publikację jego książek w formie, być może, ocenzurowanej, selektywnej w kraju, tak też czczenie jego pamięci przez ten ciągle jeszcze na poły post-PRL-owski Sejm, Sejm Rzeczypospolitej trzeciej i pół, mógłby uznać wręcz za zniewagę. Lubicie powtarzać wybrane frazy: Jedynie prawda jest ciekawa. Przypomnijcie, że mówił także: Ignorancja mas rośnie wraz z upowszechnieniem czytelnictwa. Mimo wszystko moment jest dość wzruszający i przełomowy, jeśli dochodzi do procedowania nad tą uchwałą w atmosferze, jak widzę, koncyliacyjnej, ogólnej niekontrowersyjności tej postaci, chociaż gdyby, powtarzam, była wam lepiej znana jego twórczość, pewnie chcielibyście go wyświęcić z tej sali i z życia publicznego Rzeczypospolitej, tak jak chciał to uczynić Adam Michnik, w swoim czasie nominując Mackiewicza na zoologicznego antykomunistę. Jednak jest jakiś postęp w przyrodzie. Dzięki temu, że tu, w Sejmie, to nazwisko i imię pada, jeszcze parę osób o nim usłyszy.

Gdyby koledzy i koleżanki z klubu Lewicy mieli tę lekturę w odpowiednim momencie na nocnym stoliku, to może w ogóle nie przystąpiliby do tych formacji, które dziedziczą tradycje formacji rabusiów i zbrodniarzy. Cześć pamięci Józefa Mackiewicza!

Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza. Szanowni Państwo!

Pisarz, dziennikarz, publicysta polityczny, zagorzały antykomunista, laureat emigracyjnych nagród za twórczość literacką, nominowany do Literackiej Nagrody Nobla. Wiarygodność i rzetelne przedstawienie prawdy wbrew panującym w tamtym czasie politycznym uwarunkowaniom nie zniechęciły go do przedstawiania rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Pisał często na złość całemu światu, publikował felietony, artykuły i reportaże, w których opierał się przede wszystkim na relacjach naocznych świadków, w tym także swoich własnych. Już jako dziecko uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w obronie Warszawy w 1920 r., co niewątpliwie wpłynęło na ukształtowanie jego osobowości. Z jednej strony pesymistyczny poeta, historyk, publicysta, a z drugiej - zagorzały polityk. W jego twórczości zaznaczały się dwa nurty - interesował go człowiek jako jednostka oraz dzieje mas. Jego powieści odznaczają się precyzją konstrukcji, szczegółowością, żywością języka i świetnym osadzeniem w realiach geograficznych.

Uczestnicząc w ekshumacji w Katyniu, opracował białą księgę o morderstwie katyńskim, niezbity dowód zbrodni popełnionej przeciwko narodowi polskiemu. Czesław Miłosz napisał o dwóch jego tekstach: dopóki będzie istnieć polskie piśmiennictwo, te dwa zapisy grozy XX w. powinny być stale przypominane. Mackiewicz piętnował zacieranie prawdy. Nie bał się głośno krytykować postępowania, zachowania, które mogłoby tuszować fakty historyczne. Zacytuję jego wypowiedź: „Skoncentrowane kłamstwo ludzkie posiada siłę, której granic na razie nie znamy”

Koło Parlamentarne Polska 2050 będzie głosowało za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Bardzo proszę, pierwsze pytanie pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Józef Mackiewicz to pisarz potrafiący w bardzo dosadnych słowach przekazywać swoje myśli, człowiek, którego dorobek został uhonorowany ufundowaniem specjalnej nagrody jego imienia, o czym mowa była w uzasadnieniu. Ale trzeba też jasno powiedzieć, że w kapitule przyznającej owo wyróżnienie zasiada człowiek wydalony dość niedawno z jednego z największych krajów Europy ze względu na głoszone wartości, które nie są akceptowane przez demokratyczne społeczności. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Pani Marszałek! Ja już wiele powiedziałem na temat samego przyszłego patrona, natomiast mam pytanie do rządu i proszę o odpowiedź na piśmie: Jakie działania rząd podejmie w związku z ustanowieniem tego patrona 2022 r. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Komunizm był największym wrogiem Józefa Mackiewicza.

I to, że dzisiaj Lewicy i Platformie Obywatelskiej przeszkadza to, że w kapitule Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza zasiada Rafał Ziemkiewicz, któremu odbierane są prawa obywatelskie i który nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, tylko i wyłącznie wystawia wam świadectwo.

Dziękuję, panie pośle. Tak, trafne spostrzeżenie, słuszna uwaga.

Jeśli lewica z lewej i lewica z prawej jednogłośnie czczą pamięć Józefa Mackiewicza, to wygląda na to, że wszystko już straciło tu znaczenie, słowa się zdewaluowały. Opinie, które tutaj są formułowane, mogą w dowolny sposób być oderwane od rzeczywistości, jaką pozostają właśnie np. biografie zasiadających w Wysokiej Izbie posłów.

Dziękuję. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam przerwę do godz. 15.45.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę państwa posłów o zajmowanie miejsc. Informuję, że Senat przyjął bez poprawek następujące ustawy: o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, o zmianie ustawy o sporcie. W związku z tym planowane punkty 22. i 23. porządku dziennego stały się bezprzedmiotowe. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, - o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1714, 1715, 1713 i 1709. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu. Proszę się uspokoić, to będzie słychać. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 1716. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozparzenie tego wniosku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 1689. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 1678, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 1548. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 1548, zechce nacisnąć przycisk. Po uchwałach, proszę państwa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 1600. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 1600, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 441 - za, 1 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Są wnioski formalne. Proszę. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o odroczenie obrad do 3 listopada, do godz. 10, celem umożliwienia rządowi Rzeczypospolitej przedłożenia ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną. Dzisiaj, szanowni państwo, jeżeli to posiedzenie Sejmu nie uchwali tej ustawy, to polscy podatnicy za wasz upór zapłacą do następnego posiedzenia blisko 100 mln zł. 100 mln zł to jest kara nałożona przez Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę i premiera Morawieckiego na polskich podatników. Tak, drodzy państwo. To pan, panie prezesie, wycofuje się podobno z Izby Dyscyplinarnej, ale czy jest pan tak słaby i tak bardzo boi się, że nie ma wystarczających głosów, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną? Pomożemy panu, zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną i odblokujemy środki dla Polski, które dzisiaj wasz rząd blokuje.

Pani Marszałek! Szanowni państwo. Państwo mają zwolnienia lekarskie, proszę pana. Jest głos przeciw do wniosku formalnego. Proszę doczytać regulamin, panie pośle. Proszę doczytać regulamin, panie pośle, jak wygląda wniosek formalny i głos przeciw do niego. Szanowni Państwo! To jest moment, w którym rzeczywiście ważą się losy przyszłości Polski i przyszłości Unii Europejskiej. Tej Unii Europejskiej, w której niedługo rozpęta się burza we wszystkich państwach z powodu kosztów energetycznych, z powodów kosztów życia, jakie. ideologiczna Komisja Europejska narzuca. I to jest właśnie ten fundamentalny moment, w którym państwo polskie musi powiedzieć jasno: niepodległość nie na sprzedaż. stanowienia prawa w Polsce i instytucji jest nie na sprzedaż. od rządu polskiego w tym momencie. Dziękuję, panie pośle. Ponieważ padł wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Proszę. Szczęść Boże. Dzisiaj na wokandę wjeżdża projekt: stop segregacji sanitarnej. Przyjmijcie go wy, wszyscy, którzy nie jesteście zwolennikami dyskryminacji własnych rodaków. Od ubiegłego tygodnia wiedzę z urzędu o istnieniu ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych o bezprawności nakazu zamaskowania posłów na Sejm RP posiada pani marszałek. Pod rozwagę i materiał do przemyślenia dla Stirlitza. Już po pogrzebie, ale komu nie wrosły w serce jego sceny, jego filmy. Wachmistrz Soroka, major Hubal oraz inni - bardzo często - funkcjonariusze. Teraz, panie pośle. Panie pośle, po pierwsze, to, co pan przedstawił, nie jest opinią BAS-u, tylko opinią zewnętrzną. Po drugie, 27 października wojewódzki sąd administracyjny na skargę, jaką pan złożył na mnie za to, że kazałam panu opuścić salę posiedzeń za nienoszenie maseczki. Pańska skarga została przez sąd wojewódzki odrzucona. Sąd uznał, że marszałek Sejmu ma prawo wydawać zarządzenia, w tym to zarządzenie o obowiązku noszenia maseczek. Dziękuję, panie pośle. Laryngolog, panie pośle, się kłania. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica, z wnioskiem formalnym. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rozmawiamy o wielu kwestiach, ale nie o podstawowej, dlatego składamy wniosek formalny o przerwę i wprowadzenie do porządku obrad informacji ministrów i premiera o programie drożyzna+. Inflacja w Polsce sięga 7% w październiku. Podstawowe produkty drożeją. Nierozmawianie o tym, że drożyzna+ wpędzi Polaków w święta, które będą najbiedniejsze od 6 lat. To jest wasza odpowiedzialność. Wstydzicie się tego, że w waszych miastach, powiatach musicie się tłumaczyć z drożyzny. Ale ona jest faktem. Premier i minister powinni dzisiaj powiedzieć, dlaczego rząd nie reaguje. Nie wystarczy powiedzieć: nie będziemy zmniejszali akcyzy. Ponieważ został zgłoszony wniosek formalny o przerwę w obradach, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Pani Marszałek! Koledzy i Koleżanki Posłowie! Polska 2050, panie pośle. Koleżanki i Koledzy! Bardzo się cieszę z waszego aplauzu i z mojej decyzji. To bardzo dobrze świadczy o możliwościach dalszej współpracy z wami. Bardzo się cieszę. Zatem w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 chciałem złożyć wniosek o zmianę sposobu prowadzenia obrad. Otóż, panie prezesie. Polska to wielka odpowiedzialność. Panie pośle, marszałek Sejmu prowadzi obrady. Rozumiem, że pan do mnie to kieruje. Chciałem. Dzisiaj.

Panie pośle. Panie pośle. Panie pośle Zalewski, czy pan słyszy, co ja do pana mówię? Panie pośle Zalewski, panie pośle Zalewski, panie pośle, proszę się odwrócić do mnie twarzą. Teraz pan słyszy? Stamtąd nic nie słychać, co marszałek mówi? Nie prowadzimy w tej chwili żadnej debaty. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość.

Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi Terleckiemu, że na szczęście zakończył tę tęczową wystawkę pana Czarzastego. Już kilkudziesięciu posłów podpisało się pod wnioskiem o odwołanie pana marszałka, który wczoraj urządził seans nienawiści przeciwko 140 tys. obywateli.

Gdzie pan był? To, co pan wczoraj zrobił, to jest hańba dla tej Izby. To nie był wniosek formalny. Ale nie było, panie pośle, żadnego wniosku formalnego, więc nie ma wniosku przeciwnego. Nie, nie ma wniosku. Przepraszam, pan nie był wywoływany. Nie było wniosku, panie pośle. Była wypowiedź pana posła. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1622. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1622, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Działa, już teraz działa. Kto jest przeciw?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1683. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1683, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1684. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1684, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju. Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przystępujemy do trzeciego czytania projektu uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 1661. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 1661, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1607, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1710 i 1713)

Przepraszam, były zgłoszone trzy poprawki Senatu i komisja wnioskuje o odrzucenie tych poprawek.

W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Wszystkie poprawki zgłoszone zostały do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1711 i 1714) Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła uchwałę Senatu z 28 października tego roku z druku nr 1711 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Uchwała wprowadziła do projektu 10 poprawek. Po dyskusji i głosowaniu cztery poprawki komisja przyjęła, pozostałe poprawki komisja odrzuciła.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Poprawki od 1. do 7. zgłoszone zostały do ustawy o podatku od towarów i usług. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 8. i 10., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1712 i 1715) Proszę pana posła Andrzeja Kosztowniaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedłożenia sprawozdania Komisji Finansów Publicznych z druku nr 1715 o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1712.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 2. i 54., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 7. poprawce Senat proponuje m.in. skreślić art. 66. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 16. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 20. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 22. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za nie był nikt, 439 - przeciw, wstrzymało się 4. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 24. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 28. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosowało 441 posłów.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 29. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 30. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 32. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 40. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 42. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W 46. poprawce Senat proponuje m.in. nie nadawać nowego brzmienia pkt 11 w art. 4 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 46. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 47. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 48. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 49. poprawce do art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 49. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 53. poprawce Senat proponuje dodać zdanie drugie w art. 50 ustawy nowelizującej. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 53. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 58. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 59. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 61. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (druki nr 1687 i 1709) Proszę pana posła Michała Jacha o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie i Panowie Premierzy! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, druk nr 1687. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 27 października 2021 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Z poprawką tą łączy się poprawka 5. Głosujemy. Kto jest przeciw? Już działa. Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 - za, przeciw - 443, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 7. poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie art. 8. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1646-A. Proszę pana posła Jarosława Sachajkę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Panie pośle.

Wysoka Izbo! Na dzisiejszym posiedzeniu komisji rozpatrzyliśmy poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Uprzejmie proszę o poparcie tego projektu. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1646. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 4. i 5., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1646, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1680-A. Proszę pana posła Jerzego Polaczka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury rekomenduje, aby Wysoki Sejm przyjął załączony projekt ustawy.

Pierwszy to wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, a drugi to poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi, również z pijanymi kierowcami. Koszt społeczny wszystkich wypadków i kolizji drogowych w Polsce rocznie to ponad 55 600 mln zł. Myślę, że Wysoki Sejm poprzez przyjęcie tej regulacji znacznie ograniczy bardzo dotkliwe i liczone w setkach tysięcy gorzkie skutki wypadków, liczbę osób rannych, tych, którzy ponieśli śmierć.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 440 posłów. Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 7. poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie art. 12 ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1680, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1666-A. Proszę pana posła Piotra Króla o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1633. Sejm na 40. posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1666 do Komisji Infrastruktury oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1666. Komisje przedstawiają również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Wszystkie poprawki zgłoszono do art. 1 zawierającego zmiany do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 3. poprawce do art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy nowelizowanej wnioskodawcy proponują, aby dodać lit. Głosujemy. Kto z pań i z panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu z druku nr 1666, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1679-A. Proszę panią poseł Bożenę Borys-Szopę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1675. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu w dniu 29 października 12 poprawek wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie dziewięciu i odrzuceniu pozostałych oraz o uchwalenie ustawy. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 9. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Poprawka 9. stała się bezprzedmiotowa. Poprawki od 10. do 11. zgłoszone zostały do art. 2 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1679 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 431 - za, 10 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1678-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Leszka Dobrzyńskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Komisja rozpatrzyła ww. projekt i opiniuje przyjęcie go w całości. Jednocześnie opiniujemy odrzucenie wszystkich poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1678.

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 9. poprawce do art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioskodawcy proponują zmiany w ust. 1. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1705-A. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła pięć wniosków mniejszości i dwie poprawki do rządowego projektu ustawy o podatku akcyzowym. Wszystkie wnioski mniejszości komisja odrzuciła. Przy głosowaniu nad poprawkami poprawka nr 1 została przez komisję przyjęta, a poprawka nr 2 została odrzucona. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tego bardzo ważnego projektu ustawy. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Wszystkie wnioski mniejszości oraz poprawka 1. zgłoszone zostały do ustawy o podatku akcyzowym. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 1. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1707-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę panią poseł Iwonę Arent o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Sejm na 40. posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1707 do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawki zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja rozpatrzyła zarówno wniosek, który mówił o odrzuceniu projektu w całości, jak i poprawkę dotyczącą innego modelu ustalania rynkowej ceny energii elektrycznej. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1707. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawkę. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1707, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Przypominam, że uprawnione podmioty złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego: - Koło Poselskie Konfederacja o punkty: - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Stop segregacji sanitarnej, - Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie przymuszania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w eksperymencie medycznym zwanym szczepieniami przeciwko COVID-19 i praktykowanej bezprawnej, niekonstytucyjnej, nieregulaminowej dyskryminacji niezaszczepionych; - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) o punkt: - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu negocjacji z Republiką Czeską w kontekście postępowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego Turów; - Koło Poselskie Polska 2050 o punkt: - Informacja Prezesa Rady Ministrów o skali nepotyzmu w spółkach skarbu państwa; - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody w systemie ochrony zdrowia, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, - Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, - Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, druk nr 918, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, druk nr 646, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, druk nr 582, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, druk nr 580, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 436, Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk nr 1226, Sprawozdanie komisji o senackim projekcie ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, druki nr 1019 i 1217. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań.

Ponieważ są to wnioski tożsame i zgłoszone zostały przez ten sam podmiot, Sejm nad tymi wnioskami będzie głosował łącznie. Przystępujemy do głosowania nad tożsamymi wnioskami w sprawie uzupełnienia porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie projektu ustawy Stop segregacji sanitarnej zgłoszonymi przez Koło Poselskie Konfederacja. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tych wniosków, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji Ministra Obrony Narodowej w sprawie przymuszania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w eksperymencie medycznym zwanym szczepieniami przeciwko COVID-19 i praktykowanej bezprawnej, niekonstytucyjnej, nieregulaminowej dyskryminacji niezaszczepionych. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu negocjacji z Republiką Czeską w kontekście postępowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji Prezesa Rady Ministrów o skali nepotyzmu w spółkach skarbu państwa. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody w systemie ochrony zdrowia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, druk nr 918. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 919. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, druk nr 646. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, druk nr 580. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 436. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk nr 1226. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym sprawozdania komisji o senackim projekcie ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, druki nr 1019 i 1217. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1716)

Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy głosowania i wyczerpaliśmy porządek dzienny 40. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Zamykam listę posłów zgłoszonych do oświadczeń. Ogłaszam przed oświadczeniami 2 minuty przerwy porządkowej.

Wznawiam posiedzenie. Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Lorka. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę przez szacunek dla występującego pana posła wyciszyć rozmowy, ewentualnie przenieść je poza salę sejmową. Jan Stanisław Jankowski wielki zapomniany. Wczoraj w jednym z moich wystąpień opowiedziałem historię jednej z najstarszych polskich szkół, piotrkowskiej Sorbony, czyli dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Wydana jakiś czas temu przez długoletniego dyrektora tej szacownej placówki Zenona Bartczaka monografia obejmująca spis jej słynnych absolwentów zawierała jedno ze znanych nazwisk. Był to Stanisław Jankowski. Jan Stanisław Jankowski urodził się w Krasowie Wielkim w maju 1882 r. Po ich ukończeniu pracował jako asystent w Katedrze Chemii Rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wczesnej młodości był zaangażowany patriotycznie, działał w podziemiu w różnych organizacjach niepodległościowych. Był aktywny na niwie związków narodowych, służył także w Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Był członkiem Centralnego Komitetu Narodowego. Po odzyskaniu niepodległości rzucił się w wir pracy politycznej. Był współzałożycielem Narodowej Partii Robotniczej, ministrem pracy w rządzie Witosa w 1921 r. Zamach majowy nie zakończył jego kariery. Nadal aktywnie wspierał umiarkowane organizacje o narodowej proweniencji. Po wybuchu wojny i wykształceniu się struktur Polskiego Państwa Podziemnego w 1941 r. został dyrektorem Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu RP na Kraj, pod koniec 1942 r. został zastępcą delegata rządu na kraj, a w kwietniu 1943 r. samym delegatem. W 1944 r. został mianowany wicepremierem i kierował Krajową Radą Ministrów. Zatwierdził zgodę na wybuch powstania warszawskiego, tak tłumacząc swoją decyzję: „My tu nie mamy wyboru. Walki w mieście wybuchną, czy my tego chcemy, czy nie. Za dzień, dwa lub trzy Warszawa będzie na pierwszej linii frontu Trudno sobie wyobrazić, że nasza (...) młodzież, którą myśmy szkolili od lat (...) daliśmy jej broń do ręki, będzie się biernie przyglądała albo da się Niemcom bez oporu wywieźć do Rzeszy? Jeżeli my nie damy sygnału do walki, ubiegną nas w tym komuniści.

Razem z innymi przywódcami państwa podziemnego został przewieziony do Moskwy i bezprawnie osądzony w sfingowanym procesie. Został skazany na 8 lat. Na 2 tygodnie przed końcem wyroku wycieńczony został najprawdopodobniej zamordowany we Włodzimierzu nad Klaźmą. Symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach. Bardzo dziękuję za wygłoszone oświadczenie.

Szczęść Boże. Wysoka Pustawa Izbo! Panie Marszałku!

Mam okazję spojrzeć w oczy paru posłom, którzy reprezentują tutaj demodyktaturę większości parlamentarnej i stanowią, o, w niektórych przypadkach nawet prominentne postaci grupy aktualnie trzymającej władzę. Odrzuciliście zatem właśnie nasz projekt „Stop segregacji sanitarnej” Tego projektu nie musielibyśmy składać, gdyby prawo w Rzeczypospolitej obowiązywało, gdyby rodził się pewien automatyzm prawny. Bezprawie jest diagnozowane, ścigane, wykrywane i podlega penalizacji. Zło jest naprawiane, przestępcy są hamowani w swoich zapędach. Wasze zapędy - wasze, większości parlamentarna, i tu muszę przenieść spojrzenie na drugą stronę Izby, bo to jest przecież zjednoczona koalicja COVID-owa - do tego, żeby segregować, a przez segregację dyskryminować własnych rodaków, są, jak widać, nieokiełznane. Przymuszanie do udziału w eksperymentalnych procedurach medycznych, a w niektórych przypadkach pseudomedycznych, bo np. wtykanie ludziom patyka w różne otwory ciała pod pretekstem zwalczania chorób zakaźnych jest w tej chwili praktyką rozpowszechnioną i wymusza się to, korzystając z relacji podległości, i na żołnierzach, i na artystach, i na policjantach, i na ludziach innych służb mundurowych, cywilnych, administracji państwowej. Przymus zamaskowania wielokrotnie zdemaskowany jako procedura znachorska, a jednak medyczna. Znachorska, ponieważ szereg badań wykazuje nieskuteczność, niecelowość, a niektóre studia wykazują również szkodliwość tej procedury. Najmniej szkodliwa z tego wszystkiego autointoksykacja, niedotlenienie, które niewątpliwie tutaj daje się we znaki. To jest być może najmniej drastyczny z tych elementów całego tego teatru absurdów, który tutaj zbudowaliście.

Jedna nadeszła, jak to się mówi, z miasta, a druga nadeszła z Biura Analiz Sejmowych.

Wczoraj niejako z ostrożności procesowej złożyłem oświadczenie poselskie na piśmie, ale ponieważ ono się nie uwidoczniło jeszcze w protokole tego posiedzenia, w związku z tym ponownie zwracam uwagę Wysokiej Izby i Prezydium Sejmu na istnienie tych ekspertyz. Te ekspertyzy, szanowni państwo, w sposób dla mnie samego zadziwiający, bez ezopowej prawniczej mowy, bez niuansowania i dzielenia włosa na czworo, te ekspertyzy profesorów Chmaja i Grabowskiej jednoznacznie diagnozują stosowanie przymusu zamaskowania (Dzwonek) posłów na Sejm Rzeczypospolitej jako bezprawne, a kary, represje, nie mówiąc o nękaniu i mobbingu, z tego wynikające traktują również jako bezprawne, bezpodstawne.

Proszę o zakończenie oświadczenia i proszę nie robić tu żadnych wystawek. Jak będę chciał, to sobie sięgnę. Polecam lekturę. Pan poseł Lisicki. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Miała ona za zadanie zreformować samorząd warszawski i połączyć Warszawę w jeden organizm, ponieważ wcześniej Warszawę tworzyło kilkanaście gmin. Obecnie Warszawa składa się z 18 dzielnic, które mają swoje władze, statuty i skromne kompetencje. W Warszawie cały czas mamy do czynienia z centralizacją. Prezydent Warszawy, który aktualnie nie ma za bardzo czasu na zarządzanie największym miastem w Polsce, ma jednocześnie olbrzymie kompetencje. Dzielnice, a szczególnie rady dzielnic, które są jednostkami pomocniczymi, a które są jednocześnie blisko mieszkańców, nie mają w zasadzie żadnych kompetencji uchwałodawczych pozwalających na stanowienie prawa, ponieważ ich uchwały może zawiesić prezydent i anulować rada Warszawy. Rada dzielnicy może wybrać co prawda zarząd, ale duża część kompetencji, np. kompetencje kadrowe, jest w gestii prezydenta. Prezydent może udzielić tych kompetencji burmistrzowi dzielnicy, ale może ich także nie dać, co w Warszawie dotyczy tych burmistrzów, którzy nie podobają się władzom Warszawy. Odbija się to na ważnych sprawach, bo np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są uchwalane w radzie Warszawy, a w dzielnicy są tylko opiniowane. Stąd też duże opóźnienia w uchwalaniu miejscowych planów w Warszawie. Obecnie jedynie 40% obszaru miasta jest objęte miejscowymi planami. Jednocześnie w każdej dzielnicy jest urząd oraz jednostki budżetowe. Radnych dzielnic jest około 400 - to bardzo duży koszt dla budżetu miasta. Rady dzielnic oraz urzędy dzielnic to znaczny koszt dla budżetu miasta, ale jednocześnie, a może przede wszystkim, to znaczne niewykorzystane możliwości.

Zwłaszcza że obecny włodarz stolicy ma czas zwiedzać miasta na całym świecie, ale nie ma czasu odwiedzić swojego miejsca pracy. Proszę o wygłoszenie oświadczenia panią poseł Teresę Hałas. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Listopad to miesiąc, w którym Polska odzyskała niepodległość. To miesiąc zadumy i pamięci, miesiąc wszystkich świętych i wszystkich zmarłych.

Każdy, kto choć raz stanął na cmentarzu Orląt Lwowskich, ten poczuł i zrozumiał wiele, jeśli nie więcej niż wiele. To właśnie te białe krzyże mówią wszystko o bohaterach walczącego Lwowa. Mieli po kilkanaście lat, a czasem nawet i mniej, kiedy dla potrzeb obrony sami wybierali nocne warty i służby w okopach. Ich hasło: nie damy Lwowa wydawało się szaleństwem, bo przecież to one, dzieci, miały zmierzyć się z zaprawionymi w bojach ukraińskimi żołnierzami, świetnie uzbrojonymi i doświadczonymi. Byli uczniami w szkolnych mundurkach, studentami czy słynnymi lwowskimi batiarami, dziećmi ulicy, które od najmłodszych lat zarabiały na chleb.

I tak po kolei: Jurek Bitschan, czternastolatek, symbol wszystkich Orląt, tych znanych z nazwiska i tych bezimiennych, który wychodząc z domu, zostawił taki list: Kochany tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest, gdy wojska brakuje do oswobodzenia Lwowa, iść. Z moich zadań w domu zrobiłem już tyle, ile trzeba. Walczył w pierwszym szeregu, kiedy został trafiony dwiema kulami na cmentarzu Łyczakowskim. Tadzio Jabłoński, czternastolatek. On też uciekł z domu, by dołączyć do obrońców Lwowa. Bił się jak bohater, szedł zawsze w pierwszym szeregu, by jak najszybciej zobaczyć mamę, która została w zajętej przez Ukraińców części miasta. Nie spotkał jej już nigdy. Walczył na Górze Stracenia, a potem poszedł za swoim dowódcą bronić Persenkówki. Tam został ciężko ranny i zmarł po 3 tygodniach cierpień w szpitalu. To on rozmawiał ze swoją mamą, mówiąc: Ja biłem się tak samo jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Helenka Grabska poległa ze swoim bratem Jankiem, Janeczka Prus zginęła, ratując rannego żołnierza. I wiele innych, pięknych, z warkoczykami i sercem na dłoni. Jako jedyne miasto w Polsce został odznaczony orderem Virtuti Militari za niespotykane męstwo i dzielność lwowskich dzieci. Niech to świadectwo dzisiaj, w chwilach pamięci i zadumy listopadowego święta, napełni wielu z nas dumą z wielkiego czynu Orląt Lwowskich. Niech będzie ono pięknym i docenionym przykładem szlachetnego serca dla ich dzisiejszych kolegów, rówieśników, młodych mieszkańców wolnej Polski. Może niejeden odłoży na chwilę smartfona i przeniesie swoją myśl do czasów trudnych, znaczonych wojną, walką i oddaniem w sprawie najwyższej wagi - narodowej godności i wolności. Głęboko w to wierzę, bo wierzę w młode, piękne, wrażliwe, otwarte i dobre serca. Wieczna chwała bohaterom! Pokój tobie, Polsko! Bardzo dziękujemy za tak wzruszające oświadczenie.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Tak się składa, że w ostatnich dniach wielu z was w rozmowie ze mną cytuje pewną rymowankę: od morza aż do Tatr rządzi dzisiaj Polski Ład. Wobec powyższego chciałbym na samym początku podziękować kolegom i koleżankom parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości w osobach prezesa okręgu Marka Asta, pana wojewody Władysława Dajczaka, pani europosłanki Elżbiety Rafalskiej, pani poseł Elżbiety Płonki, posła Jurka Materny, że razem, wspólnie, w soczystym dialogu gospodarskim, rozważaliśmy listę rekomendacyjną dla Polskiego Ładu i owocem tej debaty wspólnotowej wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości było to, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której 677 mln trafiło na ziemię lubuską. Każdy z nas, taka jest natura parlamentarzysty, stroi się w piórka sprawcy tego wydarzenia, ale to przecież jest działanie zespołowe. I za tę pracę zespołową każdej z was i każdemu z was, koledzy i koleżanki posłowie i posłanki, dziękuję. Oczywiście warto powiedzieć o spektakularności programu Polski Ład, który na ziemi lubuskiej odnotowany jest m.in. takimi propozycjami wsparcia finansowego jak to, co się wydarzyło w powiecie krośnieńskim.

Dobra. Pięćdziesiąt parę tysięcy mieszkańców tego powiatu dzisiaj może się radować, że nie będą musieli ani do Gorzowa, ani do Zielonej Góry się tarabanić, po prostu u siebie, w swoim szpitalu, będą mogli się diagnozować. W ramach tych pieniędzy jest 46 mln na powiat krośnieński, gdzie np. jedna z gmin, gmina Maszewo, absolutnie nie rządzona przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, dostaje 7600 tys. i załatwia tym samym wszystkie swoje potrzeby w zakresie inwestycji drogowych. Po prostu tak jest. Następna rzecz, słuchajcie, tutaj mam dużą satysfakcję, bo lubię takie klimaty.

Sprawa niebywale ważnej rangi. To znaczy, że kultura wysokiej jakości będzie również mogła w dobrej rzeczywistości infrastrukturalnej realizować się w gminie Otyń.

Z panem wójtem po wielokroć rozmawialiśmy o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest budowa centrum kultury górali bukowińskich. Przecież wiecie doskonale, że Lubuszanie to przybysze z wielu regionów Polski. Tego typu podział, nie tylko na drogi, nie tylko na kanalizację, na kwestie sanitarne, ale na szkoły, na ośrodki kultury, na potrzeby wyższego rzędu, to jest piękny wachlarz oferty Polskiego Ładu dla ziemi lubuskiej i całej Polski. To są dobre nowiny. Oświadczenie teraz wygłosi pani poseł Anna Ewa Cicholska. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu pana premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami w Nidzicy. Ktoś może powiedzieć: rządowa propaganda. Otóż nie. Po spotkaniu w Nidzicy zaprosiłam samorządowców z powiatów mławskiego i ciechanowskiego, starostów, burmistrzów i wójtów różnych opcji politycznych. Samorządowcy wyrażali uznanie dla działań rządu, a Program Inwestycji Strategicznych pozwoli im na realizację wielu potrzebnych inwestycji. Polska lokalna nie potrzebuje polityki, potrzebuje zrównoważonego rozwoju, potrzebuje środków finansowych. Polski Ład i zawarte w nim programy dają jej szansę na nowe drogi, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków, odnawialne źródła energii, nowoczesną sieć ciepłowniczą, rozbudowę infrastruktury sportowej, kulturalnej, oświatowej. Nie sposób wszystkiego wymienić. Warto pamiętać jednak, że przekazane środki finansowe to pobudzenie aktywności inwestycyjnej samorządów, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy i poprawa warunków życia obywateli. Proszę o zabranie głosu pana posła Czesława Siekierskiego. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Chcę wyrazić wielką troskę, jeśli chodzi o sytuację w rolnictwie. Oto plony na skutek warunków pogodowych na wielu polach nie zostały zebrane w znacznej części. To dotyczy wielu gmin, że wspomnę tylko gminy z mojego okręgu, myślę tu o gminach Pacanów, Nowy Korczyn. Zostały poniesione koszty, nie ma, nie będzie dochodów. Sytuacja wygląda tak, że rolnicy będą mieli problemy z zapewnieniem pasz dla zwierząt. A więc resort rolnictwa powinien podjąć działania, aby tych rolników wspomóc specjalnymi programami.

To wszystko powoduje taką sytuację, że poziom dochodów z tytułu sprzedaży nie zapewni, nie da możliwości pokrycia kosztów produkcji, kosztów odtworzenia tej produkcji, kosztów jej utrzymania. I oto do takiej trudnej sytuacji dochodzą wyjątkowo trudne problemy wynikające z sytuacji na rynku paliw, gazu, energii. Mamy taki skutek, że nawozy zdrożały w ciągu ostatniego okresu dwu-, trzykrotnie. A więc jeśli przeanalizujemy tę trudną sytuację, o której mówiłem wcześniej, to zobaczymy, że rolnicy nie będą mieli za co kupić środków produkcji potrzebnych do realizacji kolejnego cyklu produkcyjnego. To wejdzie oczywiście do przyszłych kosztów produkcji, bo te koszty będą znacznie wyższe. Rolnicy nie będą mogli wyłożyć takich środków i takich nakładów, które by zapewniły odpowiedni poziom produkcji. A chodzi o to, żeby rolnictwo było konkurencyjne na rynku. To musi doprowadzić także do zmniejszenia produkcji, ale także wzrostu cen na produkty rolne, a w konsekwencji wpłynie na ceny artykułów spożywczych, za które zapłaci konsument, w tym także rolnik, mieszkańcy wsi, my wszyscy jako konsumenci.

Oczywiście to zużycie będzie się zmniejszało na skutek galopującego wzrostu cen. Do tego dokłada się rosnąca inflacja.

Rolnicy, panie ministrze, oczekują (Dzwonek) na pana działania, aby poprawić ich sytuację. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia pana posła Waldemara Andzela. Panie Marszałku! Z tego miejsca chciałbym skierować podziękowanie na ręce prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego za pierwszą edycję rządowego funduszu Programu Inwestycji Strategicznych. Zgadzam się ze słowami pana premiera, iż jest to program bezprecedensowy i wyjątkowy, dzięki któremu do polskich samorządów trafią 23 mld zł. Jest to element Polskiego Ładu, który konsekwentnie jest wprowadzany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Do województwa śląskiego, z którego pochodzę, trafi ponad 2 mld zł. Program Inwestycji Strategicznych daje szansę na rozwój i polepszenie warunków życia absolutnie w każdej gminie w kraju. Inwestycje te to rozwój infrastruktury drogowej, tak potrzebnej zwłaszcza na terenach wiejskich, to budowa i rozbudowa obiektów kulturalno-oświatowych, poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej i wiele wiele innych. Wyrażam głęboką nadzieję, że przed polskimi samorządami kolejne edycje tego niezwykle ważnego programu. Dziękuję bardzo. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Maciej Kopiec. Nie ma, zatem. Oj, przepraszam bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję zapoznać się z zaleceniami Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród Studentów i Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, które mówią m.in. o tym, że studenci swoim strojem nie powinni naruszać zasad obyczajowości oraz wzorców kulturowych. Oraz że wygląd i strój studentów i studentek mają wpływ na kształtowanie się relacji z pacjentami i nauczycielami akademickimi obu płci. Wytyczne te mówią m.in., że unikanie noszenia bluzek z głębokim dekoltem i spódnic krótszych niż do połowy uda, unikanie wysokich obcasów czy prośba o zakrywanie tatuaży to cudowne sposoby na rozwiązywanie wszelkich problemów. Te zalecenia to wyjątkowo nieodpowiedzialna reakcja na wydarzenia, które miały miejsce na uczelni w roku 2020, kiedy to spłynęły oskarżenia o molestowanie, mobbing oraz gnębienie uczących się na terenie tej uczelni osób przez wykładowców. Sytuacja ta, łącznie z coraz częściej spływającymi informacjami ze szkół z całej Polski o ograniczeniach dotyczących ubioru, to również pokłosie wypowiedzianych przez ministra Czarnka słów o cnotach niewieścich oraz chęć przypodobania się władzy centralnej przez poszczególne placówki naukowo-dydaktyczne. Jeden z doradców premiera mówił: kluczowe jest rozwijanie cnoty i położenie nacisku na właściwe wychowanie kobiet. To skandal. Dyskryminacyjne, szowinistyczne bzdury zaczynają mieć istotny wpływ na sytuację na uczelniach, które powinny być centrum nauki i wiedzy, a nie ideologii, szowinizmu i patriarchatu. Tymczasem treść wydanego zalecenia sugeruje, że odpowiedzialność za wydarzenia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z ubiegłego roku ponoszą studentki i studenci. Edukacja, wolność, poszanowanie dla różnorodności - to podstawy dobrze funkcjonującego demokratycznego państwa. Tylko odpowiednia rzetelna edukacja i odpowiedzialni ludzie pełniący funkcje publiczne są w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Nie jest ono zależne od tego, w co się ubieramy, jak wysokie mamy obcasy, jakiego koloru założyliśmy koszulę i jakie tatuaże mamy. To nic innego jak indywidualna ekspresja i styl bycia. Jeśli ktokolwiek czuje się sprowokowany do czynu zabronionego jakimkolwiek elementem tej ekspresji, problemu powinien poszukać w sobie. Czas najwyższy, aby szkoły postawiły na rzetelną edukację seksualną i antydyskryminacyjną, a nie na ograniczanie młodych, poszukujących swojej tożsamości ludzi, którzy zasługują na dostęp do jak najlepszej wiedzy i możliwość bycia sobą w każdej sytuacji życiowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia pana posła Piotra Adamowicza. Dziękuję, panie marszałku. Panie i Panowie! Ale na razie do rzeczy.

Apel dotyczy zatrzymania destrukcji polskiego systemu edukacji. Ponieważ on jest skierowany do parlamentarzystów, pozwalam sobie go przedstawić. Planowane zmiany w ustawie - Prawo oświatowe są wyrazem bezkompromisowego dążenia do dominacji władzy centralnej. Doprowadziłyby do ograniczenia możliwości współpracy placówek oświatowych z partnerami społecznymi do organizacji koncesjonowanych przez kuratorium oświaty. W konsekwencji skutkowałyby kształtowaniem programu edukacyjnego wyłącznie w oparciu o ideologię przyjętą przez partię rządzącą. Procedowane zmiany ściśle podporządkowują szkoły kuratorium oświaty, czyli terenowemu organowi administracji rządowej. Kuratoria będące obecnie organami nadzoru pedagogicznego nad szkołami staną się organami decydującymi w kwestiach tak ważnych jak wybór dyrektora szkoły, pozaprogramowa oferta edukacyjna, tworzenie sieci szkół itd. Dyrektorom będą groziły sankcje karne, w tym pozbawienie wolności, niewspółmierne do niedookreślonego w doktrynie prawnej przekroczenia uprawnień. Edukacja nie jest polityczna, szkoła nie jest polityczna. Polska oświata jest miejscem wzrastania i tworzenia się polskiego społeczeństwa, którego przyszłość jest uzależniona od doświadczenia, jakie dzisiejsi uczennice i uczniowie, a także pracownicy szkół wynoszą i będą z niej wynosić. Wszelkie zmiany w oświacie przynoszą efekty długofalowe. Błędy rzutują na całe pokolenia, a ich naprawa, o ile możliwa, trwa latami. Chcemy, aby Polska była krajem wolnym, demokratycznym, praworządnym i konkurencyjnym pod względem ekonomicznym, naukowym i społecznym. Tego samego oczekujemy od polskich szkół i przedszkoli. Potężny chaos wywołany deformą oświaty w 2017 r. znacznie pogorszył warunki edukacyjne dzieci i młodzieży, a zignorowanie strajku nauczycieli 2 lata temu pozostawiło to środowisko w stanie zniechęcenia. Pandemia wywołała w szkolnych społecznościach głęboką traumę i frustrację. Naszą wspólną pilną odpowiedzialnością jest wsparcie społeczności szkolnych. W obliczu obecnych wyzwań musimy skoncentrować się na tworzeniu dobrych warunków pracy w atmosferze zaufania i wsparcia dla kadry nauczycielskiej, budowaniu wśród uczennic i uczniów kompetencji uczenia się i rozumienia skomplikowanych procesów zachodzących we współczesnym świecie, współpracy na rzecz rozwiązywania problemów w miejsce zideologizowanych programów nauczania. Szkoła i przedszkola muszą wychodzić naprzeciw wyzwaniom przyszłości, fascynować wiedzą, uczyć krytycznego myślenia, empatii i umiejętności dbania o siebie i dobro wspólne. Wobec powyższego, mając na względzie dobro uczennic, uczniów, kadry nauczycielskiej, społeczności szkolnych oraz całego społeczeństwa, Rada Miasta Gdańska apeluje do prezesa Rady Ministrów, posłów na Sejm oraz senatorów RP o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zatrzymania destrukcji polskiego systemu edukacji. Zostało mi jeszcze 60 sekund, postaram się je wyczerpać.

Bo być może mniejsze miasta zyskają. Jest tam wszystko dokładnie przez gminy wyliczone. Dobrego wieczoru. Bardzo dziękuję panu posłowi. Jako samorządowiec mogę powiedzieć tylko, że w dużej mierze zgadzam się z opinią pana posła co do tego szczęścia, które spotkało miasta, szczęścia w cudzysłowie. Proszę bardzo, pani poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. Wysoka Izbo! Przyznam, że ja dzisiaj pierwszy raz wygłaszam oświadczenie poselskie, a właściwie sytuacja zmusiła mnie do tego, ponieważ wczoraj nie mogłam zabrać głosu, bo ograniczono prawa posłów, ograniczono możliwość zadawania pytań podczas pierwszego czytania projektu: stop LGBT. Bardzo mnie to zasmuciło i dlatego chciałam dzisiaj parę słów powiedzieć na ten temat. To przede wszystkim trudne słowa, które wczoraj usłyszałam, smutne słowa. Przytoczę je państwu, bo to słowa, które wygłosiła osoba reprezentująca wnioskodawców.

Nie zamierzamy przepraszać za sformułowanie: ideologia LGBT, bo to rzekomo ludzie, a nie ideologia. Za każdą ideologią stoją ludzie, tak jak stali np. za ideologią komunistyczną, nazistowską. Przeczytałam państwu te słowa, tak jak już wcześniej powiedziałam, ze smutkiem, bo nigdy takie słowa w naszej Izbie nie padły. Chcę państwu powiedzieć, że wczoraj wieczorem poznałam młodych ludzi - nie tylko młodych - którzy protestowali przed Sejmem. Nazywa się Franciszek Broda. Zapytałam go, dlaczego protestuje przeciwko nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. Powiedział, że to jest projekt, który łamie konstytucję, łamie europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Stwierdził, że nie ma nic przeciwko np. pielgrzymkom na Jasną Górę, z czym zresztą w pełni się zgadzam i absolutnie nie mam nic przeciwko temu. Młody człowiek powiedział, że nie chce wykluczenia postulatów osób LGBT plus z przestrzeni publicznej. Wysoka Izbo!

Nawet nie sugeruje, tylko mówi do nas wprost, że obowiązujące prawo w pełni odpowiada na obawy związane z możliwym naruszeniem reguł dotyczących moralności, obyczajowości, znieważenia symboli państwowych czy przedmiotów kultu religijnego, a projekt wprost godzi w wolność zgromadzeń i dąży do wykluczenia osób LGBT plus. Czy tak powinno się dziać? Czy przyzwoici ludzie powinni to poprzeć? Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia pana posła Fryderyka Kapinosa. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Bez wielkiej determinacji mielczan, m.in. europosła pana Tomasza Poręby, ale również marszałka województwa podkarpackiego pana Władysława Ortyla, oraz bez ich zaangażowania i pracy nie byłoby obecnie właśnie tego, że wspomniana linia kolejowa jest czynna dla przewozów pasażerskich, a 32 km trasy kolejowej z Mielca do Dębicy zostały zmodernizowane, łącznie z przystankami, bezpiecznymi przejazdami oraz infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych. To bardzo ważne, że od 1 września tego roku młodzi ludzie mogą dojeżdżać do szkół podstawowych, zawodowych oraz średnich. Jest również przygotowany dla studentów przejazd z Mielca do Dębicy w niedzielę, który umożliwia im dotarcie do Krakowa czy też do Rzeszowa, a z uwagi na duże zainteresowanie już od stycznia 2022 r. będzie również realizowany tego typu przejazd oraz dodatkowo dedykowany studentom przejazd w piątki po południu. Mielec i powiat mielecki słyną nie tylko z samolotów, nie tylko z piłki nożnej, nie tylko z pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej, ale przede wszystkim z dobrych, uczciwych, pracowitych i przedsiębiorczych mieszkańców, a powrót kolejowych przewozów pasażerskich na linii Mielec - Dębica to dla nich powód do dużej radości i ogromne ułatwienie komunikacyjne. W swoim wystąpieniu skupiam się na moim rodzinnym regionie, jednak nie sposób nie odnaleźć w nim analogii do sytuacji z innych części Polski. Mamy tu bowiem do czynienia z działaniem w znakomity sposób wpisującym się w politykę rządów Prawa i Sprawiedliwości, podczas których odtworzono 400 km linii kolejowych. Mówienie o zwiększaniu dostępności komunikacyjnej w wydaniu czy to kolejowym, czy też autobusowym jest od 6 lat przekuwane w realne działania oraz inwestycje.

W 2018 r. był już rozstrzygnięty przetarg, w 2019 r. zostały rozpoczęte roboty, a dzisiaj możemy się cieszyć właśnie z kursów pociągów pasażerskich na trasie Mielec - Dębica, za co wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, które dało Mielcowi kolejowe okno na świat, na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim, bardzo serdecznie dziękuję. Warto również wspomnieć, że to nie koniec pozytywnych zmian związanych z koleją dla miasta Mielca i powiatu mieleckiego, gdyż trwają działania mające na celu remont linii kolejowej na trasie Mielec - Padew Narodowa, jak również rewitalizację budynku dworca kolejowego w Mielcu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie ma sprawnego działania Policji bez pracowników cywilnych Policji. To duża, prawie 25-tysięczna grupa profesjonalistów: informatyków, finansistów, techników, analityków i innych specjalistów, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie ani Komendy Głównej Policji, ani komend i jednostek Policji żadnego szczebla i żadnej specjalności. Pracownicy cywilni Policji to także niestety kolejna grupa zawodowa, która po 6 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości zderza się z nieuczciwym traktowaniem, drożyzną oraz comiesięczną batalią o związanie końca z końcem. Z danych Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wynika, że aż 6 tys. pracowników cywilnych, czyli aż 1/4, spełniała w 2021 r. warunki do otrzymania wyrównania pensji - uwaga - do wysokości płacy minimalnej. To wstyd, wstyd dla Policji, wstyd dla rządowej instytucji w państwie, w którym - jak twierdzą politycy PiS - mamy pieniądze, nieograniczone zasoby, a premier chwali się comiesięczną wielomiliardową nadwyżką.

Pracownicy cywilni Policji są rozczarowani Policją i mają już dość nieuczciwego traktowania. Dają temu upust w listach i mailach kierowanych zarówno do ministra, jak i do parlamentarzystów. Dlatego ciśnie się na usta pytanie: Jak komendant główny Policji chce osiągnąć taki efekt, by Polacy szanowali Policję, skoro Policja nie szanuje sama siebie? Jak komendant może apelować o szacunek do Policji ze strony obywateli, skoro sam nie szanuje własnych pracowników, o czym świadczą ich paski wynagrodzeń? Jak Policja chce dbać o bezpieczeństwo obywateli, skoro nie dba o bezpieczeństwo finansowe swoich pracowników? Zwracam się również do pana ministra Mariusza Kamińskiego: bez kompetentnych, a jednocześnie właściwie wynagradzanych pracowników cywilnych nie będzie sprawnej Policji, bo inaczej pracę cywili będą musieli wykonywać policjanci. Dlatego apeluję do pana ministra o zmianę polityki ministerstwa i zwiększenie budżetu Policji jeszcze w 2021 r. w celu przyznania pracownikom cywilnym adekwatnych podwyżek.

Był już czarny piątek w wykonaniu pracowników cywilnych Policji, a od minionego czwartku w wielu jednostkach garnizonu łódzkiego nie ma żadnego pracownika cywilnego, gdyż postanowili podreperować swoje zdrowie. W przyszłym tygodniu kolejni pracownicy cywilni w kolejnych garnizonach polskiej Policji zamierzają korzystać ze zwolnień lekarskich. Panie Ministrze! W ubiegłym tygodniu zapowiedział pan program modernizacji służb mundurowych MSWiA.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pracownicy administracji dowiedzieli się (Dzwonek), że do grupy 24 tys. beneficjentów, którzy otrzymają dodatkowe środki budżetowe, należą księża, natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne policjantów komendant główny Policji musi wygospodarować środki sam. Panie ministrze, tym reprezentantom pracowników cywilnych naprawdę było bardzo przykro. Wierzę, że pan spotka się z tymi pracownikami, wierzę, że pan znajdzie rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi Janowi Szopińskiemu, ale, panie pośle, chciałem podziękować także obecnemu na sali posłowi Siekierskiemu, dzięki któremu sens miał zwrot pana posła: Wysoka Izbo. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.